Stwierdzam, że pan poseł Andrzej Szlachta oraz pan poseł Jacek Kurzępa złożyli ślubowanie poselskie. Gratuluję.

Po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów podjęłam decyzję o skreśleniu z porządku dziennego bieżącego posiedzenia punktów: - Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia, druk nr 35, Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, druk nr 37. Na 3. posiedzeniu Sejm nie przeprowadził głosowań nad skierowaniami do komisji obywatelskich projektów ustaw: - o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, druk nr 31, - o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 34. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące te głosowania. Grupa posłów przedłożyła projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, druki nr 158 i 158-A. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący pierwsze czytanie tego projektu ustawy. Proponuję, aby w przypadku druku nr 158-A Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 37 ust. 4 regulaminu Sejmu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Komisja Zdrowia przedłożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, druk nr 110. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.

Stanowiska komisji to odpowiednio druki nr 123 i 124. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 126 i 125. W związku z tym, na podstawie art. 95e regulaminu Sejmu, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Właściwe komisje przedłożyły sprawozdania o projektach ustaw: - o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, - o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Sprawozdania to odpowiednio druki nr 156, 165, 166 i 168. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, podjęłam decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpatrzenie tych sprawozdań. Proponuję, aby w tych przypadkach Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 44 ust. 3. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Prezydium Sejmu proponuje, aby Sejm wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła w dyskusjach nad wszystkimi punktami porządku dziennego. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Informuję, że Konwent Seniorów jednomyślnie zaopiniował propozycję rozpatrzenia na bieżącym posiedzeniu informacji w sprawie programu Mały ZUS Plus, Pakietu Przyjazne Prawo oraz innych ułatwień dla przedsiębiorców, o której przedstawienie wnosił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Punkty porządku dziennego bieżącego posiedzenia będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu i Konwent Seniorów. Informacja w tej sprawie, a także wykaz ustaw, które Senat przyjął bez poprawek, jest dostępna w Systemie Informacyjnym Sejmu. Przed ogłoszeniem komunikatów - wnioski formalne. Pan poseł Marek Rząsa, Koalicja Obywatelska.

Na podstawie art. 184 ust. 1 i 3 pkt 1 regulaminu Sejmu wnoszę o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w celu rozszerzenia porządku obrad o informację prezesa Rady Ministrów w sprawie dramatycznej sytuacji na Podkarpaciu, a sprawa dotyczy Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.

Zagrożone są programy społeczne, inwestycyjne, oświatowe.

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

Informacje o tym, że w wyspecjalizowanej służbie specjalnej, która ma chronić pieniądze podatników, giną pieniądze, że są stamtąd wynoszone pieniądze, to coś, co pokazuje skalę rozkładu państwa pod rządami aktualnej władzy.

Natomiast co słyszymy od ministrów rządu PiS-u? Od rzecznika CBA słyszymy, że wszystko jest w porządku, a od pana ministra Ziobry słyszymy, że trwa postępowanie prokuratorskie. Już czas, aby przeciąć te spekulacje, aby pan premier Morawiecki wyjaśnił, co zdarzyło się w CBA.

Pytanie zada pani. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów z powodu skandalicznej afery GetBacku.

Przez te lata nic nie zrobiono, co więcej, kiedy komisja się tym zajmowała, ludzie, społeczeństwo, obywatele, ci, który doznali szkody w wyniku tej afery, nie zostali wpuszczeni na salę. Co się dzieje?

Tak że bardzo proszę, pani marszałkini, o włączenie tego punktu do porządku obrad. Dziękuję. Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

Bardzo proszę o uczczenie jego pamięci.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek formalny w sprawie zwołania Konwentu Seniorów, przerwy i włączenia do porządku obrad informacji ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie prac nad zwiększeniem świadczeń emerytalnych i rentowych.

Został on odrzucony, pomimo, że przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej wielokrotnie mówili, że te sprawy zostaną uregulowane systemowo.

Proszę zatem o włączenie tego punktu do porządku obrad. Był rządowy projekt ustawy, który przyjęliśmy na poprzednim posiedzeniu Sejmu, dotyczący dodatkowej emerytury i waloryzacji emerytur. Dziękuję bardzo. Proszę posła sekretarza o odczytanie komunikatów. Proszę bardzo, panie pośle. Na podstawie art. 184 regulaminu wnoszę o przerwę w obradach, zwołanie Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku obrad o informację ministra sprawiedliwości i ministra spraw zagranicznych dotyczącą projektu uchwały Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy stwierdzającej rażące naruszenie praworządności w Polsce. W najbliższy wtorek, 28 stycznia, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy odbędzie w Strasburgu debatę dotyczącą funkcjonowania instytucji demokratycznych w Polsce i podejmie odpowiednią uchwałę. W tej uchwale zrówna sytuację w Polsce, sytuację instytucji demokratycznych, z sytuacją w innych niedemokratycznych krajach świata. W związku z tym uważam, że żądanie informacji od ministra spraw zagranicznych i ministra sprawiedliwości jest w tym momencie zasadne, gdyż ta debata, ta uchwała może być kolejnym ciosem w rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim w Rzeczpospolitą Polską. Po pierwsze, wniosek jest nieregulaminowy, a po drugie, panie pośle, rozumiem, że wniosek o sprawdzenie praworządności we Francji też powinien być rozpatrywany, prawda? Jeżeli nie jest. Bardzo proszę. Kłaniam się. Szczęść Boże!

Obywatelski projekt. Ponad 200 tys. podpisów wpłynęło na ręce pani marszałek. Po raz pierwszy od niepamiętnych czasów Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ma szansę zadziałać aktywnie, a nie reaktywnie.

Panie pośle, chciałam poinformować, że wniosek jest, po pierwsze, nieregulaminowy i powinien pan o tym wiedzieć, a po drugie, w tej chwili faktycznie wpłynął wniosek obywatelski i zgodnie z procedurami sprawdzany jest pod względem formalnym w Kancelarii Sejmu. Zgodnie z przepisami w ciągu 3 miesięcy znajdzie swój finał. Nie, panie pośle. Znajdzie swój finał tutaj, w Sejmie. Bardzo proszę, pan poseł Maciej Gdula, Lewica, z wnioskiem formalnym. Wysoka Izbo! Zgłaszam wniosek o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów w sprawie informacji premiera i ministra koordynatora służb specjalnych dotyczącej CBA. To jest niezwykle istotna kwestia, bulwersująca opinię publiczną. Opinia publiczna chce mieć jasną informację, co dzieje się w instytucji powołanej do walki z korupcją. Dziś w instytucji, która jest powołana do walki z korupcją, ma miejsce defraudacja. Tak nie może być, [[Oklaski]] że pojawiają się różne kwoty. Najwyższe kwoty, które się pojawiają, proszę państwa, stanowią 7% budżetu tej instytucji. Nie możemy tego tolerować. Premier i minister powinni nam opowiedzieć, co dzieje się w CBA. Powinniśmy mieć jasność. Powtórzę to raz jeszcze: tą kwestią zajmie się powołana do tego Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Ten wniosek już padł wcześniej, tak że dziękuję panu posłowi. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Proszę o zarządzenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów. Wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego złożenia przez ministra finansów i Komisję Nadzoru Finansowego informacji dotyczącej restrukturyzacji upadłości Podkarpackiego Banku Spółdzielczego. oraz poinformowanie Wysokiej Izby, co to za nowy projekt wprowadzono celem restrukturyzacji tego banku. Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny zastosowały prekursorską, mało znaną metodę restrukturyzacyjną.

Pan chyba nie zwrócił uwagi na to, że powtórzył pan wniosek, który już padł w tej Izbie.

Wysoka Izbo! Chciałbym złożyć wniosek o przerwanie posiedzenia do godz. 11 oraz przygotowanie w tym czasie przez panią marszałek informacji na temat sytuacji związanej z listami poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Mamy bardzo czytelny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przesądził, że listy poparcia mają być jawne. Mamy również wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego, który powiedział, że przepisy RODO nie mają zastosowania, gdy o ujawnienie pewnych dokumentów zwraca się sąd. Wczoraj mieliśmy do czynienia z paniczną decyzją last minute prezesa olsztyńskiego sądu rejonowego Macieja Nawackiego, sędziego we własnej sprawie, który w domu na kartce papieru napisał. zarządzenie prezesa sądu w sprawie odwołania delegacji pana sędziego Pawła Juszczyszyna.

Proszę odróżnić marszałka Sejmu od Kancelarii Sejmu. Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się następujące posiedzenia Komisji: - Finansów Publicznych - godz. 10.30, - do Spraw Energii i Skarbu Państwa - godz. 10.30, - Infrastruktury - godz. 11, - Kultury i Środków Przekazu - godz. 11.30, - Spraw Służb Specjalnych - godz. 12, - do Spraw Petycji - godz. 12, - Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - godz. 12, - Łączności z Polakami za Granicą - godz. 12, - Administracji i Spraw Wewnętrznych - godz. 13, - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 13, - Polityki Senioralnej - godz. 13, - do Spraw Petycji - godz. 13, - Finansów Publicznych - godz. 13.30, - Edukacji, Nauki i Młodzieży - godz. 14, - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 14, - Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - godz. 14, - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 14.30, - Regulaminowej Spraw Poselskich i Immunitetowych - godz. 15, - Finansów Publicznych - godz. 16, - Obrony Narodowej - godz. 16, - Gospodarki i Rozwoju - godz. 16, Zdrowia - godz. 18, Finansów Publicznych - godz. 19.

Dziękuję, pani poseł. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 158 i 158-A) Proszę pana posła Jarosława Krajewskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę tych posłów, którzy nie są zainteresowani tym projektem, o to, żeby prowadzili rozmowy w kuluarach, bo to naprawdę przeszkadza. Bardzo proszę pana posła Jarosława Krajewskiego o przedstawienie uzasadnienia projektu ustawy. Bardzo proszę, panie pośle.

Panie Premierze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. To jest bardzo istotna nowelizacja, którą możemy określić systemowym i komplementarnym usprawnieniem pracy administracji rządowej. Ta nowelizacja, którą przedstawiliśmy Wysokiej Izbie, doprowadzi przede wszystkim do utworzenia dwóch nowych działów administracji rządowej: pierwszego działu - aktywa państwowe i drugiego działu - klimat. Te dwie generalne zmiany, które są zawarte w tym projekcie ustawy, będą również skutkowały zmianami, które będą dokonane w prawie 100 innych ustawach. to szczególnie pokazuje, jak szereg propozycji, które znalazły się w tej nowelizacji, w naszej ocenie jako wnioskodawców przyczyni się do usprawnienia działań administracji i realizacji nowych wyzwań, o których za chwilę powiem. Ponieważ mówimy o administracji rządowej, trzeba przede wszystkim podkreślić, że silne i sprawne państwo to w dużej mierze sprawna i skuteczna administracja rządowa. I w tym kierunku dążymy jako przedstawiciele wnioskodawców - żeby wyjść naprzeciwko tych wyzwań, które się pojawiały i które były zawarte choćby w exposé pana premiera Mateusza Morawieckiego, w programie Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o to, żeby zorganizować pracę administracji rządowej tak, żeby za 4 lata po raz kolejny można było powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymało słowa danego Polakom, że przede wszystkim naszym znakiem rozpoznawczym jest wiarygodność. Ale żeby to zrealizować, musimy dokonać tych zmian. Otóż ten projekt opiera się na trzech filarach i podstawowych celach, które przyświecały wnioskodawcom. Po pierwsze - optymalizacja, po drugie - racjonalizacja, a po trzecie - zwiększenie skuteczności w zarządzaniu.

Ten projekt możemy oczywiście uznać za naturalną zmianę, która wynika również z doświadczenia 4 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale także za dojście do wniosków, które mają z jednej strony wzmocnić zarządzanie aktywami państwowymi, a z drugiej strony przede wszystkim poprawić efektywność prowadzonej polityki klimatycznej, polityki energetycznej i polityki ekologicznej. W kilku szczegółach chciałbym przedstawić Wysokiej Izbie podstawowe informacje dotyczące tych dwóch działów: aktywa państwowe i klimat. Otóż zgodnie z uzasadnieniem, w celu zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania mienia państwowego, co warto podkreślić - zwiększenia jego wartości oraz realizacji najważniejszych celów polityki gospodarczej państwa, proponujemy wyodrębnienie działu aktywa państwowe. Tutaj przede wszystkim chcemy skoncentrować się na zakresie gospodarowania mieniem państwowym, wykonywania praw majątkowych i osobistych, przysługujących Skarbowi Państwa, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa. Chcemy to uzyskać poprzez zwiększenie spójności działań podejmowanych w tych obszarach.

W tym momencie możemy mówić o koncentracji tych uprawnień w zakresie kompetencji ministra aktywów państwowych. Natomiast w celu prowadzenia skutecznej polityki ekologicznej, skutecznej polityki klimatycznej proponujemy wyodrębnienie z działu środowisko nowego działu - klimat. Jest to oczywiście odpowiedź na wzrastające zainteresowanie i nowe wyzwania dotyczące polityki klimatycznej - zarówno w ujęciu krajowym, zwiększającej się percepcji obywateli w zakresie polityki klimatycznej, ale również w zakresie współpracy z Unią Europejską, jak i współpracy międzynarodowej. Warto choćby przypomnieć odbywający się niedawno szczyt klimatyczny w Katowicach, tę deklarację katowicką. Myślę, że Polska tutaj ma bardzo dużo wyzwań, które muszą skutkować również wzmocnieniem działu klimatu. W tym zakresie, o którym mówiłem, nie mieści się też. Dotyka to też kwestii związanych z polityką zagraniczną. Tutaj proponujemy przepisy, które dokonują zmian w zakresie spraw objętych działem członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Jest to doprecyzowanie także niektórych kompetencji ministra kierującego tym działem. O tym jeszcze za chwilę powiem w kilku zdaniach, żeby Wysoka Izba miała pewność co do tego, jaki mamy obrany kierunek jako wnioskodawcy tego projektu. Jeżeli mówimy o. Jeszcze na chwilę wrócę do aktywów państwowych. Otóż dział ten obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, wykonywania praw majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa oraz ochrony interesów Skarbu Państwa z wyjątkiem spraw, które na mocy odrębnych przepisów pozostaną we właściwości innych działów. Minister właściwy do spraw aktywów państwowych będzie reprezentował Skarb Państwa w zakresie gospodarowania mieniem państwowym. Jeśli chodzi o dział klimat, to obejmuje on sprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju. Te projektowane przepisy określają szczegółowy zakres zadań, tych spraw, którymi będzie zajmował się minister klimatu, takich jak: wdrażanie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, gospodarka odpadami, a także efektywność energetyczna oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W ramach proponowanych zmian określamy również zakres spraw należących do działu członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Przenosi się z tego przedmiotowego działu do działu sprawy zagraniczne sprawy dotyczące działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz o polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie. Warto też poinformować Wysoką Izbę, że przykładowo w ramach tych propozycji ze strony wnioskodawców chcemy również zapisać ochronę interesów Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach z instytucjami i organami Unii Europejskiej i wyraźnie wskazać monitorowanie wykonywania wyroków organów sądowych Unii Europejskiej. Jeśli wrócimy jeszcze do kilku kwestii, które są według mnie istotne, jeżeli spojrzymy na zadania w ramach działu aktywa państwowe, to warto przypomnieć, że w tym projekcie znajduje się m.in. rozwiązanie, które obliguje ministra właściwego do spraw aktywów państwowych do tego, żeby być organem właściwym w zakresie wyrażania zgody na zakup lub budowę nieruchomości na potrzeby organów administracji rządowej. Oczywiście jeśli chodzi o projektowane zmiany, te podstawowe, które mają znaczenie dla proponowanej reformy zarządzania aktywami państwowymi, to warto przypomnieć, że ta proponowana nowelizacja zakłada zebranie przedmiotowych kompetencji głównie we właściwości ministra właściwego do spraw aktywów państwowych w porównaniu do stanu obecnego, kiedy to zarówno prezes Rady Ministrów, jak i poszczególni ministrowie odpowiadają za niektóre podmioty Skarbu Państwa. Jeżeli mówimy o tym projekcie, to warto również przypomnieć, że część zmienianych przepisów jest implementacją aktów prawa Unii Europejskiej. W tym zakresie należy wskazać ustawę Prawo energetyczne czy ustawę Prawo ochrony środowiska. Część zmian, tak jak wspomniałem na samym początku, ma charakter redakcyjny związany z wyodrębnieniem dwóch działów aktywa państwowe i klimat. Ale warto również - i myślę, że będziemy nad tym pracować w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych - pracować nad szeregiem rozwiązań merytorycznych, które zmierzają do sprawnej administracji rządowej i do zagwarantowania optymalizacji i racjonalizacji i zwiększenia skuteczności administracji rządowej. Chciałbym również wspomnieć o autopoprawce złożonej do tego projektu, która przewiduje, że pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania będzie sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rodziny. Spieszę od razu z informacją dla Wysokiej Izby, że dzisiaj jest to sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jeżeli mówimy o vacatio legis, bo myślę, że będą również o to pytania, proponujemy, żeby ustawa weszła w życie 7 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem dwóch artykułów, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. To są kwestie związane z nakazem poinformowania w ciągu 7 dni pracowników o zmianach dotyczących ich stosunku pracy. Jeżeli mówimy o vacatio legis, to chciałbym też odnieść się do apelu, który był kierowany ze strony posłów Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej, którzy apelowali do rządu o jak najszybsze przyjęcie ustawy o działach. Mam nadzieję, że posłowie i posłanki opozycji przyczynią się do tego, żeby ta ustawa bez problemów, sprawnie została przeprowadzona w parlamencie, tak żeby można było przystąpić w sposób komplementarny, całościowy do realizacji priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości i rządów Zjednoczonej Prawicy. Na koniec jeszcze raz warto podkreślić, żeby każdy poseł, który będzie głosował nad tą ustawą, nad tym projektem, żeby pamiętał o sprawach fundamentalnych. A tak oceniam kwestię związaną z tym, że naszym celem jako wnioskodawców, a moim jako przedstawiciela wnioskodawców jest to, żeby doprowadzić do optymalizacji, racjonalizacji i zwiększenia efektywności i skuteczności administracji rządowej. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jako pierwszy pan poseł Zdzisław Sipiera, klub Prawo i Sprawiedliwość.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiany dzisiaj w pierwszym czytaniu projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej jest bardzo ważnym dokumentem dotyczącym porządkowania tego, co istotne w administracji, czyli adekwatności do tego, co wynika z potrzeb i tego, co się dzieje wokół nas, jak również potrzeb, które rząd w trakcie swojego zarządzania widzi i w związku z którymi dochodzi do wniosku, że takie zmiany powinny być dokonane.

Aktywa państwowe zbierają z wielu dziedzin i z wielu działów kompetencje. Uwzględniając doświadczenia, które były i do tej pory funkcjonowały, wydaje się, że akurat ten projektowany element jest bardzo istotny i bardzo ważny, dlatego że on porządkuje i sytuuje w jednym miejscu najważniejsze funkcje, które będzie miał minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

W jednym miejscu, w jednym ręku i pod jednym kierownictwem.

Prawa dewizowego, pomoc publiczna dla przedsiębiorców, kontrola i nadzór dotyczące zobowiązań koncesyjnych, zwiększenie liczby członków rady Banku Gospodarstwa Krajowego, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Nabywanie od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego. Zwiększenie udziału nadzoru właścicielskiego poprzez dwóch przedstawicieli w Poczcie Polskiej. Organ likwidujący jednostkę budżetową. To bardzo ważna rzecz, decyzja była w różnych miejscach, w tej chwili będzie w jednym - właśnie w rękach ministra aktywów państwowych. Umarzanie, odraczanie i rozkładanie na raty. Wyrażanie zgody na zakup lub budowę nieruchomości na potrzeby organów administracji rządowej. W jednym miejscu - konkretnie będzie to minister aktywów państwowych. I jeszcze kilka innych kompetencji - bardzo wiele, w jednym miejscu, w dużym skomasowaniu. To bardzo dobre rozwiązanie. Uważamy, że również jest to bardzo ważna rzecz, na ten temat były wielokrotnie dyskusje prowadzone.

W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej pani poseł Gabriela Lenartowicz. Panie Marszałku! Ja w ślad za posłem sprawozdawcą - który notabene zapomniał się podpisać pod tym projektem - apeluję tym razem do pana premiera. Są rzeczy fundamentalne. Jedną ze spraw fundamentalnych jest dobre zarządzanie państwem i kierowanie najważniejszym organem wykonawczym, czyli rządem. A tu mamy do czynienia z sytuacją taką, że od czasu powołania mamy de facto rząd wydmuszkę, by nie powiedzieć: masę upadłościową złożoną z resortów, których bądź już nie ma, np. technologii i przedsiębiorczości, energii i Skarbu Państwa czy środowiska, bądź de facto jeszcze nie ma, bo bez przypisania konkretnych kompetencji. To przede wszystkim klimat i aktywa państwowe. Nic. Dzisiaj procedujemy nie nad propozycją premiera czy rządu dotyczącą urządzenia władzy wykonawczej, a nad zgłoszonym przez posłów PiS koszmarkiem. Zmiana ma 58 stron, dotyczy kilkudziesięciu ustaw, podczas gdy pierwotna ustawa jest o połowę mniej obszerna. Przyjrzyjmy się zatem temu, jak to ktoś premierowi urządza rząd. Bo w grupie posłów - rzekomych autorów nie ma ani koalicjantów, ani członków rządu, których to dotyczy. Nawet sprawozdawca, jak wspomniałam, zapomniał się podpisać i musiał uzupełniać, że też popiera. Nie ma też posła członka Rady Ministrów w oczekiwaniu na tekę, niejakiego ministra Wosia, którego premier przecież w rozporządzeniu zobowiązał do przygotowania zakresu zadań, którymi w kadłubowym Ministerstwie Środowiska ma się zająć. Niestety w tym projekcie wbrew zapewnieniom klimatu też nie ma, bo nie wystarczy coś nazwać, by się stało. Z ministerstwa, które miało być do spraw polityki klimatycznej, została nazwa, czyli to, co już było w resorcie środowiska, plus kadłubkowe OZE, bo nawet nie wszystkie kompetencje w tym zakresie. Oczywiście bez najważniejszej kwestii związanej z klimatem ściśle, bez polityki energetycznej, która zostaje w dziale energia przypisanym ministrowi Sasinowi. Wygląda na to, że sprawy klimatyczne PiS sprowadza ewentualnie do smogu i śmieci oraz ugłaskania Brukseli i wyciągnięcia na ten cel pieniędzy z Unii. Nie dziwi to, bo w narodowym funduszu ochrony środowiska, który pozostaje w gestii ministra klimatu, pieniędzy już prawie nie ma, bo wydaje się je na inne rzeczy albo kieruje do Torunia albo na drogi samorządowe, a to przecież nie jest środowisko. A resort, dział środowisko?

I wreszcie najważniejsze, aktywa państwowe, czyli: wszystko, co mamy, Sasinowi oddamy, pozbawiając oczywiście koalicjantów fruktów, samemu premierowi też ograniczając wpływ. Patrząc na rozporządzenie premiera, jak i rozporządzenie ministra aktywów, które koncentrują władzę nad wszystkimi złotonośnymi, jeśli chodzi o posady i pieniądze, spółkami Skarbu Państwa w jednych rękach właśnie, możemy zobaczyć, że - jedno rozporządzenie premiera o wykazie spółek, które ukazało się w grudniu, drugie teraz właśnie, ministra Sasina, jeszcze przed tą ustawą, którą dopiero dzisiaj zaczęliśmy procedować - resortowi aktywów państwowych będzie podlegać ponad 200 podmiotów, spółek, instytutów. Oczywiście największe spółki, energetyka w rękach wicepremiera. Całość dobrze ilustruje filozofię rządzenia PiS: chaos i podział łupów. Ktoś, panie premierze - pana nie ma tu, to nie jest fundamentalna rzecz - urządza panu rząd. Czy pan o tym wie, czy pan może chce uniknąć odpowiedzialności?

Teraz głos ma pan poseł Wiesław Szczepański, klub Lewicy. Panie Premierze! W imieniu Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie nasze stanowisko co do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką, zawartego w drukach nr 158 i 158-A. Potrzebne są zatem zmiany w działach określających kompetencje poszczególnych ministrów. To kompetencja premiera. Na projekt ustawy w tym zakresie czekaliśmy ponad 2 miesiące. Chciałbym zapytać pana premiera: Czy brak było zgody w rządzie na podział kompetencji dla nowych ministrów? Dlaczego tak długo państwo czekaliście? Czy zaskoczył państwa podział łupów wśród koalicjantów po wyborach? Zaciekawia wywiad udzielony przez dziś jeszcze ministra bez teki pana Michała Wosia, który już 2 miesiące temu chwalił się, że będzie ministrem środowiska. Cóż pan minister powiedział? Na pytanie, co robił, będąc ministrem bez resortu, przez ostatnie 2 miesiące, i za co mu płacimy, odpowiedział: „W pierwszej kolejności za przygotowanie podziału. To rzeczywiście jest bardzo skomplikowana sprawa. Ta ustawa... zgodnie z moją wcześniejszą zapowiedzią nazajutrz po naszej ostatniej rozmowie 2 miesiące temu przekazałem panu premierowi projekt ustawy. To jest ustawa, którą wypracowaliśmy. Oczywiście ustawa, która dzieliła Ministerstwo Klimatu od Ministerstwa Środowiska czy w jakiś tam sposób przekształcała Ministerstwo Energii w Ministerstwo Klimatu, a z Ministerstwa Środowiska wyjmowała dwa departamenty, ta ustawa przerodziła się w większą ustawę, bo oczywiście doszły jeszcze aktywa państwowe” Projekt nie jest rządowy, lecz poselski, bo, jak twierdzi pan minister Michał Woś, „doszliśmy do wniosku wspólnie, że nasi posłowie taki projekt przedłożą, z tej racji, żeby sprawnie tego podziału dokonać” A może dlatego, że premier wstydził się firmować ten projekt i dostał polecenie polityczne, bo góra urodziła mysz? A więc za pieniądze publiczne pan minister Woś przez najbliższe miesiące w oczekiwaniu na wymarzony resort środowiska będzie, jak twierdził, dzielił, bo to nie są proste sprawy.

Również uzasadnienie projektu nie odpowiada przepisom art. 34 ust. 2 pkt 2 regulaminu Sejmu. Przedłożony projekt ustawy zakłada utworzenie działu administracji rządowej klimat. Część zakresu spraw objętych tym działem stanowi powtórzenie zakresu spraw objętych działem środowisko. Z projektowanej ustawy nie wynika, jaki zakres ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystania jego zasobów będzie należał do każdego z właściwych ministrów. Wątpliwości co do właściwości rzeczowej wydają się zasadne z uwagi na fakt, iż w projektowanym art. 28 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia projektodawca użył zwrotu „w szczególności”, co przesądza o przykładowym charakterze tego wyliczenia. Może zatem dojść do sporu kompetencyjnego pomiędzy ministrem właściwym do spraw klimatu a ministrem właściwym do spraw środowiska. W przypadku możliwej kontroli głównego inspektora ochrony środowiska przez obu ministrów wnioskodawcy nie wskazali, na jakiej podstawie zostanie wskazany organ, który wykonuje zadania kierownika jednostki kontrolującej wynikające z ustawy o kontroli administracji rządowej. Utworzenie działu administracji rządowej aktywa państwowe oznacza przywrócenie treści normatywnej istniejącego kiedyś działu Skarb Państwa. Nazwa ta wiąże się z obecną nazwą ministerstwa: Ministerstwo Aktywów Państwowych, w którego skład wchodzą komórki organizacyjne obsługujące sprawy z zakresu działów energia i gospodarka złożami kopalin. To nadzór nad mieniem państwowym, nad spółkami Skarbu Państwa. To tworzenie, panie premierze, taniego państwa, budowa Bizancjum, bo przecież tworzone ministerstwo otrzymuje dodatkowe miejsca w radach nadzorczych spółek, w fundacjach, agencjach, specjalnych strefach ekonomicznych, Banku Gospodarstwa Krajowego. Dziesiątki miejsc dobrze opłacanych, oczywiście dla swoich, za które zapłacą te podmioty. Domniemywam, że dziś są to nowi członkowie rady nadzorczej, a jutro będą to nowi członkowie zarządu. Ile to będzie kosztowało? Ile takich miejsc państwo potrzebujecie? Pełnię władzy minister aktywów przejmuje również w Radzie do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. Odwołujecie państwo wszystkich dotychczasowych członków, a w to miejsce powołujecie nowych, swoich. Projekt zakłada (Dzwonek) powstanie nowego ministerstwa związanego. Projekt zakłada powstanie również ministerstwa związanego z Unią Europejską, lecz - nie wiadomo dlaczego - sprawy związane z działalnością informacyjną i edukacyjną dotyczącą Unii przejmie minister spraw zagranicznych. Chciałbym zapytać, dlaczego to on będzie promował Unię Europejską, a nie minister właściwy do spraw Unii Europejskiej. Naprędce otrzymaliśmy wczoraj wrzutkę przenoszącą pełnomocnika do spraw równego traktowania z kancelarii premiera do ministerstwa polityki społecznej. Proponowane w ustawie 7-dniowe vacatio legis wydaje się zbyt krótkie, aby umożliwić reorganizację właściwych departamentów poszczególnych ministerstw, jeśli samo pisanie ustawy zajęło państwu 3 miesiące.

Dziękuję bardzo panu posłowi. Proszę teraz, aby w imieniu klubu parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 głos zabrała pani poseł Urszula Nowogórska. Szanowny Panie Marszałku! Przepraszam za głos, ale przeziębienie dopada czasem w najmniej odpowiednim momencie. Ale do rzeczy. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku sejmowym nr 158, wraz z autopoprawką, zawartą w druku sejmowym nr 158-A.

Jej szczególny charakter polegał na tym, że rozproszony po wielu ustawach zakres działalności administracji rządowej został po raz pierwszy uregulowany niemal w całości w jednej ustawie. Ustawa została oparta na konstrukcji działu administracji rządowej, rozumianego jako wydzielona część obszaru działania administracji rządowej co do zasady kierowana przez ministra. Dziś proponowane są kolejne zmiany w tej ustawie. Projekt zakłada dokonanie przesunięć niektórych zakresów spraw pomiędzy działami administracji rządowej, związanych z wyodrębnieniem dwóch nowych działów administracji rządowej, tj. aktywa państwowe oraz klimat. Dział aktywa państwowe, jak napisano w uzasadnieniu noweli, obejmuje sprawy dotyczące gospodarowania mieniem państwowym, w tym wykonywania procedur majątkowych i osobistych przysługujących Skarbowi Państwa, z wyjątkiem spraw, które na mocy przepisów odrębnych pozostaną we właściwości innych działów. Minister do spraw aktywów państwowych będzie reprezentował Skarb Państwa w zakresie gospodarowania mieniem państwowym. Proponuje się również, aby minister ten posiadał kompetencję inicjowania polityki państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego. Dział klimat natomiast będzie obejmował sprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju. W projekcie ustawy, który dzisiaj przechodzi pierwsze czytanie, zmierza się do zmian w ustawie o działach administracji rządowej, a także w 92 innych ustawach. Skala tych zmian, można powiedzieć, troszeczkę poraża. Ponadto przewiduje się szereg zmian w zakresie spraw objętych działem członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że projekt ustawy nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. Nasuwa się zatem pytanie, jaka rzeczywiście jest intencja wnioskodawców. Nasuwa się szereg różnych pytań. Po pierwsze, dlaczego tak szybko albo czemu tak późno? Minęły 3 miesiące. Na kolanie przygotowano autopoprawkę i przedstawiono nam ją bardzo, bardzo szybko. Czy nie powinno tam być napisane, że minister klimatu powinien zająć się programem „Czyste powietrze” Wyborcy w terenie, mieszkańcy różnych okręgów sygnalizują, że są bardzo poważne problemy z rozliczaniem tych projektów. Czy przypadkiem nie chodzi tu o dofinansowanie upadających spółek? Wcześniejsze zmiany doprowadziły do ogromnego rozproszenia. Powstały spółki matki, spółki córki. Czasem trudno się zorientować, kto czym rządzi i kto za co odpowiada. Jakie będą pozytywne efekty nowelizacji oprócz zwiększenia liczebności rad nadzorczych i zwiększenia wydatków na ten cel? Zastanawiamy się również, czy nie powstanie spór kompetencyjny pomiędzy Ministerstwem Klimatu a ministerstwem środowiska w wyniku wyodrębnienia działu klimat, ponieważ jak wynika np. z art. 13a ust. 1 ustawy o działach administracji rządowej, minister do spraw klimatu sprawuje nadzór nad głównym inspektorem ochrony środowiska, a organ ten zajmuje się m.in. monitorowaniem przyrody. W odniesieniu do działu aktywa państwowe wydaje się, że wnioskodawca zamierza przywrócić treść normatywną działu Skarb Państwa pod nazwą: dział aktywa państwowe, czyli można wnioskować, że to, co działało wcześniej, przez 8 lat, było rzeczywiście dobre. Szanowni Państwo! Klub Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 jest przeciwko wprowadzeniu chaosu i rozproszenia. Nie popieramy pisania prawa, pod którym kryją się ukryte mechanizmy. Nie podoba nam się pisanie prawa bez konsultacji, na kolanie i pod dyktando określonej grupy interesów, ale zależy nam na sprawności administracji państwowej i skuteczności państwa. Dziękuję bardzo, pani poseł. Teraz w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja głos zabierze pan poseł Krzysztof Bosak. Szanowni Państwo! Dokładnie w grudniu 2016 r. rząd przedstawił i uchwalił tutaj, w Sejmie, projekt likwidujący Ministerstwo Skarbu Państwa. Przypomnijmy, że odbyło się to po negatywnej ocenie sprawowania funkcji ministra skarbu państwa przez polityka PiS-u, który swoim postępowaniem doprowadził do tego, że rząd zapowiedział likwidację tego ministerstwa. Szanowni Posłowie PiS-u! Szanowni Ministrowie! To żaden wstyd wycofać się z błędnej decyzji. Bardzo dobrze, że po 4 latach poszli państwo po rozum do głowy i doszli do tego prostego wniosku, że jeżeli państwo jest właścicielem tak wielu spółek, to ktoś musi tym wszystkim zarządzać. Przejrzysta struktura, w której jest dział administracji rządowej odpowiadający za nadzór właścicielski, jest dobrą strukturą. Przypomnę tylko, że obiecywali państwo 100 mln zł oszczędności na ograniczeniu biurokracji i prognozowali państwo, że po 10 lat tych oszczędności będzie 1 mld. Minęły 4 lata, wycofują się państwo ze swoich strategicznych planów. Co więcej, żeby było śmiesznie, wycofujecie się państwo pod pretekstem projektu poselskiego. To jest jakiś żart, że proponujecie to państwo jako projekt poselski. Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt, a mianowicie że nadzorem właścicielskim przywracanego obecnie Ministerstwa Skarbu Państwa, które dla niepoznaki, żeby nie przyznać się do błędu, nazywacie w tej chwili Ministerstwem Aktywów Państwowych. Poza jurysdykcją tego ministerstwa będą ważne podmioty w naszym organizmie państwowym, które oczywiście nadzorują bardzo ważne spółki, kontrolowane pośrednio przez Skarb Państwa, a mianowicie przez Agencję Rozwoju Przemysłu i przez Polski Fundusz Rozwoju. Szczególnie w tym ostatnim podmiocie dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy, które są poza radarem opinii publicznej. Chciałbym też zwrócić uwagę, że wyzwaniem, które będzie stało przed odtwarzanym przez was obecnie, a wcześniej przez was zlikwidowanym, Ministerstwem Skarbu Państwa pn.: Ministerstwo Aktywów Państwowych, jest dokończenie prywatyzacji spółek, które nie mają charakteru strategicznego, tzw. resztówek. Drugą sprawą, której oczekujemy od rządu, jest prawidłowe zabezpieczenie interesów narodowych w spółkach o strategicznym znaczeniu, szczególnie w tych, w których rząd Platformy Obywatelskiej nieroztropnie, w celu zwiększenia swoich dochodów budżetowych, wyprzedał akcjonariat, schodząc na pakiety mniejszościowe i nie przewidując tego, że Unia Europejska może ingerować w zakres nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa nad tego typu spółkami.

Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zabranie głosu pana posła Grzegorza Brauna. Kłaniam się. Szczęść Boże, komu jeszcze nie mówiłem. Konfederacja nie popiera gry w trzy karty z obywatelami. Herbata od samego mieszania nie zrobi się słodsza. Szanowni państwo, nazywacie to ministerstwem aktywów, a my nazywamy to zintegrowanym systemem dostępu do koryta. Rozrywa was dwojaka tendencja: jednej strony zrobić dobrze własnym towarzyszom partyjnym, zwiększyć, pomnożyć liczbę stołków do obsadzenia, a z drugiej strony zrobić dobrze urzędnikom brukselskim, skonformizować Rzeczpospolitą względem poprawności politycznej. Tworzycie więc Ministerstwo Klimatu.

Zobaczcie: jest Ministerstwo Klimatu, a już na święta dzieci śniegu nie miały. Zastanówcie się nad własną twórczością. To w ogóle nie jest w porządku, że rząd - bo ma rację mój przedmówca, konstatując, że to jest w istocie projekt rządowy - zarządza, nie zaś wykonuje to, co tutaj Wysoka Izba by postanowiła. Dziękuję bardzo panu posłowi. Do pytań zapisało się dziewiętnaścioro państwa posłów.

Czas na zadanie pytania ustalam na 1 minutę. Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Chciałbym na początku powiedzieć, że to symptomatyczne, że rozmawiamy o przebudowie i reorganizacji rządu i nie przysłuchuje się tej dyskusji rzekomy autor tej zmiany, czy prawdziwy autor tej zmiany, czyli pan premier.

A zatem może potrzeba stworzenia nowego stanowiska. Mamy kolegę, który musi zostać ministrem, więc stwórzmy dla niego nowe stanowisko i nowe ministerstwo. Szanowni Państwo! Co jest prawdziwym powodem tego, że projekt jest sygnowany przez grupę posłów? Nie chcemy rozmów, dyskusji, boimy się rozmów o poważnych sprawach, bo to przecież ważne sprawy, te, którymi mają się zajmować nowe ministerstwa. W tej kadencji byłem już świadkiem sytuacji, w której rzekomi autorzy projektu, grupa posłów, i sprawozdawca występujący w ich imieniu nie znali odpowiedzi na elementarne pytania. To jest jeszcze większe kuriozum, że posłowie podpisują się pod zmianą dotyczącą kształtu polskiego rządu. Kim są posłowie? Bardzo proszę o udzielenie jeszcze odpowiedzi na pytanie, jakie będą koszty tej reformy, na piśmie. Dziękuję bardzo. Pytanie teraz zada pan poseł Ryszard Wilczyński, Koalicja Obywatelska. Rząd PiS ma 24 członków, historyczny rekord. Gratulacje.

Wiceministrów nikt nie policzy, jest to niepoliczalne, bo się kocą, i co chwila jest jakiś nowy. Panie ministrze, ilu macie wiceministrów w rządzie w tej chwili? Lepsze są tylko Węgry, w cudzysłowie, a więc mamy Budapeszt nad Wisłą, jeżeli chodzi o skład Rady Ministrów i liczbę wiceministrów. Kompetencje rządu są odwrotnie proporcjonalne do wielkości tego rządu, skoro posłowie muszą przedkładać ustawy o działach. Kompromitacja. Mateusz Morawiecki ogłasza votum separatum w sprawie zdolności Polski do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Polska nie spełni w 2020 r. wymagań co do 15-procentowego udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, ale za to mamy Ministerstwo Klimatu bez klimatu. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie zada pan poseł Waldy Dzikowski. Wysoka Izbo! Projekt ustawy zakłada wprowadzenie dwóch działów: aktywa państwowe i klimat. Ustawa o działach administracji rządowej jest fundamentem działania Rady Ministrów, w związku z tym nie tyle wydaje się, ile powinno tak być, że wymaga ona odpowiedniej rzetelności i staranności. Pamiętam, a wielokrotnie pracowałem w Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, że tam toczyła się żywa i bardzo czasochłonna debata. Zmiana ustawy o działach administracji rządowej wymaga oczywiście przeprowadzenia konsultacji przez Radę Ministrów z poszczególnymi ministrami, jak i przez komitet stały, w związku z tym oczywiście wydłuża to ścieżkę, ale to jest tak ważna ustawa, taki, że tak powiem, fundament działania Rady Ministrów, że ona wymaga takiej ścieżki.

Proszę o zadanie pytania pana posła Macieja Koniecznego, Lewica. Wysoka Izbo! Dlaczego zgłaszają to posłowie, a nie premier? Tego nie wiadomo. Co wiadomo?

Jak zadbać o dobrą rotację, to zmieści się sześciu. Do tego dojdą jeszcze jakieś sute odprawy i co, koledzy odwdzięczą się, wpłacając na partię, wpłacając na zaprzyjaźnione fundacje. Dobrzy koledzy to się odwdzięczą. Parafrazując klasyka: Dobrze się żyje, panie i panowie z PiS-u, dobrze się żyje. Szkoda, że głównie wam. A emerytom żałowaliście 1600 zł na minimalną emeryturę, ręka w rękę z liberałami z Platformy głosując przeciwko projektowi Lewicy. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Marek Dyduch. Nie, przepraszam bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

Rzeczywiście one będą coraz większe. Pytanie jest takie, czy będą zwiększały się również składy rad nadzorczych i zarządów w spółkach Skarbu Państwa, bo w tym projekcie ustawy jest wiele punktów dotyczących tego, że trzy ministerstwa ze sobą będą musiały uzgadniać różne rzeczy. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie zada pani posłanka Daria Gosek-Popiołek, klub Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od lat ekolodzy aktywiści alarmują, że główny inspektor ochrony środowiska tego środowiska nie chroni, podobnie jak regionalne inspektoraty. Ministerstwa Środowiska to właściwie do tej pory nie obchodziło. Kontrowersyjne decyzje, jak choćby w sprawie lokalizacji ferm przemysłowych na terenach cennych przyrodniczo - przykład Krynek i Kruszynian - zapadają i nikogo w ministerstwie to nie obchodzi. A teraz nie będzie to obchodziło aż dwóch ministerstw, bo zgodnie z przedstawionym projektem GDOŚ podlegać będzie de facto obydwu ministerstwom. Czy to celowe działanie? Bo to już nie jedno, ale dwa ministerstwa - i środowiska, i klimatu - będą udawały, że działanie i decyzje GDOŚ i regionalnych inspektoratów nie są ich sprawą. Dziękuję bardzo. Proszę teraz o zadanie pytania panią poseł Gabrielę Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Ale jak doniósł kolega z Lewicy, już się podobno przyznał minister Woś. Myślę, że kto pisał, to być może wiemy, ale nie wiemy, kto czytał. Mam wrażenie, że nikt.

Tymczasem tak nie jest. Kwestie polityki klimatycznej tylko w wąziutkim zakresie (Dzwonek) rozmawiania z Brukselą są przekazane, ale wszystkie kompetencje pozostają w dziale: energia i są przypisane ministrowi Sasinowi. Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Nie oceniając merytorycznie zawartości tego projektu ustawy, chciałbym zwrócić uwagę na procedurę i formy procedowania nad niniejszym projektem. Są oczywiście ustawy, które wymagają zastosowania tzw. szybkiej ścieżki legislacyjnej, ale składanie projektu ustawy o działach administracji rządowej przez posłów bez zachowania procedur i wymogów określonych dla projektów rządowych, czyli bez konsultacji i bez opinii, to z całą pewnością nie jest właściwa droga. Z zasadami prawidłowej legislacji, o której uczymy nasze dzieci w szkołach podstawowych i średnich, a studentów na studiach, nie ma to absolutnie nic wspólnego. I na koniec: nie chciałbym, żeby to było odebrane jako pewnego rodzaju zgryźliwość, ale jeżeli grupa posłów jest w stanie przygotować świetny projekt ustawy, liczący kilkadziesiąt stron, a nie jest w stanie zrobić tego rząd, to chyba niezbyt dobrze świadczy to o rządzie. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Konrada Frysztaka, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tym razem będziecie meblować gabinet premiera Morawieckiego, ale to wasza sprawa. Dzielicie między siebie łupy, w tym przypadku Polską Grupę Zbrojeniową. Polską Grupę Zbrojeniową, która powstała dzięki decyzji rządu Ewy Kopacz. To wtedy w Radomiu została zarejestrowana Polska Grupa Zbrojeniowa, która podlegała pod Ministerstwo Obrony Narodowej. A w tej chwili? Takie, że pan premier Sasin przeniesie sobie to do innego miasta ze szkodą dla Radomia, dla Radomia, który reprezentuję.

Proszę o zabranie głosu pana posła Tadeusza Tomaszewskiego, klub Lewica. Wysoki Sejmie!

Ale jest też jedna spółka specjalna, mianowicie jest spółka PL.2012+ w wykazie ujętym pod pozycją 186.

Natomiast członków rady nadzorczej i zarząd przejmuje (Dzwonek) pan minister Sasin. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania panią posłankę Magdalenę Biejat, klub Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie - właściwie nie wiem, czy do wnioskodawców, czy do rządu - dotyczące podziału Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Klimatu. Czemu to ma służyć? Wielokrotnie z tej mównicy i poza nią punktowaliśmy jako posłowie i posłanki Lewicy rząd, wskazując, że działania, które podejmuje, w najlepszym wypadku są pozorne, jeśli chodzi o ochronę klimatu, i nie robi się tutaj nic, żeby zapobiec katastrofie klimatycznej, w wyniku której już teraz zaczyna brakować latem wody w miastach, a ceny żywności zaczynają gwałtownie rosnąć. A więc pytam raz jeszcze: Czemu ma służyć wydzielenie Ministerstwa Klimatu i Ministerstwa Środowiska, wydzielenie w dodatku tak niekompetentne, że nie udało się dobrze podzielić obowiązków jednego i drugiego resortu?

Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Wiesław Szczepański, klub Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam dwa pytania.

Pytanie do posła sprawozdawcy: Jakie są powody, że część zadań dzisiaj przypisanych do części europejskiej, a więc promocja, informacja o Unii Europejskiej, znajduje się w sferach wpływu ministra spraw zagranicznych? Dlaczego o resorcie, który będzie zajmował się działaniem Polski w Unii Europejskiej, ma informować i chwalić Unię Europejską minister spraw zagranicznych?

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pani poseł Maria Małgorzata Janyska, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Pan poseł wnioskodawca, przedstawiając ten projekt, powiedział, cytuję: zawiera on priorytety, które chcemy realizować jako rząd PiS-u. Panie Morawiecki, czy pan abdykował, czy pan jeszcze o czymś nie wie, o czym wie pan poseł?

Dwóch premierów przemykało się tu co chwilę, ale widocznie jest to dla nich tak nudne, że szkoda ich czasu na tak ważny temat. Pan poseł powiedział również, że ta ustawa m.in. doprecyzowuje kompetencje ministrów. Doprecyzowuje kompetencje ministrów, a premierów nie ma, proszę państwa. Czy nie zależy im na kompetencjach, czy generalnie mają w nosie to, co się dzieje tutaj? Pan poseł powiedział także (Dzwonek), że dzięki temu projektowi będzie silna administracja rządowa, a silna administracja rządowa to silne państwo. Bardzo wiele zapisów, które są zawarte w tym projekcie, trzeba przerzucić na samorządy, bo one zagwarantują dobre rządzenie, a nie manipulacje polityczne. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wtedy opinia publiczna pod wpływem polityków Prawa i Sprawiedliwości, wtedy koalicji PO oczywiście, bardzo grzmiała, że zawłaszczamy państwo, że kolesiostwo, że partyjniactwo itd.

Co takiego się wydarzyło, że ci wszyscy, którzy nas wtedy umoralniali, że Lewica zawłaszcza władzę, dzisiaj zmieniają zdanie? Co takiego się wydarzyło, gdzie ta moralność? Zmieniła się Polska? Jest oszczędne rządzenie krajem? Bardzo dziękuję. Proszę o zadanie pytania panią poseł Małgorzatę Tracz, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej nie pozostawia żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia de facto z podziałem łupów, podziałem stanowisk w Lasach Państwowych, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spółkach węglowych pomiędzy koalicjantami Zjednoczonej Prawicy, koteriami i frakcjami. Ten projekt oraz ostatnie działania rządu nie dają nam żadnej podstawy do uznawania nowo powstałego Ministerstwa Klimatu za coś więcej niż ordynarny greenwashing waszego rządu. Nie dają nam żadnych złudzeń co do tego, jak traktowane są przez was kwestie kryzysu klimatycznego, transformacji energetycznej oraz ochrony przyrody. Złożony przez Koalicję Obywatelską projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu dotyczący powołania stałej komisji sejmowej do spraw klimatu trafił do sejmowej zamrażarki. Bo jak inaczej można interpretować to, że wciąż nie został rozpatrzony przez komisję regulaminową, do której trafił 22 listopada ub.r. [[Dzwonek]] projekt uchwały, który był wyrazem naszej woli współpracy z nowym ministerstwem na rzecz klimatu? Dlatego moje pytanie brzmi: Kiedy wyjmiecie projekt uchwały dotyczący powołania stałej komisji sejmowej do spraw klimatu z zamrażarki? Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Romuald Ajchler, klub Lewica. Wysoka Izbo! Lewica nie poprze tej ustawy. Boimy się jednej rzeczy, o której wspomniał pan poseł Dyduch. Poparlibyśmy każdą ustawę, która nie tworzy bytów politycznych, a ta ustawa właśnie to czyni. Ja osobiście się boję, że znowu powstaną nowe rady nadzorcze w tych nowych bytach. Trzeba będzie wypłacić ogromne pieniądze na odprawy różnym ludziom. Ale przede wszystkim ta ustawa charakteryzuje się tym, że jest dla tzw. swoich. Nie róbcie tego, nie idźcie tą drogą, jak mówił klasyk, jeszcze jest szansa. Wysoka Izbo! Otóż nie rozumiem jednej rzeczy.

Chodzi o to, żeby w tych kwestiach, o których decyduje większość, decyduje rząd, była zgoda, a nie żeby to był, jak się mówi, podział łupów. Ta ustawa właśnie to niesie. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Marek Sowa, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 3 lata temu politycy PiS-u pod szczytnym hasłem oszczędności likwidowali Ministerstwo Skarbu Państwa. Wówczas oczywiście nie chodziło o żadne oszczędności, chodziło tak naprawdę o dokonanie podziału łupów pomiędzy poszczególnych polityków PiS-u. Część trafiła do pani premier Szydło, część do Morawieckiego, do Ziobry, Gowina. Można by było wiele wymieniać. Sami się o tym przekonaliście, widząc, że to tak naprawdę doprowadza tylko do wielkich konfliktów wewnątrz waszego obozu. Dzisiaj przywracacie Ministerstwo Skarbu Państwa - zmieniona nazwa nic tutaj nowego nie wnosi. Ale co obserwujemy? Na czele komitetu, który będzie sterował podziałem łupów, postawiliście zaufanego człowieka prezesa Kaczyńskiego i on ma tam tych swoich przedstawicieli każdej grupki z waszego obozu. To jest skandaliczne i naganne zachowanie, to absolutnie w niczym nie doprowadzi do tego, aby zwiększyć efektywność zarządzania zasobami, aktywami państwowymi. Od 10 miesięcy w rządzie premiera Morawieckiego jest minister Woś. Chciałbym się zapytać: Co przez te 10 miesięcy robił, skoro nie miał resortu? Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zadanie pytania pana posła Tomasza Piotra Nowaka. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałoby się powiedzieć: panie premierze, ale pan premier jak zwykle Sejm ma. Delikatnie mówiąc, ma zdystansowany stosunek do Sejmu. A więc my jako zdystansowany Sejm zadajemy panu premierowi pytanie o zadania, które stoją przed tym rządem. A zadaniem fundamentalnym, które jest w tej chwili, jest transformacja przemysłu, energetyki, transformacja polskiej gospodarki w stronę gospodarki zeroemisyjnej. Jest to zadanie, na które trzeba odpowiedzialnie odpowiadać, czyli trzeba tak skonstruować ten rząd, ażeby realizował w pełni określone zadanie. Tymczasem mamy podział na ministerstwo aktywów i Ministerstwo Klimatu z niejasnymi kompetencjami i z niejasnymi wpływami jednego ministerstwa na drugie.

Teraz pytanie zada pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Nowelizacja ustawy o działach to projekt, który wcale nie wzmacnia aktywów państwowych, lecz wzmacnia pisiewiczów i podział łupów, czyli pracę dla swoich, jak to zwykle bywało. Ta ustawa jest nie do przyjęcia. Jak to jest, panie pośle sprawozdawco? Mówi pan, że celem tej ustawy jest doprowadzenie do optymalizacji i racjonalizacji oraz skuteczności administracji publicznej. To co, w chwili obecnej administracja publiczna jest nieskuteczna? Jak to jest, panie pośle? Dlaczego vacatio legis jest tak krótkie - 7 dni? W ciągu 7 dni to jest niewykonalne. Dlaczego ta ustawa jest projektem poselskim? Gdzie konsultacje społeczne, gdzie opinie? Tak nie można stanowić prawa. Piąty rok rządzicie, a niczego się nie nauczyliście. To zakłamanie to już po prostu. Jest tutaj na sali pan minister Woś. Panie ministrze, może miałby pan na tyle cywilnej odwagi i przyszedłby pan tutaj, powiedziałby pan, że napisał pan tę ustawę, że jest pan twórcą tej ustawy, bo tak pan powiedział w jednej ze stacji radiowych 20 stycznia i chwalił się pan, że pan napisał tę ustawę i przekazał premierowi. Niech pan się przyzna. Przestańcie kłamać. Bardzo dziękuję. Proszę teraz o zadanie pytania panią poseł Paulinę Hennig-Kloskę, Koalicja Obywatelska. Panie i Panowie Posłowie! Resortowi aktywów państwowych według rozporządzenia pana ministra będzie podlegać ponad 200 podmiotów, m.in. spółek, instytutów. Pan minister Sasin będzie nadzorować osobiście 27 spółek, w tym m.in. spółki energetyczne. Ale przy tej okazji chciałam pana ministra zapytać przede wszystkim o to, czy dalej będzie utrzymywała się tak duża rotacja na stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa, na zasadzie, żeby jeden robił miejsce drugiemu, bo każdy musi trochę zarobić, czy w końcu zacznie się jakieś strategiczne zarządzanie nakierowane na optymalizację zysków w tych spółkach. Natomiast chciałam też przy tej okazji zapytać pana premiera Gowina, czy stanowisko dla Zbigniewa Gryglasa i nadzór nad 69 spółkami w ramach ministerstwa aktywów (Dzwonek) to zapłata za poparcie ustawy kagańcowej, bo przecież nawet wasz senator mówił otwarcie w trakcie debaty w Senacie, że ta ustawa jest niezgodna z polską konstytucją, i chciał w tej sprawie składać poprawki.

Pytanie teraz zada pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Wysoka Izbo! To, że ta ustawa pozwoli jeszcze szybciej rosnąć najszybciej rosnącej grupie milionerów w Polsce, czyli milionerom z Prawa i Sprawiedliwości, jest oczywiste. Natomiast jedna rzecz, jedna zmiana budzi moje zaniepokojenie. Otóż tą ustawą Prawo i Sprawiedliwość przenosi pełnomocnika ds. równego traktowania z kancelarii premiera do ministra właściwego do spraw rodziny. To jest oczywiście, po pierwsze, taka zmiana, która de facto, można powiedzieć, obniża rangę funkcjonowania tego urzędu. Zmiana jest według wnioskodawców podyktowana koniecznością lepszej współpracy z pełnomocnikiem do spraw osób niepełnosprawnych.

Pytanie do wnioskodawców: Co spowodowało tak drastyczną zmianę, tak drastyczne obniżenie w tym projekcie rangi tego pełnomocnika? Pytanie zada pani poseł Krystyna Skowrońska, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku!

Przecież to jest rzecz skandaliczna. Państwo proponujecie, jak ma wyglądać ustawa, tzn. przygotowaliście ustawę o działach.

Pan premier to powiedział 5 marca. W 2015 r. zatrudnienie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wynosiło 559 osób, a w styczniu 2020 r. - 719. Czy chcecie państwo tym projektem ustawy powiedzieć, że aktualne będą słowa premiera?

Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Krutul z klubu parlamentarnego Lewica zamyka listę posłów zapisanych do zadania pytania. Wysoka Izbo! Proszę państwa, gdzie są konsultacje społeczne dotyczące tej ustawy? W którym miejscu suweren, o którym tak często wspominacie, może zabrać głos i wyrazić swoje stanowisko? Jak powiedział klasyk: ojczyznę dojną racz nam dać, Panie. Zastanówcie się. Dziękuję bardzo. Proszę o wystąpienie zastępcę szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pana Pawła Szrota. Bardzo proszę.

Szanowna Pani Przewodnicząca Skowrońska! Nie powinno być dla nikogo tajemnicą ani zaskoczeniem, ani jakimś szczególnym odkryciem, że projekt ten wnioskodawcy pisali w ścisłym porozumieniu, w ścisłej współpracy i w ścisłych uzgodnieniach ze stroną rządową.

Oczywiście rząd popiera rozwiązania zawarte w tej ustawie. Chodzi o uzgodnienie tego ze stroną parlamentarną.

Pan poseł Sowa pytał, co robił do tej pory minister Woś. Minister Woś został powołany na ministra członka Rady Ministrów odpowiedzialnego za organizowanie Ministerstwa Środowiska. Efekt jego pracy również dzisiaj szanowna Wysoka Izba rozpatruje. Jeśli chodzi o pytania, które były bezpośrednio kierowane do Rady Ministrów, chciałem udzielić właśnie tylu odpowiedzi. Na resztę pytań z całą pewnością odpowie przedstawiciel posłów wnioskodawców.

Dziękuję bardzo. W imieniu wnioskodawców głos zabierze pan poseł Jarosław Krajewski. Panie Marszałku!

Mogę je państwu, Wysokiej Izbie, przedstawić. Chodzi przede wszystkim o to, że projekt może spowodować skutki finansowe, które zostaną pokryte w ramach budżetu na 2020 r. Z moich informacji wynika, że w projekcie budżetu przedstawionym przez Radę Ministrów propozycje dotyczące zmian działów administracji rządowej zostały uwzględnione.

Otóż nie kto inny, jak dwie parlamentarzystki Platformy Obywatelskiej apelowały do rządu i do polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Wiecie państwo, co mówił wtedy pan poseł Wójcik reprezentujący klub Platformy Obywatelskiej? Mówił, że to jest naturalne prawo, że jest to prawo kształtowania przez większość parlamentarną, przez rząd, działów administracji rządowej. Nie jest to żaden precedens, nie dajcie sobie państwo tego wmówić. Niejednokrotnie projekty dotyczące działów administracji rządowej były przedstawiane jako projekty poselskie.

Otóż my jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość bardzo cenimy sobie dobrą współpracę z administracją rządową. Ten projekt, tak jak powiedział pan minister Szrot, był omawiany i konsultowany. Dobra współpraca ze stabilną większością parlamentarną jest wartością dodaną.

Jest również kwestia związana z tym, że państwo mówicie, jakie są intencje. Chodzi o optymalizację, racjonalizację i większą skuteczność zarządzania.

Kwestia konsultacji społecznych. Wiecie państwo, że jesteśmy osobami otwartymi na dialog, konsultacje i szukanie kompromisu.

Kwestia ochrony interesów Skarbu Państwa - temat wywołany przez pana posła Krzysztofa Bosaka. Panie pośle, proponujemy następujące rozwiązanie - minister aktywów państwowych będzie miał możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec decyzji o likwidacji przedsiębiorstwa państwowego.

Trudno jest mi wyobrazić sobie, żeby na tej sali w polskim parlamencie był parlamentarzysta, który miałby inny cel. Pani poseł mówiła, że wskazujemy, że silne i sprawne państwo potrzebuje przede wszystkim sprawnej administracji rządowej. Przez prawie 10 lat byłem samorządowcem w mieście stołecznym Warszawie i zdaję sobie sprawę z tego, jakie zadania spoczywają na administracji rządowej i jakie obowiązki spoczywają na jednostkach samorządu terytorialnego.

Myślę, że bardzo dobrze to świadczy, że poseł wnioskodawca identyfikuje się i wspiera rząd w tym zakresie, żeby przygotować rozwiązania prawne, które usprawnią i umożliwią wyjście naprzeciwko oczekiwaniom, również w kwestii klimatu. Mówiłem o polityce energetycznej, klimatycznej i ekologicznej. z tego powodu, że zdajemy sobie sprawę z tego, że rośnie choćby zainteresowanie obywateli polityką klimatyczną. Codziennie - myślę, że we wszystkich mediach albo w większości mediów - pojawia się informacja o smogu. A ja mieszkam w Warszawie, więc wiem, jaki to jest problem w mieście zarządzanym przez Platformę Obywatelską i prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Niestety wiem również o tym, że w tym zakresie Platforma Obywatelska w Warszawie zrobiła bardzo niewiele. Kwestia jeszcze jednego pytania - o pełnomocnika rządu ds. równego traktowania. Ta propozycja, która znalazła się w projekcie, zakłada jednoznacznie, że przeniesienie kompetencji pełnomocnika ds. równego traktowania do kompetencji ministra, który odpowiada za rodzinę, będzie równoznaczne z tym, że pozostaje zasada, że ten pełnomocnik jest oczywiście powoływany i odwoływany przez prezesa Rady Ministrów. W żadnym wypadku nie jestem w stanie zgodzić się z zarzutem, że jest to jakiekolwiek deprecjonowanie pełnomocnika. Te wszystkie zasady, które są określone w ustawach, które spoczywają dzisiaj na pełnomocniku, na panu ministrze, będą realizowane. Tutaj jest kwestia usprawnienia tej współpracy z ministrem, który odpowiada jako pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Taką rolę będzie pełnił pełnomocnik, ale - zgodnie z naszą propozycją - w ministerstwie, które jest odpowiedzialne za dział rodzina. Myślę, że ta sprawa nie wywołuje większych kontrowersji. Tych kontrowersji nawet teraz nie widzę na sali plenarnej. Dziękuję bardzo panu posłowi, przedstawicielowi wnioskodawców. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druki nr 46 i 110) Proszę pana posła Tomasza Latosa o przedstawienie sprawozdania komisji. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Zdrowia mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, druki odpowiednio nr 110 i 46. Szanowni Państwo! Jest to niezwykle potrzebna nowelizacja, o której mówiło się tak na dobrą sprawę od kilku lat. Mówiąc najkrócej: jedna z najważniejszych rzeczy, których ta ustawa dotyczy, jest związana z pionizacją struktury inspekcji sanitarnej, tak aby powiatowi inspektorzy byli w większym stopniu, niż to jest w tej chwili, niezależni od władzy lokalnej, aby mogli dla dobra bezpieczeństwa obywateli podejmować skuteczne, skuteczniejsze działania niż do tej pory w ramach swojej służby. To ustawa niezwykle ważna, niezwykle potrzebna. Żeby nie przedłużać - ponieważ mamy za chwilę głosowania - chciałem przekazać, że Komisja Zdrowia rekomenduje przyjęcie tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Wznawiam obrady. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam pod głosowanie. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia. Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy zawartego w drukach nr 158 i 158-A, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?

Sejm wniosek odrzucił, a tym samym skierował ten projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. proszę państwa,

Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 2. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Proszę zatem o zabranie głosu pana posła Czesława Hoca, który wygłosi oświadczenie w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli nie ma pana posła, to proszę, aby w imieniu klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej głos zabrał pan poseł Rajmund Miller. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, druk sejmowy nr 46.

uniemożliwiają panu wystąpienie, także koleżanki. Proszę bardzo.

Otóż ministerstwo nie zdecydowało się na powołanie tej komisji rządowej i zmiany, które dotyczą tak naprawdę części, która podlegała dotąd samorządowi, zostają wprowadzone bez zgody samorządu.

Nie może to następować ze złamaniem porządku prawnego. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten rząd w jednym jest do bólu konsekwentny, a mianowicie w okradaniu i deprecjonowaniu samorządu terytorialnego w Polsce.

Obniżyliście dochody samorządu terytorialnego.

Nie może być na to zgody parlamentu. Szanowni Państwo!

Samorządy terytorialne, samorządy powiatowe pomagają, również finansowo, w funkcjonowaniu powiatowych inspektoratów sanitarnych.

Szanowni Państwo!

Jeżeli odbierzecie im wszelkie kompetencje, również w zakresie nadzoru nad Państwową Inspekcją Sanitarną czy powiatową inspekcją sanitarną, to w jaki sposób będą oni mogli skutecznie wypełniać swoje obowiązki? A są za to odpowiedzialni. Szanowni Państwo! Ten projekt jest z natury zły, wpisuje się w tendencję rządu PiS-u do niszczenia samorządu terytorialnego, do odbierania mu kompetencji, w związku z tym nie ma na to zgody Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo, panie pośle. Już na sali jest pan poseł Czesław Hoc, który wygłosi oświadczenie w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Trudno się poważnie odnosić do takich argumentów. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić opinię w sprawie zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, druki nr 46 i 110. Można na wstępie stwierdzić: najwyższy czas. Nareszcie nastąpi powrót Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zarządzania hierarchicznego, dojdzie do przywrócenia funkcjonalnego podporządkowania merytorycznego. Wszystko po to, by usprawnić, ujednolicić i uporządkować funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu skutecznego, lepiej skoordynowanego nadzoru w zakresie zdrowia publicznego, wszak chodzi o zdrowie i życie obywateli, albowiem wszelkie decyzje w chwili zagrożenia epidemiologicznego bądź innych zagrożeń muszą być podejmowane bezzwłocznie, spójnie, profesjonalnie i efektywnie. Współczesna Państwowa Inspekcja Sanitarna to już nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa żywienia i żywności, warunków higieniczno-sanitarnych dotyczących personelu, sprzętu oraz pomieszczeń medycznych. To nie tylko profilaktyka chorób czy też nadzór nad warunkami w kwestii higieny środowiska w zakładach pracy, higieny radiacyjnej, procesów nauczania i wychowania czy też higieny wypoczynku i rekreacji. To także, a może nade wszystko, współczesne wyzwania: współdziałanie z innymi służbami w kwestii afrykańskiego pomoru świń, ognisk ptasiej grypy i świńskiej grypy, zapobieganie gruźlicy wielolekoopornej i koinfekcji gruźlicy i HIV.

Czy państwo wiecie, że od wielu lat nie ma ciepłej wody w budynkach Parlamentu Europejskiego ani w Strasburgu, ani w Brukseli? Być może nie mają tak sprawnych i profesjonalnych służb sanitarnych jak my w Polsce.

Jedynie pionowa struktura umożliwi ministrowi zdrowia sprawowanie skutecznego nadzoru w zakresie zdrowia publicznego oraz podejmowanie decyzji umożliwiających bezzwłoczne i adekwatne do zagrożenia działania służb sanitarno-epidemiologicznych w całym kraju. Skąd o tym wiemy? Po pierwsze, z kilkunastoletniego doświadczenia. Mieliśmy przykład niespójnego, nieskoordynowanego funkcjonowania w zakresie kompetencji organizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Chodzi o jasne zasady powoływania i odwoływania wojewódzkiego inspektora sanitarnego i powiatowego inspektora sanitarnego.

W tym momencie pragnę serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, że pomimo niedogodności organizacyjnych, znacznych problemów w nadzorze na poszczególnych szczeblach władzy oraz niezbyt satysfakcjonujących poprzednich uposażeń potrafili odpowiedzialnie, merytorycznie i z wielkim zaangażowaniem pracować na rzecz bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zasadniczo scentralizowanie struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również ustanowienie państwowego powiatowego inspektora można uznać za krok we właściwą stronę. Jest to jednak krok niewystarczający. Ten krok - zresztą nie pierwszy raz - to jest ustawa zrobiona, można powiedzieć, trochę po łebkach. Dlaczego? Warto w tym miejscu przytoczyć cytat z opinii Biura Analiz Sejmowych: „Celem projektu zmiany ustawy jest poprawa kompleksowości i skuteczności nadzoru nad Państwową Inspekcją Sanitarną, w skrócie PIS” Odnosząc się do konkretnych zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie ma żadnych racjonalnych przesłanek do odebrania organom jednostek samorządu terytorialnego prawa do występowania z wnioskami o podjęcie działań w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego lub o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia. Według Związku Powiatów Polskich - ale trzeba pamiętać, że podczas obrad komisji związek nie został dopuszczony do głosu, czyli strona społeczna - nie są znane przypadki, aby samorządy nadużywały do tej pory tej kompetencji. A wykreślony zapis z tego projektu ustawy umożliwiał szybkie reagowanie w przypadku zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców. Kto inny jak nie samorządy lokalne jest bliżej spraw obywateli i wydarzeń, które dzieją się w powiecie, gminie czy nawet dzielnicy.

Bardziej lokuje nas w okolicach koczowniczych plemion stepów centralnej Azji sprzed kilkuset lat. Wobec powyższych zastrzeżeń klub Lewicy przedkłada Wysokiej Izbie dwie poprawki do niniejszego projektu. Jedna dotyczy przywrócenia właściwych uprawnień samorządom, a druga - zapisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Dziękuję bardzo panu posłowi.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiam opinię Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 w sprawie rządowego projektu zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej planowane były przez obecną ekipę rządzącą praktycznie od 3 lat. Decyzyjność w tej sprawie Prawa i Sprawiedliwości jest zdumiewająca. Tak długo czekaliśmy na zmianę, która koncentruje się praktycznie jedynie na pionizacji podległości służbowej. Nie na takie zmiany czekała inspekcja sanitarna, szczególnie że miały one następować we właściwym czasie i były planowane od dłuższego czasu. Sanepid czekał na wsparcie finansowe, systemowe, przede wszystkim dotyczące wynagrodzeń pracowników, wsparcia laboratoriów, zmian organizacyjnych, uzbrojenia inspekcji w dodatkowe kompetencje, na unifikację procedur i działań przeciwepidemiologicznych oraz mechanizmów wprowadzenia polityki bezpieczeństwa sanitarnego oraz wielu, wielu innych kwestii, które wynikają z długiej praktyki działania sanepidu szczególnie na poziomie lokalnym. Zmiany, które planuje się w sanepidzie, polegają głównie na sposobie powoływania urzędników, co jedynie jest kolejnym etapem centralizacji władzy publicznej w Polsce. Dotyczyły one ośrodków doradztwa rolniczego, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, zarządów melioracji wodnej i urządzeń wodnych, spraw związanych z koordynacją świadczeń rodzinnych, 500+, które zostały cofnięte z urzędów marszałkowskich do wojewodów, nawet Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

A pamiętamy niedawną debatę dotyczącą BDO. Co by było, gdyby ktoś wcześniej pomyślał i zadania dotyczące przyjmowania wniosków skierował chociażby do powiatów? Nie byłoby tych dantejskich scen w urzędach marszałkowskich, które były w wielu miejscach naszego kraju. Bardzo żałuję, że przez te 3 lata pracy nad zmianą tej ustawy rząd nie wymyślił niczego, co moglibyśmy tu wspólnie zaakceptować.

Moja ocena dotychczasowego działania sanepidów, szczególnie w powiatach, jest dobra, szczególnie w tych uwarunkowaniach finansowych, w których inspekcja musiała się poruszać. Wiele dobrych inicjatyw własnych, bardzo dobra współpraca z samorządem i powiatowym, i gminnym, realizacja w 100% wszystkich programów krajowych z rozszerzeniem dotyczącym specyfiki danego powiatu. Wystawiam lokalnemu, powiatowemu sanepidowi za to co najmniej piątkę, jeżeli nie szóstkę, bo często sanepid wykraczał poza swoje dotychczasowe możliwości, które naprawdę nie były szerokie. Natomiast takim sztandarowym przykładem dobrego radzenia sobie na gruncie lokalnym i wykorzystania we właściwy sposób tej, można powiedzieć, niezależności, niespionizowania się, byłby chociażby przykład dotyczący dopalaczy kilka lat temu. Widzieliśmy wtedy, jak w tej sytuacji, która rozpoczęła się w Łodzi, a później miała miejsce we wszystkich częściach kraju, sanepid wespół z samorządem sobie radził, szczególnie z tymi sklepami, które mnożyły się i powstawały. Wtedy trzeba było nie lada sposobu i współpracy z odpowiedzialnym za to samorządem powiatowym, starostą, prezydentem, który pełni także funkcję starosty. Tylko dzięki właśnie takiej własnej inicjatywie i niezależności można było użyć sposobów, które uniemożliwiały powstawanie tych sklepów i zagrożenia ze strony dopalaczy dla młodzieży. Mówię w kontekście tego, w jakim stanie samorząd przejmował sanepid. Wszyscy, którzy byli w tamtym czasie starostami bądź działali w samorządzie powiatowym, pamiętają, że trzeba było dokupywać samochodów, trzeba było te budynki wyposażać, remontować. Wiele pieniędzy i zaangażowania powiaty włożyły w to, żeby ten sanepid wyglądał tak, jak dzisiaj wygląda. A dzisiaj co? Głos związku powiatów, głos związku miast nie był wysłuchany.

Stosowną poprawkę przedkładam na ręce pana marszałka. Dziękuję bardzo panu posłowi za wystąpienie w imieniu klubu parlamentarnego. Teraz pan poseł Janusz Korwin-Mikke, a następnie pan Grzegorz Braun zabiorą głos w imieniu Koła Poselskiego Konfederacja. Wysoka Izbo! Klub Konfederacji będzie głosował przeciwko. Nie widzimy powodu, żeby naruszać zasadę pomocniczości i centralizować coś, co scentralizowane być nie musi. Przy okazji chciałbym sprostować pewne użycie słów. Autorytarne to jest państwo oparte na autorytecie, a tu mamy do czynienia z budową państwa, które może wszystko. Nieprawda, chcą państwa prawa. To PiS jest partią demokratyczną i mając większość, ma prawo robić, co chce, bo demokracja polega na tym, że to jest tyrania większości i większość może robić z nami, co chce. Chcieliście państwo - tfu! - demokracji, to właśnie ją macie. Proszę państwa, ludzie pomordowani byli obywatelami polskimi i czy to byli Żydzi, czy nie, to trzeba by w każdym przypadku sprawdzać za pomocą ustaw norymberskich, czy to rzeczywiście byli Żydzi. Kolega Braun ma głos. Dziękuję, panie prezesie, za to sprostowanie. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak jest, Konfederacja to jest koło tworzone przez polskich państwowców, którzy z wielką powagą traktują potrzebę istnienia sprawnego, silnego państwa polskiego, ale silne państwo silnym będzie tylko wtedy, kiedy przestanie rozpraszać swoje siły na sprawy, którymi zajmować się nie musi, a nawet nie powinno. Sanepidy już dały się we znaki Polakom, którzy pragną zachować wolność w wyborze procedur medycznych, np. aplikowanych ich maleńkim dzieciom. W uzasadnieniu tego złego, niedobrego projektu zmiany prawa czytamy jakieś wzięte z sufitu dane na temat rzekomego wzrostu liczby Polaków, którzy nie aplikują swoim dzieciom przymusowych szczepień.

Powiadam: sanepidy dały się już we znaki, dlatego że jest tu ewidentny konflikt interesów. Sanepid z jednej strony jest obowiązany tym totalniackim, wciąż jeszcze na piśmie niesformułowanym, ale praktykowanym nakazem ścigać rodziców dzieci, którzy - powtarzam - żądają wolności i żądają respektu dla praw rodzicielskich w dziedzinie np. procedur medycznych, ale z drugiej strony sanepidy mają rejestrować przypadki występowania tzw. niepożądanych odczynów poszczepiennych.

No i skoro dzieje się to na szczeblu lokalnym w przypadku sanepidów, jeszcze rozśrodkowanych, lękamy się, że jeśli będziemy mieli jednego, centralnego, totalniackiego urzędnika od tych spraw, to także te niepożądane odczyny poustawowe będą jeszcze wzrastały. Stąd nie możemy popierać tego projektu, ale pragnę, żebyście państwo odnotowali, że nie czynimy tego ze skłonności do anarchizowania życia publicznego, tylko wręcz przeciwnie: z powodu naszego przywiązania do tradycyjnej, wspomnianej tutaj przez mojego znakomitego przedmówcę, zasady pomocniczości. To jest fundament naszej cywilizacji. Tej konstrukcji się trzymajmy. Dziękuję bardzo. Do pytań zapisało się 10 państwa posłów. Jeżeli nie, to zamykam listę. Ustalam jednocześnie czas na zadanie pytania na 1 minutę. Proszę, żeby pytanie zadał pan poseł Waldy Dzikowski, Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Otóż ten projekt, projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, to następny krok ku centralizacji naszego kraju.

Od dłuższego czasu toczy się debata, gdzie powinno być umiejscowione bezpieczeństwo np. sanitarne czy żywnościowe.

PiS wyznaje jednak zasadę taką, że silne państwo to duży rząd. My uważamy wręcz odwrotnie, że państwo obywatelskie, państwo zdecentralizowane, bliżej obywatela, pod jego kontrolą jest państwem bezpiecznym i takim, które daje gwarancję życia w zgodzie ze wszystkimi instytucjami i ze sobą. Dziękuję bardzo. Proszę o zadanie pytania pana posła Jacka Protasa, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Nie przedstawiliście żadnego argumentu, powtarzam: żadnego argumentu za tym, że konieczna jest pełna centralizacja inspekcji sanitarnej, że potrzebne jest odsunięcie samorządów, a konkretnie starostów czy też prezydentów miast na prawach powiatów od wpływu na funkcjonowanie powiatowych inspekcji sanitarnych. Moje pytanie brzmi: Czy macie dowody na to, macie przykłady tego, że starostowie nie radzą sobie we współpracy czy nie radzą sobie z pewnym nadzorem nad powiatowymi inspektorami sanitarnymi? Czy starostowie przeszkadzają? Czy te zapisy, które są dzisiaj, przeszkadzają w prawidłowym funkcjonowaniu powiatowych inspektoratów sanitarnych? Ja byłem starostą dwie kadencje i muszę wam powiedzieć, że gdyby nie pieniądze z budżetu powiatu, inspekcja sanitarna w powiecie (Dzwonek) by nie funkcjonowała.

Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Czesław Hoc, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Oto argumenty. Przykład jednego z absurdalnych rozwiązań poprzedniego systemu funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W województwie zachodniopomorskim wojewódzki inspektor sanitarny musiał pokonać drogę ze Szczecina do Sławna, ponad 200 km, by dokonać czynności kontrolno-nadzorczej dla podmiotów, których organem prowadzącym bądź założycielskim był powiat, np. szpital, dom pomocy społecznej, wszystkie szkoły ponadpodstawowe, bo nie mógł tego dokonać powiatowy inspektor sanitarny z powodu bezpośredniej podległości pod starostę, który powoływał i odwoływał powiatowego inspektora. Czyli nie mogła to być niezawisła decyzja i też byłby konflikt interesów. Ustawowy koszmarny, kosztowny absurd.

Dziękuję bardzo. Teraz pytanie zada pan poseł Zdzisław Wolski, klub parlamentarny Lewica. Ta ustawa jest dość typowa, bo istniały pewne nieprawidłowości i z jednej strony dobrze, że rząd się tym zajął - pewne sprawy porządkuje, ale niestety nie te dla sanepidu najważniejsze. Typowo dla siebie pokazuje swoje fobie, uprzedzenie, realizuje politykę wykluczeń, odpowiedzialności zbiorowej - myślę o tych elementach dezubekizacyjnych - ale jednocześnie z konsekwencją żelazną i niedobrą odbiera kolejne kompetencje samorządom. Nie ma. Przedmówcy o tym mówili.

Mówili o tym moi przedmówcy.

Dziękuję bardzo.

Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej podobno ma na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców. Ani z treści ustawy, ani z uzasadnienia nie wynikają jakiekolwiek korzyści dla przedsiębiorców, ale widać wyraźnie, że w tym projekcie odbiera się kolejne uprawnienia samorządom, w tym wypadku starostom, przenosząc je do administracji rządowej. W trakcie posiedzenia Komisji Zdrowia przewodniczący nie dopuszczał do głosu przedstawicieli Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich. Twierdził, że powinni uzgodnić, który z nich ma zabrać głos, a następnie, przy omawianiu kolejnych artykułów ustawy, twierdził, że już się wypowiadali, ignorując fakt, że wypowiadali się, ale w innej sprawie i w innym punkcie obrad komisji. Jeżeli rzeczywiście projekt tej zmiany ustawy nie był poddany opiniowaniu przez komisję wspólną, to jest to nie tylko kolejny przejaw arogancji ze strony rządzących, ale też złamanie obowiązującego w Polsce prawa. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Wojciech Maksymowicz, Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie ministrze, czy wobec informacji, które w ciągu ostatnich 2 dni dotarły do Polski, o zagrożeniu epidemiologicznym nowym koronawirusem, który podobnie jak SARS może zabić tysiące ludzi, a jego rozprzestrzenianie jest zawsze tajemnicą, dopóki nie wystąpi.

Chodzi o kompetencję i nie wypowiadajmy się w sprawach tak ważnych dla obywateli (Dzwonek), jeżeli widzimy to bardzo krótkowzrocznie i nie znając się na rzeczy. Tutaj jestem za absolutnie jasną kompetencją rządową, od góry do dołu, bo tylko to może nas uratować. Dziękuję bardzo. Pytanie zada pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ta ustawa buduje - po raz kolejny - brak zaufania do drugiego segmentu władzy publicznej, jakim są samorządy.

Przykłady pokazywały dobrą współpracę. Chciałem zapytać pana ministra, czy macie państwo informacje, jaką kwotą w ciągu 4 lat samorządy powiatowe i samorządy miejskie dofinansowały funkcjonowanie inspektorów sanitarnych na szczeblu powiatów. Po drugie, czy ta ustawa nadal zachowuje możliwość, elementy współdziałania samorządu powiatowego, samorządu gminnego z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym?

Dziękuję. Dziękuję. Pytanie zada pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! To, że nie akceptujecie samorządów, dało się odczuć wielokrotnie. Po raz kolejny działacie na szkodę jednostek samorządu terytorialnego. Jak możecie zabierać kompetencje samorządom, skoro jednocześnie chcecie, aby samorządy ponosiły odpowiedzialność? To niemożliwe. Widzicie wiele zagrożeń, a nie zauważacie tego, że najlepiej te zadania będzie wykonywał starosta, a nie - zamiejscowo - wojewoda. Te wasze zmiany są bardzo niekorzystne. Mam pytania. Czy ta reorganizacja zmieni finansowanie inspekcji sanitarnych? Czy otrzymają wystarczające środki finansowe na funkcjonowanie placówek? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o zadanie pytania pana posła Mirosława Suchonia. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To, że przedłożony projekt ustawy pozbawi inspekcje sporego wsparcia ze strony samorządów, które chcąc nie chcąc, do tej pory bardzo mocno finansowały działalność inspekcji, jest sprawą oczywistą.

I drugie pytanie: Czy w związku z tymi zmianami planowane jest wzmocnienie działań dotyczących komunikowania o zagrożeniach związanych z nieprzyjmowaniem szczepień ochronnych? Niestety istnieje spory ruch społeczny, który w oderwaniu od faktów próbuje prowadzić politykę antyszczepionkową.

Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytanie zada pan poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Mam wrażenie, że ten projekt jest kolejnym przykładem permanentnego dążenia do tego, ażeby jak najwięcej organów mających powiązanie z samorządem terytorialnym wyłączyć spod działania samorządu terytorialnego i stworzyć pionowe struktury podległe resortowi zdrowia. Na ten moment konstytucja wyraźnie wskazuje, że państwo polskie jest zbudowane na fundamencie zasady subsydiarności. A zasada ta wymaga bezpośredniego udziału poszczególnych wspólnot lokalnych i regionalnych w pełnieniu zadań administracyjnych, również dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa. I konkretne pytanie, panie ministrze: Czy Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego opiniowała ten projekt zmiany ustawy? Jest to projekt nowy, złożony w tej kadencji. Czy ten projekt stawał na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego? Dziękuję. Pytanie zada teraz pan poseł Romuald Ajchler, klub Lewica.

Ale przecież wiemy doskonale, że sanepid to nie tylko środki finansowe, to przede wszystkim sprawa zdrowia i bezpieczeństwa Polaków.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie teraz zada pan poseł Piotr Borys, Koalicja Obywatelska. Szanowny Panie Marszałku! Chciałbym zadać pytanie, które związane jest przede wszystkim ze skutecznością funkcjonowania całego systemu, który od strony konsumenta wymaga tak naprawdę tego, aby wszelkie instytucje... aby było przeświadczenie o pełnym bezpieczeństwie żywności.

Dziękuję bardzo. Lista osób zapisanych do pytań została wyczerpana.

Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za te pytania, one też pojawiły się w toku prac komisji, ale może raz jeszcze uda się udzielić na nie odpowiedzi. Zacznę od pytania pana posła Protasa, czy starostowie w jakikolwiek sposób nam przeszkadzają.

To jest sytuacja, co do której mieliśmy bardzo liczne sygnały od przedsiębiorców.

Pan poseł Hardie-Douglas pytał - i to pytanie się później powtarzało - czy ten projekt był przedmiotem opinii komisji wspólnej rządu i samorządu. Tak, oczywiście był.

Sytuacja, w której jest ta pionizacja, jest ta bezpośrednia podległość, na pewno sprzyja temu, aby ta współpraca przebiegała lepiej. Pan poseł Tomaszewski pytał, czy dysponujemy informacjami, jakimi kwotami samorząd dofinansowywał inspektorów sanitarnych.

Przecież z pewnością przyznacie mi państwo rację, mówię o krytykach tego projektu, że tymże starostom chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie swoich mieszkańców, a nie o obsadę stanowisk. Szanowni państwo, te środki były i pozostaną w części budżetowej dla poszczególnych wojewodów. W związku z tym nie ma tu jakichkolwiek przesunięć, nie ma jakichkolwiek zmian w tej kwestii. Natomiast jeżeli pytacie państwo o to, czy tych środków wystarczy, odpowiem w taki sposób: w zeszłym roku po raz pierwszy od wielu, wielu lat cała inspekcja sanitarna otrzymała istotne podwyżki. Kiedy państwo i państwa ugrupowania były u władzy tych środków na to, co w inspekcji sanitarnej jest najważniejsze, czyli na najlepszych ludzi, po prostu nie było. To też jest odpowiedź na pytanie pani poseł Pępek i na pierwsze pytanie pana posła Suchonia.

Jestem przekonany, że dalsza współpraca, tym razem już znacznie ściślejsza, pomiędzy inspekcją, głównym inspektorem a inspektorami powiatowymi przyczyni się do tego, że te działania będą jeszcze silniejsze i dadzą jeszcze lepszy efekty. Jak mówiłem, ona była.

Chcemy, żeby inspekcja sanitarna, przypomnę, że chodzi o 16 tys. pracowników na terenie całego kraju, była silniejsza, lepiej skoordynowana i w jeszcze lepszy sposób niż do tej pory wspierała obywateli, przedsiębiorców, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Pan poseł Ajchler pytał też o to, ile ta zmiana kosztuje. Według naszych szacunków nie ma mowy o żadnych dodatkowych kosztach, nie ma mowy o tworzeniu żadnych dodatkowych etatów. Raczej jesteśmy przekonani, że dzięki temu projektowi, dzięki tym zmianom ta inspekcja będzie działała znacznie lepiej niż do tej pory w ramach tych środków, które do tej pory były na to przeznaczane. Dziękuję bardzo panu ministrowi. Głos w dyskusji zabierze także sprawozdawca komisji pan poseł Tomasz Latos. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Dziękuję wszystkim państwu za dyskusję, dziękuję panu ministrowi za szczegółowe wyjaśnienia. Zostały zgłoszone poprawki, ale także wniosek o odrzucenie w drugim czytaniu. Przyznam, że z perspektywy dyskusji i na posiedzeniu komisji, i w przeszłości wokół potrzebnych zmian w inspekcji sanitarnej jest to dość zaskakujący wniosek, biorąc pod uwagę, że co do pewnych kierunków zmian do tej pory zawsze byliśmy zgodni. Komisja w dniu dzisiejszym się tym zajmie. Dziękuję bardzo panu posłowi. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Zdrowia w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedłożyła sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, druk nr 175. W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania. Marszałek Sejmu proponuje, aby w tym przypadku Sejm wyraził zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycje przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druki nr 63 i 126) Proszę pana posła Krzysztofa Szulowskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, druk nr 63.

Dodać należałoby, że niniejsza ustawa, aby kompleksowo zastąpić obecne regulacje zawarte w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, powinna wejść w życie razem z projektowaną ustawą o ochronie roślin przed agrofagami, a ta będzie procedowana jako następna. Przede wszystkim zadania z zakresu zdrowia roślin będą wykonywane, tak jak do tej pory, przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa będzie także wydawał, jak do tej pory, decyzje administracyjne w przypadku stwierdzenia występowania agrofagów kwarantannowych lub innych agrofagów podlegających obowiązkowi zwalczania. Tenże inspektor będzie także organem właściwym do prowadzenia urzędowego rejestru podmiotów zawodowych, który zastąpi rejestr przedsiębiorców prowadzony na podstawie dotychczasowej ustawy. Tenże inspektor będzie także wydawał świadectwa fitosanitarne, eksportowe oraz świadectwa fitosanitarne reeksportowe. Z kolei główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa będzie wydawał zgodę na prowadzenie prac badawczych z wykorzystaniem agrofagów kwarantannowych, agrofagów kwarantannowych dla stref chronionych oraz roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów, których wprowadzanie na obszar Rzeczypospolitej Polskiej lub stref chronionych jest zabronione. Główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa będzie także, jak do tej pory, reprezentował Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa na zewnątrz, w tym przekazywał Komisji Europejskiej oraz pozostałym państwom członkowskim Unii Europejskiej wymagane informacje z zakresu ochrony roślin. Tenże organ będzie też właściwy do wyznaczania stacji kwarantanny oraz miejsc zapewniających izolację. Szereg regulacji dotyczących organizacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa pozostaje bez istotnych zmian. Natomiast projektowana ustawa reguluje szczegółowo organizację i zasady funkcjonowania laboratoriów działających na potrzeby realizacji zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w tym zasady wyznaczania laboratoriów urzędowych i krajowych laboratoriów referencyjnych, działających w obszarze zdrowia roślin oraz środków ochrony roślin.

Stąd inspekcja będzie wykonywała zadania z zakresu kontroli i upraw GMO. Tak jak dotychczas, utrzymano uprawnienia dla głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do wydawania decyzji w sprawie przyznania odszkodowania za straty związane z wystąpieniem określonych agrofagów podlegających obowiązkowi zwalczania. Modyfikacji uległy także przepisy dotyczące powoływania i odwoływania wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Celem wprowadzanych rozwiązań jest zapewnienie większej możliwości oddziaływania głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa na pracę wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa i ich zastępców, ponieważ główny ciężar odpowiedzialności za realizację zadań wykonywanych przez wojewódzkich inspektorów spoczywa na głównym inspektorze. Zgodnie z propozycją wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa i jego zastępca powoływani byliby przez wojewodę w uzgodnieniu z głównym inspektorem ochrony roślin i nasiennictwa. Drugą istotną zmianą jest propozycja, aby wojewoda realizował obowiązki wobec wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępcy w zakresie wynagradzania i dyscypliny pracy w uzgodnieniu z głównym inspektorem ochrony roślin i nasiennictwa. Pozwoli to na uzyskanie przez głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa wpływu na motywowanie oraz wyciąganie konsekwencji służbowych wobec osób zajmujących te stanowiska. Zweryfikowane zostały także wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz ich zastępców. Uregulowane zostały zasady udzielania określonym osobom będącym pracownikami Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jak również niebędącym zatrudnionym w tej inspekcji upoważnienia do załatwiania spraw oraz przeprowadzania określonych czynności w imieniu głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Uprawnienia te będą mogły uzyskać osoby, które m.in. zdały egzamin przed komisją powołaną przez głównego inspektora z zakresu znajomości przepisów dotyczących spraw ochrony roślin przed agrofagami, środków ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzony zaświadczeniem. Ale w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie zniesiony został obowiązek cyklicznego powtarzania tego egzaminu jako nieuzasadnionego obciążenia pracowników Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W projektowanej ustawie wprowadzone zostało także pojęcie urzędowego inspektora. W ustawie przewiduje się zachowanie uprawnień Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do świadczenia określonych usług. Wprowadzono jednak warunek, iż nie może to wpływać negatywnie na wykonywanie przez nią zadań. Generalnie w oparciu o dotychczasowe regulacje określono zasady nakładania w czasie kontroli plomb w celu uniemożliwienia zmiany tożsamości lub zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów lub zmiany tożsamości agrofagów, środków ochrony roślin lub materiału siewnego, a także sposób udzielania zgody na ich zdjęcie. Wprowadzono rozwiązania umożliwiające wykonanie obowiązków właściwych organów dotyczących pobierania próbek w przypadku towarów oferowanych na sprzedaż za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w tym Internetu. Określono zasady współpracy inspekcji z innymi służbami, w tym z Policją i strażą gminną (miejską), oraz organami administracji rządowej i samorządowej. Regulacje te mają na celu zapewnienie efektywności przeprowadzanych czynności kontrolnych oraz wydawania decyzji administracyjnych. Uregulowano organizację oraz zasady funkcjonowania laboratoriów wykonujących badania na potrzeby Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa - chodzi o wyznaczanie laboratoriów urzędowych oraz krajowych laboratoriów referencyjnych i ich obowiązki. Jednym z głównych warunków wyznaczenia urzędowych laboratoriów w obszarze ochrony roślin przed agrofagami jest posiadanie przez te laboratoria akredytacji w zakresie stosowanych metod w całym zakresie analitycznym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, co musi być potwierdzone certyfikatem wydanym przez krajową jednostkę akredytującą. Do tej pory laboratoria te nie były objęte takim wymogiem. Projekt zakłada zmianę podległości laboratoriów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z podległości wojewodom w ramach wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa na podległość głównemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa w ramach Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zmiany te mają na celu zwiększenie efektywności pracy laboratoriów, lepsze wykorzystanie zasobów finansowych i osobowych oraz ograniczenie kosztów związanych z realizacją zobowiązań. W toku procedowania ustawy zgłoszono szereg poprawek, ale tylko o charakterze legislacyjnym. W głosowaniu przyjęto projekt ustawy bez głosów sprzeciwu. W imieniu komisji rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie projektu ustawy. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Głos ma poseł Kazimierz Gołojuch, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko mojego klubu co do projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Projektowana ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego przepisy nowych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady regulujących sprawy zdrowia roślin.

Proponuje się przy tym zmianę organizacji laboratoriów inspekcji i przeniesienie ich ze struktur wojewódzkich w ramach wojewódzkiej administracji zespolonej na rzecz podległości głównemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa. Nadmienię, że w obszarze nasiennictwa zachowane zostaną wszelkie rozwiązania krajowe.

Projektowana ustawa określa skutki finansowe wejścia w życie zarówno tej ustawy, jak i projektowanej równolegle ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Panie Marszałku! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie projektu procedowanej ustawy. Dziękuję bardzo. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pani poseł Dorota Niedziela. Wysoka Izbo!

Jak mówiłam, jest to dosyć obszerna, techniczna ustawa, która wymaga dogłębnych analiz dokonanych przez specjalistów.

Bardzo proszę o konkretne przemyślenie sprawy zmiany definicji materiału siewnego. Dziękuję bardzo, pani poseł.

Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Lewicy w sprawie projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jest ona bardzo ważna, dotyczy m.in. bezpieczeństwa żywności i ma także rozwiązywać problemy związane z pracą inspekcji czy jakością pracy laboratoriów i ich organizacją. Mamy więc do czynienia z jednej strony z koniecznością dopasowania naszych przepisów do przepisów unijnych, a z drugiej - z kwestią organizacji pracy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Niestety ta ustawa nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z pracą pracowników inspekcji, pracą laboratoriów czy z bezpieczeństwem żywności. A zatem sygnalizujemy, że jako klub uważamy, że kontrola bezpieczeństwa żywności w Polsce jest niedostateczna, co naraża Polaków na liczne choroby wynikające ze stosowania zbyt dużych ilości często nielegalnych środków ochrony roślin, antybiotyków oraz nieprzestrzegania karencji w ich stosowaniu.

Problemem jest także brak nadzoru na poziomie powiatów i umocowanie inspektorów na poziomie województw.

Dziękuję serdecznie.

Proszę, panie pośle.

Rzeczywiście pani poseł Niedziela ma rację.

Dziękuję bardzo. Zapraszam panią poseł Jagnę Marczułajtis-Walczak z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Proszę się nie spieszyć.

Pani poseł, zapraszam serdecznie, z uśmiechem na twarzy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Czy dokumenty stanowiące dowód poniesienia strat w związku z występowaniem agrofagów zostaną określone rozporządzeniem ministra właściwego do spraw rolnictwa? Pytanie drugie: Co oznaczają „kompetencje kierownicze”, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 5? Co oznacza „wiedza w zakresie”, skoro planowana jest rezygnacja z wykształcenia rolniczego? I z jakiego powodu planowana jest rezygnacja z wymagania wykształcenia rolniczego? Wprowadzenie nowego pojęcia wymaga zdefiniowania w projektowanych przepisach. Nie jest wystarczające podanie w uzasadnieniu informacji, że (Dzwonek) jest on odpowiednikiem państwowego inspektora, zwłaszcza że zakres jego działania także - zgodnie z informacjami podanymi w uzasadnieniu - ulega rozszerzeniu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Kazimierza Plocke z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym się dowiedzieć, w jaki sposób będą rozstrzygnięte kwestie dotyczące laboratoriów. Czy obecnie funkcjonujące laboratoria w gestii państwowego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa będą przechodzić nową procedurę, żeby uzyskać certyfikację? A jeśli tak, czy to będzie w oparciu o unijne przepisy? I jeśli tak, to jaki będzie koszt tej certyfikacji?

Dziękuję serdecznie, panie pośle. Zapraszam panią poseł Dorotę Niedzielę z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Powrócę do tematu materiału siewnego i definicji dotyczącej materiału siewnego, która zostaje zmieniona. W naszej ocenie ta zmiana nie będzie dobrą zmianą.

Ale ja chciałabym zapytać, czy to rzeczywiście tak będzie, czy nie będzie dualizmu materiału siewnego, z którym będzie miała problem inspekcja nasienna.

Dziękuję, pani poseł. Zapraszam podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana ministra Rafała Romanowskiego. Panie ministrze, 15 minut jest do pana dyspozycji. Proszę bardzo. Wysoka Izbo!

Ale podczas pierwszego przedłożenia Wysokiej Izbie wyjaśniałem, dlaczego ta procedura została wydłużona. Projekt ustawy jednej i drugiej był przedłożony i przyjęty przez rząd w poprzedniej kadencji, ale właśnie w związku z tym musiał być ponownie przedłożony rządowi i przedstawiony pani marszałek do rozpatrywania. Aczkolwiek wszystkie te przepisy, które nas obowiązują, jeżeli chodzi o wykonywanie przepisów unijnych, w pełni są realizowane. Pan poseł Ajchler po raz kolejny poruszył kwestię plomby.

Kwestia postępowań konkursowych. Nadal są przeprowadzane postępowania konkursowe. Wprowadzone jest tylko i wyłącznie wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, staż pracy minimum 6-letni, w tym 3-letni na stanowisku kierowniczym. Tak jak państwo słusznie zauważyli, jest wykreślone wymagane wykształcenie rolnicze, ale to tylko i wyłącznie ze względu na praktykę i doświadczenie głównego inspektora sanitarnego. Po prostu w bardzo wielu postępowaniach konkursowych wielu kandydatów nie spełniało tych podstawowych warunków i postępowania konkursowe w województwach były z tego powodu powtarzane do momentu znalezienia właściwego kandydata, który spełniał to ustawowe kryterium. Stąd m.in. właśnie ta zmiana w ustawie, jeżeli chodzi o strukturę laboratoriów, które przejdą ze struktury wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa pod głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Tak jak przecież w przedłożeniu przedstawiałem, te laboratoria będą wymagały nowej akredytacji, zgodnie z przedmiotowymi rozporządzeniami Unii Europejskiej.

Obejmuje ona wszystkie takie nasiona, tj. nasiona, które są kwalifikowanym materiałem siewnym, oraz nasiona, które nie były poddawane ocenie i tych wymagań nie spełniają, ale są przeznaczone do siewu. W praktyce oznacza to, że do obrotu, czyli do sprzedaży z przeznaczeniem do siewu, nie będzie można wprowadzać niekwalifikowanego materiału siewnego. Taka reguła będzie miała zastosowanie do wszystkich podmiotów, tj. przedsiębiorców prowadzących obrót materiałem siewnym oraz rolników, którzy będą sprzedawać niekwalifikowany materiał siewny innym rolnikom. Taka regulacja przyczyni się do porządkowania rynku materiału siewnego, będzie chronić rolników przed przedsiębiorcami sprzedającymi do siewu niekwalifikowany materiał siewny. Przyniesie również korzyści przedsiębiorcom legalnie wprowadzającym materiał siewny do obrotu. Zasady w nasiennictwie dotyczą obrotu nasionami, tj. nie mają zastosowania do stosowania nasion we własnym gospodarstwie. To też powinno wybrzmieć, bo nad tym też dyskutowano bardzo mocno na posiedzeniu komisji rolnictwa. Natomiast kwestie wnoszenia przez rolników dla hodowców opłat od rozmnożeń własnych dotyczących odmian chronionych wyłącznym prawem dla odmiany są uregulowane w ustawie o ochronie prawnej odmian roślin. A ta ustawa o ochronie prawnej odmian roślin nie jest zmieniana, jeżeli chodzi o przedmiotowy projekt. Dziękuję serdecznie. O głos proszę sprawozdawcę komisji pana posła Krzysztofa Szulowskiego. Panie pośle, 15 minut do pana dyspozycji. Proszę bardzo. Wysoka Izbo! Nie było tutaj pytań wprost skierowanych do mnie. Mimo obszerności ustawy, mimo tego, że materia tej ustawy jest tak obszerna, prace przebiegły sprawnie, nie było wielkich kontrowersji. Chciałbym się tylko odnieść do jednej kwestii, do bardzo ważnej kwestii, która jest poruszana w ustawie, dotyczącej akredytacji laboratoriów badawczych.

Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druki nr 62 i 125) Bardzo proszę pana posła Zbigniewa Dolatę o przedstawienie sprawozdania komisji. Proszę, panie pośle. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Zawarta jest ta ustawa w druku nr 62, a sprawozdanie - w druku nr 125. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła projekt ustawy na posiedzeniu w dniu 7 stycznia.

Projektowana ustawa ma zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o ochronie roślin z 18 grudnia 2003 r. Przyjęcie przepisów zawartych w projekcie ustawy jest bardzo ważne w kontekście konieczności udoskonalenia systemu chroniącego zdrowie roślin narażonych na liczne, w tym nowe, agrofagi oraz zapewniającego bezpieczeństwo w międzynarodowym obrocie produktami pochodzenia roślinnego. W trakcie prac komisji zgłoszono i przyjęto jedną poprawkę. Poprawkę tę zgłosiła pani poseł Dorota Niedziela. Poprawka dotyczy art. 56 i odnosi się do pobierania opłat za kontrolę przez głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa lub wojewódzkich inspektorów ochrony roślin. Precyzuje ona, że opłaty za kontrole niezbędne do wydawania świadectw eksportowych będą pobierane 14 dni po doręczeniu rachunku, a nie przed kontrolą. Pragnę w tym miejscu podkreślić, że poprawka była zgłoszona przez polityka opozycji. Opozycja często podkreśla albo skarży się, że poprawki są odrzucane. To nieprawda. Jeśli są merytoryczne, to są przyjmowane. Mam nadzieję, że będzie więcej właśnie takich przykładów solidnej, merytorycznej pracy, a nie krytyki dla krytyki. Ponadto komisja przyjęła szereg poprawek redakcyjno-legislacyjnych, które zostały zgłoszone przez Biuro Legislacyjne. Komisja jednogłośnie przyjęła projekt ustawy i dlatego w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwracam się z wnioskiem, aby Wysoki Sejm raczył uchwalić projekt ustawy z druku nr 125. Dziękuję serdecznie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Zapraszam serdecznie pana posła Jerzego Małeckiego z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt kolejny raz przedstawić oświadczenie dotyczące rządowego projektu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, który zawarty jest w druku nr 62. Projekt dotyczy wprowadzenia rozwiązań ograniczających ryzyko zawleczenia do Polski tzw. nowych agrofagów, m.in. obcych wirusów, bakterii, grzybów czy szkodników, które atakują rośliny. Jego celem jest także wprowadzenie do krajowego porządku prawnego postanowień prawa europejskiego. Ochrona roślin przed agrofagami ma istotne znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska naturalnego. Zwalczanie nowych patogenów wymaga dodatkowych zabiegów ochronnych, co podnosi koszty produkcji. Wystąpienie nowych patogenów może negatywnie wpływać także na eksport naszych płodów rolnych. Myślę, że potrzeba przyjęcia tego projektu nie budzi żadnych wątpliwości. Dano temu wyraz - jak to przed chwileczką przedstawił pan sprawozdawca komisji rolnictwa - właśnie podczas prac sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która jednogłośnie go przyjęła. W związku z powyższym Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość opowiada się za przyjęciem rządowego projektu ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Zapraszam pana posła Kazimierza Plocke z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze! Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska poprze rządowy projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami. Pierwsze dotyczy środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, a drugie dotyczy kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych w celu zastosowania prawa paszowego, żywnościowego, zdrowia roślin i środków ochrony roślin. Ochrona roślin przed agrofagami na bardzo duże znaczenie gospodarcze. Jest ważna z punktu widzenia gospodarki narodowej, a także środowiska naturalnego. Proces ochrony roślin w Polsce uzyska nowy wymiar prawny, który będzie odbywał się w oparciu o nowe rozwiązania zaproponowane przez rząd, a wynikające z przepisów europejskich. Ważność tego projektu polega na ograniczaniu ryzyka introdukcji na obszar konkretnego państwa nowych organizmów szkodliwych dla roślin mogących spowodować stratę w uprawach rolnych bądź leśnych. Dobrze wiemy, że temu procesowi w ostatnich latach towarzyszy, po pierwsze, intensywny rozwój handlu zagranicznego czy też zmiany klimatyczne. Przyjęcie zaproponowanych rozwiązań zwiększy kontrolę nad obrotem produktami i towarami pochodzenia roślinnego w wymianie międzynarodowej. Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Żeby nie przedłużać: Projekt został omówiony bardzo dokładnie i szczegółowo, dlatego jeszcze raz powtarzam, że nasz klub będzie głosował za przyjęciem analizowanego projektu ustawy. Zapraszam pana posła Romualda Ajchlera z klubu parlamentarnego Lewicy. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Otóż, jak pan widzi i słyszy, projekty ustaw rolniczych mają szczęście.

Bo na pewno nie ma i nie byłoby zgody Lewicy na to, aby poprzeć projekt ustawy, który nie odpowiada naszym warunkom. Ten projekt ustawy mało tego, że odpowiada warunkom Lewicy i pozostałej opozycji, ale także odpowiada przede wszystkim polskiemu rolnictwu i bezpieczeństwu żywnościowemu, a także bezpieczeństwu tych, którzy spożywają artykuły rolno-spożywcze. A tutaj, w tym przypadku, jeśli chodzi o sprawy roślinne, to także zabezpiecza te rośliny przed agrofagami.

Zresztą wie pan doskonale, że przy tego typu ustawach są głosy „za” i są głosy „przeciw” Rzeczywiście pani poseł Niedziela była autorką poprawki, z którą nie mogliśmy się wszyscy jako opozycja zgodzić, ale m.in. ja również w imieniu Lewicy podpisałem tę poprawkę, bowiem uważam, że jeśli się wykonuje przez instytucje państwa jakąś usługę, to już kto jak kto, ale państwo nie powinno wchodzić w to przed wykonaniem tej usługi, tylko w normalnym interesie jest, aby dokonało tego po. Ale podczas tej debaty zapytałem pana ministra.

My nie dyskutujemy, przyglądamy się tylko tej kwestii.

Bo ja oceniam - i prosiłbym, aby pan minister sprostował, jeśli nie mam racji, zresztą możemy na ten temat podyskutować - że 80% tej ustawy to jest twórczość naszych urzędników, którzy w różny sposób przypisują sobie uprawnienia, a 20% jest to autentycznie kwestia przystosowania przepisów do prawa unijnego.

Przed chwilą debatowaliśmy na temat innych ustaw.

Macie pomysły na to, co zrobić, żeby obniżyć podatki i zmniejszyć przez to wpływy samorządów, jeśli chodzi o dochody, to musicie mieć pomysły na to, w jaki sposób zrekompensować także im utratę tych dochodów.

Ale, jak mówię, wystrzegajcie się tego państwo.

do prawa unijnego. Nie korzystajcie z tej okazji i niech pan ograniczy twórczość swoich urzędników, wtedy Lewica na pewno was poprze. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W rządowym projekcie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami, druki nr 62 i 125, przewidziano rozwiązania ograniczające ryzyko zawleczenia do Polski tzw. nowych agrofagów, tj. m.in. wirusów, bakterii, grzybów czy szkodników, które atakują rośliny. Zmiana przepisów dostosowuje polskie prawo do rozporządzeń i dyrektyw unijnych. Ochrona roślin przed agrofagami ma istotne znaczenie zarówno dla gospodarki, jak i środowiska naturalnego. Agrofagi niszczą m.in. plony, a także powodują znaczne ubytki w drzewostanach. Ich zwalczanie wymaga dodatkowych zabiegów w zakresie ochrony chemicznej lub działań kwarantannowych, co podnosi znacznie koszty produkcji. Wystąpienie w Polsce nowych agrofagów może mieć negatywny wpływ na eksport płodów rolnych.

Agrofag ten spowodował w Irlandii katastrofalny głód. W ostatnich dekadach w Europie odnotowano przypadki wystąpienia nowych agrofagów, co uzasadnia wzmocnienie dotychczasowych przepisów dotyczących eksportu i importu. Przykładem może być nowa bakteria, która zagraża ponad 300 gatunkom roślin. Najczęściej porażane są przez nią gatunki roślin o znaczeniu gospodarczym dla Polski. Mówimy tutaj o wiśni, czereśni, śliwie, tudzież innych gatunkach. Najważniejsze zadania związane ze zdrowiem roślin będą wykonywane jak do tej pory przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Organem, który będzie przeprowadzał kontrolę dotyczącą spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu unijnym, jak również kontrolę występowania agrofagów, będzie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa. Wojewódzki inspektor będzie także wydawał jak obecnie decyzje administracyjne w razie stwierdzenia występowania tzw. agrofagów kwarantannowych lub innych agrofagów podlegających zwalczaniu. Nowością będą możliwości wyznaczania obszarów wolnych od określonych agrofagów, co powinno ułatwić eksport towarów do państw trzecich, poza Unię Europejską. Obszar wolny od określonego agrofaga będzie ustanawiał wojewoda. Ograniczenia lub nakazy obowiązujące na takim obszarze będą natomiast wynikały z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Komisja przyjęła poprawkę dotyczącą zmiany terminu dokonywania opłaty pobieranej przez głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa bądź właściwego wojewódzkiego inspektora. Opłaty uiszczane będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia rachunku.

Zasadne by było, aby obligatoryjnie były to studia wyższe o kierunku rolniczym lub pokrewnym. Właściwe pod względem merytorycznym wykonywanie obowiązków wymaga posiadania ogromnej wiedzy rolniczej, specjalistycznej wiedzy.

Chciałbym ponadto zwrócić uwagę - mam prośbę do pana ministra - że jeśli chodzi o pracowników tej sfery, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo żywnościowe narodu, wysokość stawki wynagrodzenia korpusu służby cywilnej zależy od kwoty bazowej i mnożnika.

Pracownicy dzisiaj pracują na prowizorium budżetowym. Nie wiedzą, jakie będą otrzymywać pensje w tym roku.

Pracownicy tej administracji, którzy odpowiadają za tak ważną dziedzinę gospodarki narodowej, apelują o przyjrzenie się ich pensjom (Dzwonek), tym bardziej że jest to w skali kraju 1870 zatrudnionych osób. Dziękuję serdecznie. Przechodzimy do zadawania pytań. Ustalam czas zadawania pytań na 1 minutę. Zapraszam pana posła Romualda Ajchlera z klubu parlamentarnego Lewicy, tak mając dystansik, mówię, że Lewicy, a nie SLD, panie pośle. To są przyzwyczajenia. Za chwilę pewnie się ich wyzbędę, ale to jeszcze kwestia chwili. Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Chciałbym się dowiedzieć, czy macie państwo jakieś wyliczenia, co nam grozi w tych sprawach, jakie jest niebezpieczeństwo.

Uporaliśmy się z tym. Boję się, żeby czasem, przypadkiem nie dotyczyło to produkcji roślinnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Panie ministrze, ma pan 15 minut. Jak będzie krótko, to będę się do pana ciepło uśmiechał. Wysoka Izbo!

Ale kilka takich dosyć istotnych informacji, które pojawiły się i wręcz wzbudziły mój głęboki niepokój. Panie Pośle Ziejewski! Znamy się wiele lat. Prowizorium budżetowe, ustawa budżetowa to jest jedyna ustawa, która podlega czterem czytaniom. Zależy tylko i wyłącznie od trybu procedowania przez Wysoką Izbę, kiedy budżet państwa będzie przyjęty. Pamiętajmy o jednej podstawowej rzeczy: w ustawie budżetowej w roku 2018, jeżeli chodzi o Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, została zagwarantowana podwyżka dla tej inspekcji dla każdego etatu w wysokości 400 zł. W roku 2019 było to 530 zł. W roku 2020 w projekcie ustawy budżetowej, który jest w tej chwili procedowany, jest 6% zagwarantowanej podwyżki dla Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, więc nie wiem, z czego pan poseł wyczytuje, że w ramach prowizorium budżetowego, jeśli chodzi o 1/12, w budżecie prowizorium nie ma pieniędzy na wynagrodzenia czy też nie ma zagwarantowanych wynagrodzeń w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Pan poseł Ajchler podnosił kwestię samotwórczości albo bardziej pracowników administracji, urzędu centralnego, jakim jest ministerstwo rolnictwa. Panie pośle, chciałbym bardzo wyraźnie zaznaczyć, że w wypadku akurat tej ustawy i praktycznie wszystkich ustaw, które realizują postanowienia Unii Europejskiej i wdrażają prawodawstwo unijne, proporcje są zdecydowanie odwrotne, czyli, jak pan to nazywa, radosna twórczość pracowników ministerstwa to jest 10%, maksymalnie 15% i dotyczy bardzo istotnych rzeczy, jeżeli chodzi akurat o tę ustawę, bo to dotyczy, drodzy państwo, eksportu roślin na rynki trzecie, czyli do krajów innych niż unijne.

Stąd właśnie pojawiają się te przepisy, ale one tylko i wyłącznie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej, gdzie ten aspekt był podnoszony.

Ona w pełni implementuje prawodawstwo unijne.

Wszystkie te uwagi, które były wniesione przez stronę społeczną podczas procedowania nad tą ustawą, jak również nad poprzednią ustawą o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zostały w pełni implementowane do tych przepisów. Dziękuję bardzo. Dziękują serdecznie, panie ministrze. Zapraszam pana posła sprawozdawcę Zbigniewa Dolatę. 15 minut, panie pośle. Wysoka Izbo! Również chciałem podziękować, przede wszystkim panu ministrowi, pracownikom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, panu głównemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa i jego pracownikom, oczywiście również państwu posłom, szczególnie państwu posłom, którzy pracowali w komisji. Była rzeczywiście merytoryczna dyskusja. Mówiłem już o tym, że poprawka opozycji zyskała uznanie. Tak dla jasności trzeba powiedzieć, że pani poseł Niedziela zgłosiła ją, ale ona została złożona przez podmiot trzeci, czyli Unię Owocową, a to świadczy o tym, że... Czujność. Tak. ...posłowie reagują na różnego rodzaju zapotrzebowanie społeczne.

Uważam, że akurat polski rząd, ministerstwo rolnictwa przede wszystkim dba o interes polskich rolników i implementujemy oczywiście przepisy unijne, ale dbamy przede wszystkim o interes Polski, interes polskich rolników, bo do tego, panie pośle, jesteśmy powołani. Dziękuję serdecznie. Panie Pośle! Przed tymi ustawami debatowaliśmy na temat m.in. działów. Niech pan się wczyta w te ustawy. Dojdzie pan do wniosku, że dużo, dużo im brakuje do tego, aby je poprzeć, aby Lewica je mogła poprzeć, bo nijak się mają do jakości pracy wykonanej przez resort rolnictwa. No dobrze. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pracowały przy tej ustawie.

Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie sprawozdania komisji. Pani poseł zmierza w naszą stronę, więc korzystając z dobrych zasad i uśmiechu na twarzy, chwilę poczekamy. Poczekamy jednak chyba na panią poseł Annę Paluch, szanując oczywiście

Proszę państwa, chętnie bym przeszedł do następnego punktu, ale nie ma sprawozdawców do następnego punktu, w związku z czym albo ogłoszę przerwę, a chciałbym chwilę poczekać, albo przepraszając za panią poseł, poczekam na nią jeszcze minutę. Nie, no właśnie nie ma, panie pośle, bo w sposób sprawny, błyskotliwy i inteligentny już bym zarządził następny punkt, ale pomimo swojej sprawności, inteligencji i błyskotliwości nie mogę tego zrobić. Dobre, ale bez zarozumialstwa. Tak że to nie wasz klub. Następny punkt - jestem.

Dzięki uprzejmości posłów sprawozdawców i panów ministrów mamy i tak czas skrócony, w związku z czym. Ale pani poseł, mamy weekend za chwilę, trzeba po prostu być tolerancyjnym, uśmiechniętym. Pokażmy, że potrafimy.

Pani poseł, dzięki sprawności prowadzenia obrad i tolerancji Wysokiej Izby nie straciła pani głowy, bo już mieliśmy zwrócić pani uwagę. Dobrze, proszę pani, ale mam do pani bardzo uprzejmą prośbę. Proszę bardzo.

Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Infrastruktury przedstawiam sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt jest zawarty w druku nr 121, a sprawozdanie Komisji Infrastruktury - w druku nr 156. Pierwsze czytanie projektu zawartego w druku nr 121 odbyło się na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu 15 stycznia tego roku, natomiast szczegółowe prace nad projektem po zakończeniu pierwszego czytania przeprowadziła podkomisja nadzwyczajna, której miałam zaszczyt przewodniczyć. W dniu wczorajszym Komisja Infrastruktury rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji i przyjęła sprawozdanie z druku nr 156, które dzisiaj Wysokiej Izbie przedstawiam. Wysoka Izbo! Zmiany zawarte w omawianym projekcie dotyczą w zakresie obowiązków inwestora takich kwestii jak: procedura uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, zasady sporządzania projektu budowlanego, przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, samowola budowlana, uregulowanie kwestii nielegalnego użytkowania obiektu czy też doprecyzowanie budzących wątpliwości i niejasnych przepisów. Ponadto wprowadzane przepisy służą zwiększeniu bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnieniu sprawności przebiegu procesu inwestycyjnego w zakresie wydawania warunków przyłączania do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych czy kanalizacyjnych, a także realizacji przyłączy do tych sieci. Dzięki nowym przepisom zostaną również uporządkowane kwestie kompetencyjne w zakresie wydawania pozwoleń na budowę obiektów budowlanych związanych z gospodarką morską, a także wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych. Wysoka Izbo! Zmiana druga w tymże art. 1 precyzuje zasady uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Doprecyzowanie tych zasad powinno wpłynąć chociażby na zmniejszenie liczby wniosków, które wymagają uzupełnienia.

Tak że problem jest istotny i warto te przepisy precyzować, żeby tych poprawek było jak najmniej i żeby procedowanie było sprawne.

Nie będzie teraz - jeśli przeprocedujemy ten projekt ustawy i ona zacznie obowiązywać - konieczności uzyskiwania zgody administracji architektoniczno-budowlanej oraz upoważnienia ministra. Zgoda na odstępstwo w zakresie przepisów przeciwpożarowych będzie mogła być udzielona w postanowieniu komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, tak jak obecnie się to dzieje przy wydawaniu zgody na zastosowanie rozwiązań zamiennych na podstawie tegoż właśnie art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wprowadzano bardzo liczne odesłania i wyjątki, co powoduje ogromne problemy z interpretacją tych przepisów. Jak by to powiedzieć, konia z rzędem temu, kto na pierwszy rzut oka rozstrzygnie, jaka procedura go czeka, jeśli chodzi o inwestorów.

Powiem to kolokwialnie: teraz każdy inwestor ma jak kawę na ławę wszystko wyłuszczone w sposób bardzo komunikatywny i jasny. Mianowicie art. 29 ust. 1 zawiera listę przedsięwzięć, których budowa nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30. Przykładowe takie inwestycje to budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce, na której budynek został zaprojektowany, albo budowanie niecek dezynfekcyjnych - przypominam, żeśmy ostatnio to procedowali w związku z walką z ASF; trzeba te niecki dezynfekcyjne w sposób łatwy i skuteczny wykonywać.

Mianowicie te przepisy, które zawarte są w omawianym projekcie, wprowadzają podział projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania działki lub terenu - jest obowiązek wykonywania go na zaklauzulowanym podkładzie geodezyjnym, mapie przyjętej do zasobu - projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. Trzeba podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami na etapie wydawania pozwolenia na budowę przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza się tylko co do zgodności z przepisami projekt zagospodarowania działki lub terenu, natomiast pozostała część projektu budowlanego jest weryfikowana tylko w zakresie kompletności, nie sprawdza się rozwiązań technicznych. Lepiej zatem przedkładać organowi administracji tylko te części projektu budowlanego, które organ weryfikuje, tzn. projekt zagospodarowania działki lub terenu czy projekt architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny jest niezbędny w momencie przystąpienia do wykonywania robót. Proponowane w niniejszej zmianie ustawy zapisy, w szczególności art. 42, który reguluje obowiązki inwestora, mówią jednoznacznie, że przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany zapewnić sporządzenie projektu technicznego i przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, o ile ten projekt jest wymagany - ale to, na podstawie przepisów, w zależności od stopnia skomplikowania zamierzenia budowlanego. Istotne jest również to, że zmniejszeniu z czterech do trzech ulega liczba egzemplarzy projektu budowlanego, który winien być przedłożony organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Wysoka Izbo! Wprowadza się w zmianie 21. przepis, że nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat - oczywiście jeżeli obiekt został wybudowany.

Zmiana 30. z kolei i następne zmiany dotyczą postępowań legalizacyjnych. Wobec licznych wątpliwości i problemów z interpretacją dotychczasowych przepisów zostają one w niniejszej zmianie ujednolicone. Wprowadzane zmiany upraszczają procedurę, wprowadzają czytelne następstwo kolejnych kroków czy etapów postępowania, które podejmuje organ nadzoru budowlanego. Niniejsza zmiana ustawy wprowadza także nowe pojęcie czy nową procedurę: uproszczone postępowania legalizacyjne dla budów zakończonych ponad 20 lat temu. Proszę państwa, legalizacja czy zmniejszenie liczby nielegalnie eksploatowanych budynków leży w publicznym interesie, bo jeżeli obiekt nie jest zalegalizowany, nie podlega przepisom dotyczącym prawidłowego użytkowania, nie ma kontroli technicznych co do utrzymania we właściwym stanie technicznym budynku i narażone jest bezpieczeństwo użytkowników. I ta sytuacja się skończy, jeżeli obiekty zostaną pod pewnymi warunkami zalegalizowane. W celu legalizacji konieczne będzie przedłożenie oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzy technicznej. W tej uproszczonej procedurze organ nie będzie badał zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego. Skoro przez 20 lat lokalny samorząd - a przypominam, że to lokalne samorządy na poziomie gminnym tworzą dokumenty planistyczne, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i inne dokumenty - organ na poziomie gminnym nie podjął żadnych działań, żeby ten obiekt tak czy inaczej zniknął z przestrzeni, to znaczy, że tak powiem, iż lokalne samorządy jakoś się pogodziły z jego wybudowaniem. Powiem nawiasem, że 20-letni okres wystarcza nawet do nabycia prawa własności przez zasiedzenie. Przepraszam, ale.

Proszę nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Uproszczone postępowanie legalizacyjne jednak nie będzie możliwe w każdym wypadku. Jeżeli mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że przed upływem tego 20-letniego okresu zostało wszczęte postępowanie czy, tym bardziej, została wydana decyzja o wstrzymaniu budowy czy rozbiórce, nie będzie można zastosować tej uproszczonej procedury. Proszę państwa, to jest oczywiste, że uproszczona legalizacja, zwłaszcza samowoli budowlanych, wobec których wydano nakaz rozbiórki, byłaby niesprawiedliwa w stosunku do osób, które wykonały np. nakaz rozbiórki konkretnej inwestycji. Dokonano zmian w części dotyczącej wydawania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także realizacji przyłączy do tych sieci. Temu służą m.in. zmiany dokonane w ustawie Prawo energetyczne.

Są one szczegółowo wymienione w odnośniku do tytułu ustawy. Z uwagi na brak czasu nie będę mogła ich tu szczegółowo omówić. W toku prac w podkomisji wprowadzono 13 poprawek merytorycznych. Pierwsze trzy poprawki służą zapewnieniu spójności ustawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ze zmianami dokonywanymi w Prawie budowlanym niniejszą ustawą. Poprawka 4. doprecyzowuje w miejsce dotychczasowego sformułowania „opis konstrukcji” zapis, cytuję, „projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych” w art. 34 w ust. 3, który precyzuje zawartość projektu technicznego. Jest jasne, że nie wystarczy opis konstrukcji, potrzebne są rysunki i niezbędne obliczenia. Poprawka 5. dotyczy wycofania się ze zwalniania inwestorów budynków jednorodzinnych z obowiązku zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót budowlanych, uznając słuszność zastrzeżeń Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, że zwolnienie z tego obowiązku inwestorów budynków jednorodzinnych będzie oznaczało w istocie brak informacji dla organu o osobie, która pełni funkcję kierownika budowy, oraz brak oświadczeń projektanta i sprawdzającego. Przywracamy obowiązek informowania nadzoru budowlanego o rozpoczęciu robót budowalnych przez wyżej wymienionych inwestorów. Poprawka 6. odnosząca się do art. 42 Prawa budowlanego w zmianie 26 prowadzi do wskazania wprost w ustawie przypadków, w których wymagane jest sporządzenie projektu technicznego, tak żeby nie było w tym zakresie żadnych wątpliwości. Art. 42, jak mówiłam, określa obowiązki inwestora. Mówi również jasno, że inwestor jest obowiązany przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny, oczywiście o ile ten projekt jest wymagany, co wynika z innych przepisów. Poprawka 7. odnosi się do już omówionej sprawy uproszczonego postępowania legalizacyjnego, a poprawki od 8. do 13. dostosowują zmiany w innych ustawach do zmian dokonywanych niniejszym projektem w ustawie Prawo budowlane. Wysoka Izbo! Na etapie prac komisyjnych wprowadzono z kolei dwie poprawki merytoryczne. Pierwsza z nich dotyczy zmiany 17. w art. 1 i uwzględnia kryterium zmiany 5% powierzchni zabudowy jako parametru, który określa istotne zmiany projektu, obok już uwzględnionych - wysokości, długości, szerokości oraz liczby kondygnacji. Druga poprawka dodaje nowy przepis przejściowy zgodnie z sugestiami Biura Legislacyjnego, który utrzymuje ważność obowiązujących gminnych dokumentów planistycznych, tzn. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wprowadzono do tekstu projektu szereg poprawek przygotowanych przez Biuro Legislacyjne. Całość projektu (Dzwonek) została przyjęta przez Komisję Infrastruktury 18 głosami za, przy 5 przeciwnych i 3 wstrzymujących. Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Infrastruktury proszę o uchwalenie projektu ustawy o zmianie Dziękuję serdecznie. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Zapraszam uprzejmie pana posła Aleksandra Mrówczyńskiego z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu dotyczące projektowanej ustawy o zmianie Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z druku nr 121. Projekt ten dotyczy, zgodnie z uzasadnieniem, uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego, m.in. wprowadzenia podziału projektu budowlanego na trzy części.

Prawo budowlane wynika z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć. Rozróżnienie elementów projektu budowlanego sprawi, że wydawanie decyzji, pozwolenia na budowę będzie przebiegało sprawniej i szybciej. Dodatkowo projekt ustawy zawiera szereg zmian. Wymienię niektóre z nich. W przepisie właśnie takie wyrażenie powstanie z powodu tego, iż Prawo budowlane winno zajmować się jedynie tą formą zagospodarowania, która dotyczy obiektów budowlanych, a zatem jedynie zabudową. W art. 9 wprowadzono zmiany w zakresie uzyskiwania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych. Zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych nie może być udzielona w ramach prowadzonych postępowań legalizacyjnych. W kontekście wprowadzonych zmian dotyczących podziału projektu budowlanego na części ważne jest podkreślenie faktu, iż w art. 20 ust. 1 pkt 1, który nie jest zmieniony przedmiotową ustawą, odnosi się do projektu budowlanego jako całości. Podstawowym celem w art. 29 proponowanych zmian jest ułatwienie inwestorom ustalenia, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia. W artykule tym wprowadzono katalog obiektów, których budowa wymaga dokonania zgłoszenia. W art. 31 wprowadzono zmiany mające na celu doprecyzowanie kwestii dotyczących zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego. W art. 33 uaktualniono pojęcia dotyczące projektu budowlanego, wynikające z jego nowego podziału, a także zmieniono wymaganą liczbę projektów będących załącznikami do wniosku o wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na budowę z czterech do trzech. Podkreślić należy, że roboty budowlane, w przypadku których wymagane było uzyskanie decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę, mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie projektu budowlanego, w tym projektu technicznego, oraz pod nadzorem kierownika budowy. Projektowany art. 36b ustawy nakłada na kierownika budowy obowiązek udostępnienia organowi nadzoru budowlanego aktualnego projektu technicznego na każde jego żądanie. W art. 53 wydzielono osobny rozdział: Zakończenie budowy, który na celu uporządkowanie przepisów dotyczących tej kwestii. W proponowanej ustawie wprowadzono zmiany w zakresie ustaw: o ochronie ppoż. Prawo energetyczne, o gospodarce nieruchomościami, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków oraz o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt wywiera jednoznacznie pozytywny wpływ na sferę przedsiębiorczości poprzez uproszczenie procedur związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Projekt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej, nie podlega notyfikacji oraz nie wymaga przedstawienia właściwy organom i instytucjom Unii Europejskiej. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość w całości popiera przedłożony projekt ustawy, druk nr 121. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Państwo Ministrowie! Wysoka Izbo! Przedstawiony projekt to kolejny bubel prawny, który będziecie poprawiać wiele razy, jak każdą ustawę z uchwalonych w takim pośpiechu, bo jest on tak niedopracowany. Czemu się tak spieszycie? Przecież inwestycje to nasz rozwój gospodarczy. Nie można wszystkiego niszczyć, rozdając, byleby tylko wygrać wybory. Projekt tej ustawy zakłada m.in. podział projektu budowlanego na trzy części: projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny. Taki podział nie przyspieszy realizacji obiektów. Będzie więcej pozwoleń na budowę, ale mniej oddanych inwestycji. Ale może o to chodzi. Sukces odtrąbiony. Obecnie dyskutuje się w ministerstwach nad wprowadzeniem technologii BIM, czyli Building Information Modeling, gdzie wszyscy branżyści pracują na jednym modelu, więc uzasadnione jest projektowanie kompleksowe, a nie wyłączenie na projekcie architektonicznym, jak zaproponowano w projekcie ustawy. W wielu krajach to już standard. Ta ustawa stoi w sprzeczności z potrzebami takiego nowoczesnego projektowania, mimo że wiele naszych krajowych pracowni już zaczyna tę technologię stosować. Taki projekt według tej nowelizacji będzie miał zatwierdzony plan zagospodarowania, następnie architektoniczno-budowalny, a potem: hulaj dusza, piekła nie ma. A jak nie będzie działać, to nawet nie będzie winnych, bo tą ustawą rozmontowany będzie system kontroli. Od 2021 r. spełnienie norm efektywności energetycznej budynków nie będzie praktycznie możliwe bez odpowiednio zaprojektowanych instalacji budynku, czyli bez projektu technicznego. Czy państwo nie będzie tego weryfikować, wydając wcześniej pozwolenie na budowę? Następna zmiana.

Szanowni Państwo! Problemem procesu budowlanego nie jest czas uzyskania pozwolenia na budowę, bo to maksymalnie 65 dni, ale ilość decyzji, pozwoleń, uzgodnień i zgód. W tym zakresie nic się nie zmienia w tej ustawie.

Wprowadza się też legalizację co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych, i to nawet tych niezgodnych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Kto będzie oceniał te 20 lat? Kto stwierdzi? Nastąpi wysyp zgłoszeń, bo się okaże, że wszystkie nielegalne budowy w Polsce są 20-letnie. Brak jest terminu, do kiedy można to zgłaszać.

Tu chodzi o te najnowsze. Ten pęd do legalizacji to nagradzanie nieuczciwości. Jest to nieetyczne wobec tych, którzy budują uczciwie i zgodnie z prawem. Wprowadzi to chaos przestrzenny w całym kraju, który będzie przynosił negatywne skutki przez dziesięciolecia. W projekcie tej ustawy partykularne interesy wygrywają z dobrem całej wspólnoty, czyli ładem urbanistycznym w naszym kraju, czyli odpowiedzialnością rządu - bo po nas choćby potop. kształtem w niczym nieprzypominające podhalańskiego stylu, które są już legendarnym przykładem polskiej brzydoty, nielegalnej zabudowy, teraz zostaną usankcjonowane na zawsze. To są bardzo duże i skutkogenne zmiany w prawie wprowadzone szybko i chaotycznie z wieloma źle dopracowanymi zapisami, więc klub Koalicji Obywatelskiej składa poprawki, a w przypadku ich odrzucenia - wniosek o odrzucenie ustawy. Dziękuję serdecznie. Pani posłanka Hanna Gill-Piątek, klub parlamentarny Lewica. Zapraszam. Szanowni Państwo! To bardzo duży projekt, który jest bardzo dużą łatką na bardzo bolesne problemy. Tylko łatką niestety, dlatego że te zmiany w Prawie budowlanym, z którymi mamy do czynienia, oczywiście przystosowują to prawo do współczesnych wymagań, oczywiście są potrzebne w wielu miejscach. Pracując w Komisji Infrastruktury i w podkomisji ds. tego projektu, staraliśmy się je ulepszyć jak najbardziej.

Bardzo się cieszę, że to się stało.

Od lat czekamy na kodeks urbanistyczno-budowlany. Prace nad tym projektem zostały przerwane i ostatnie wiadomości z 2018 r. są takie, że nie wiadomo, gdzie ten projekt zniknął.

Miał on m.in. poradzić sobie - ja to przypomnę, bo chciałabym żebyśmy wszyscy o tym pamiętali - m.in. z korupcjogennymi tzw. wuzetkami, z odszkodowaniami, które rabują kasy samorządów, z odszkodowaniami planistycznymi, ze zmorą dobrego sąsiedztwa, z chaotyczną zabudową, z tym, że postępowanie środowiskowe jest oddzielne od normalnego postępowania pozwolenia na budowę. To wszystko miało być, proszę państwa, uregulowane. My, jako Lewica postulujemy, zwracamy się do strony rządzącej i bardzo prosimy o tę reformę planowania i o kompleksowy kodeks urbanistyczno-budowlany.

Tak więc apelując do pana ministra i do całego rządu, bardzo prosimy: podejdźmy do sprawy zarówno budownictwa, jak i planowania kompleksowo. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Jacka Tomczaka z klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Kukiz15.

Wynikająca z konieczności uproszczenia i przyspieszenia procesu legislacyjnego Prawa budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć nowelizacja jest wyczekiwanym ruchem legislacyjnym. Nowela ma na celu doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności projektantów oraz organów administracji, m.in. przez podział projektu budowlanego na projekt w celu zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny. Niektóre elementy projektów będą podlegały weryfikacji przez organy administracji publicznej, z kolei za prawidłowość innych odpowiadać będą wyłącznie projektanci. Powinno to doprowadzić do usprawnienia i przyspieszenia wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę czy też przyjmowania zgłoszeń wraz z projektem. Ponadto przewiduje się, że podział projektu budowlanego spowoduje zmniejszenie obciążeń organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz umożliwi szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z projektowaną regulacją zmieniają się zakresy projektu budowlanego oraz jego poszczególnych części. Konieczne jest również wprowadzenie zmian dostosowawczych do nowej koncepcji projektu budowlanego w innych aktach prawnych. Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że projekt nowelizacji ogranicza nadmierność wymogów dokumentacyjnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę oraz ogranicza koszty konieczne do poniesienia przez inwestorów.

Nowelizacja ma na celu ułatwienie inwestorom ustalenia, jakie roboty budowlane wymagają dokonania zgłoszenia w zamian za uzyskanie pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia. W ustawie stworzono katalog robót budowlanych objętych zwolnieniem z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oparty na obecnych rozwiązaniach w tym zakresie, wprowadzający modyfikacje upraszczające proces inwestycyjno-budowlany. Projekt wprowadza zmiany ułatwiające rozwój automatyzacji usług komunikacyjnych i pocztowych, takich jak biletomaty, wpłatomaty, automaty sprzedające, paczkomaty. Wzmacnia się również pozycja inwestora względem organów administracji publicznej w związku z wprowadzeniem granicznego 5-letniego terminu dla stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Do tej pory nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę można było stwierdzić wiele lat po tym, jak budynek powstał i był użytkowany.

Nie jest on pewnie dziełem doskonałym, natomiast niewątpliwie stanowi pewne ułatwienie dla inwestorów.

Zapraszam pana posła Dobromira Sośnierza z Koła Poselskiego Konfederacja. Witam, Panie Marszałku! Konfederacja z radością wita również wszelkie przejawy chęci liberalizacji, deregulacji, redukcji biurokracji, każdą chęć ulżenia naszym obywatelom błąkającym się w tej dżungli przepisów produkowanych bez litości przez naszą Izbę w ilościach hurtowych. A to właśnie nam ta ustawa obiecuje. Mówimy tutaj o uproszczeniu procedur, o rezygnacji ze zbędnych wymagań. Niestety trzęsiecie się nad tymi zmianami jak kot nad wanną. Odwagi! To może wiele nie dać, bo w biurokracji jak się zetnie jedną głowę, to hydra natychmiast wypuszcza dwie kolejne. Na przykład likwidujemy możliwość uzyskania odstępstwa w procesie legalizacji. Skoro do tej pory można było takie odstępstwo uzyskać i świat się nie zawalił, to cóż by się złego stało, gdyby nadal można je było uzyskać, tylko już w sposób jednolity.

Nie potrzebujemy nadzoru budowlanego w ogóle.

To w ogóle jest cud, że w takim systemie jakiekolwiek budynki powstają i nie walą się na głowę. Jeśli w tym systemie się nie walą, to w żadnym innym też na pewno nie będą się waliły, więc naprawdę, jeszcze raz: odwagi! Dwa kroki do przodu, jeden krok do tyłu. W wielu krajach nie ma nadzoru budowlanego.

Z tych parytetów wynika, że w ciągu całej kadencji Konfederacja będzie miała okrągłe zero miejsc we wszystkich podkomisjach.

Opozycja często tutaj uskarża się właśnie na arogancję, na to, że Prawo i Sprawiedliwość tak bezpardonowo się z nią obchodzi. A więc nie jęczcie nad tym. Sami nie jesteście w niczym lepsi. Konfederacja mimo pewnych zastrzeżeń poprze ten projekt. Dziękuję. Dziękuję, panie pośle, serdecznie. Tak nawiasem mówiąc, nie poczułem się urażony, tylko chciałem się z panem ciepło przywitać, bo lubię pana. Proszę państwa, 12 osób zgłosiło się do zadania pytań. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby się zgłosić? Jeżeli nie, to zamykamy listę. I zapraszam serdecznie pana posła Konrada Frysztaka z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. A jeżeli nie ma, to zapraszam serdecznie pana posła Przemysława Koperskiego z klubu parlamentarnego Lewica. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Natomiast jest wniosek, prośba i zarazem pytanie: Dlaczego projektodawcy nie pokusili się o zmiany daleko idące czy idące głębiej? Właśnie wczoraj zostaliśmy zapoznani przez wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli z raportem dotyczącym nieprawidłowości w działalności powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego. Wynika z niego, że z jednej strony mamy Prawo budowlane, usprawniamy je, ale z drugiej strony nie ma w tej chwili w Polsce instytucji, która byłaby w stanie stać na straży (Dzwonek) tego prawa. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję serdecznie. Zapraszam panią posłankę Katarzynę Kretkowską z klubu parlamentarnego Lewica. Mając minutę do dyspozycji, chciałam poruszyć jedną kwestię szczegółową, drobną, ale istotną, zwłaszcza dla konserwatorów zabytków, którzy ją zgłaszają.

Czyli dach budynku i to, co jest ponad dachem, nie jest traktowane jako kondygnacja. Tymczasem inwestorzy na tych dachach umieszczają szyby windowe, umieszczają klimatyzacje, wentylacje, które szpecą te budynki (Dzwonek), i konserwatorzy. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Chciałam zapytać: Co z polderami, co z zabudową na polderach? Usłyszałam, że reguluje to Prawo wodne, co nie jest zgodne z prawdą. Też tam będziecie legalizować samowole? Bardzo proszę o odpowiedź na te dwa pytania na piśmie. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Wojciecha Saługę, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze!

Powołuję się też na ten raport NIK-u z 19 czerwca zeszłego roku, który powinien być kierownictwu resortu znany, a który pokazuje, że w niektórych obszarach państwa

Mamy zasoby nieadekwatne do potrzeb, mamy środki nieadekwatne do zadań.

Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi zagłębiowskiemu. Lubuskie? Lubuskie. Miło. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Panie Ministrze! Czy inżynierowie budownictwa będą mogli wykonywać projekty zagospodarowania terenu i działki oraz projekt architektoniczno-budowlany? Drugie pytanie. W jaki sposób, usuwając przepisy mówiące o konieczności, o obowiązku dostarczenia opinii odpowiednich instytucji wyznaczonych przez ministra dotyczących bezpieczeństwa obiektów niebezpiecznych, takich jak rafinerie, zakłady chemiczne, elektrownie atomowe chociażby, chcecie państwo zapewnić bezpieczeństwo tych obiektów, jeśli ten przepis wykreślacie? Bo ja rozumiem, że przy dostarczeniu kierownikowi budowy projektu technicznego przez inwestora nikt nie będzie w stanie sprawdzić, czy taka opinia jest czy nie. I po co kierownikowi budowy taka opinia? To musi trafić do odpowiednich instytucji, które stwierdzą, że obiekt taki nie będzie zagrażał bezpieczeństwu. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł. Pani poseł Joanna Fabisiak, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Z dyżurów poselskich - dwa palące problemy, które zgłaszają mieszkańcy, to jest długie oczekiwanie na zgodę na budowę i chaos, i próba budowania byle jak i byle gdzie. Szczególnie ta pierwsza sprawa, wydaje się, może być przez ustawę rozwiązana, ale tylko się wydaje. 3 lata. I teraz czy ustawa rozwiąże ten problem? Myślę, że nie. To, że się zapisze nieco inaczej i nieco inne dokumenty - nie tu jest trudność. Ta sprawa nie jest uregulowana, a urzędnicy domagają się jeszcze jednego i jeszcze jednego, i jeszcze jednego dokumentu, tak długo aż ten okres jest roczny, 2-letni, 3-letni, a potem trzeba zmieniać projekt (Dzwonek) i wszystko zaczyna się od nowa.

Dziękuję. Pani poseł Dorota Niedziela, Koalicja Obywatelska. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!Nie jestem specjalistą od Prawa budowlanego, jednakże biorąc pod uwagę to, że to, co najważniejsze w państwie, to bezpieczeństwo prawa i egzekwowanie obowiązków. Jakżeż to się ma do tego, że ktoś bez pozwolenia wybudował obok nas coś, co nam przeszkadza, i po 20 latach niemożności wyegzekwowania prawa, gdy ktoś bez pozwoleń, bez jakichkolwiek uzgodnień wybudował nam coś w okolicy.

Dziękuję serdecznie. Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska.

Wysoka Izbo!

W chwili obecnej wymaga się stosowania przepisów pożarowych do tych budynków, które powstały 20 lat czy nawet więcej lat temu i zostały oddane do użytkowania. Czy w związku z tą ustawą nie będzie trzeba dostosowywać istniejących obiektów do nowych przepisów? Bo wiąże się to z ogromnymi nakładami finansowymi i przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, np. domy wczasowe, hotele, ponoszą ogromne wydatki na cele remontowe, dostosowując się do tych przepisów.

Dziękuję. Pan poseł Marek Dyduch, klub parlamentarny Lewica. Wysoki Sejmie! Mam ogólne pytanie do przedstawiciela rządu. To już jest kawał czasu. Tamta ustawa, ta początkowa, którą teraz poprawiamy, miała dostosować polskie prawo do nowych warunków rynkowych - samorządy, relacje - bo Prawo budowalne dotyczyło jeszcze czasów Polski socjalistycznej. W związku z tym jest zasadne pytanie, czy po 15 latach zamiast robić tak dużo zmian w tym projekcie, który dzisiaj omawiamy, czy faktycznie rząd nie powinien zaprezentować kompleksowego nowego rozwiązania, tym bardziej że budownictwo w różnych postaciach się bardzo szybko rozwija, chodzi właśnie o Kodeks urbanistyczno-budowlany. Dziękuję. Pan poseł Romuald Ajchler, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo! Prawo budowlane już jest, było, kodeks urbanistyczny także, planowanie kompleksowe także, ale żeby wybudować, to trzeba mieć na czym wybudować. Trzeba mieć grunty, które pozwolą właśnie na tego typu sytuacje.

Kiedyś burmistrz, wójt, prezydent miasta miał bujną wyobraźnię i sobie wymyślił, że tam powstanie jedna obwodnica, a wkoło miasta trzy obwodnice. Zarezerwowano w planie zagospodarowania przestrzennego grunty, blokując jednocześnie prywatną własność.

Dziękuję. Dziękuję, panie pośle. Zapraszam. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Chciałbym, żeby to wybrzmiało z tej mównicy. Panie Ministrze! Dokładna informacja. Czy konieczny jest projekt techniczny, aby inwestor mógł prowadzić roboty budowalne?

Bardzo dziękuję.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Czy są takie plany, ażeby dalej zmieniać Prawo budowlane i zrobić kompleksową nowelizację - taką, która da większy impuls przedsiębiorcom w Polsce i szansę na to, żeby te procedury można było skrócić? Dziękuję bardzo. Pani poseł Jagna Marczułajtis-Walczak, Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Projektowane zmiany to abolicja mająca na celu legalizację bezprawia i działania przeciw ładowi przestrzennemu. To również zmiana, która ma posłużyć odblokowaniu zaśmieconych wnioskami nadzorów budowalnych, bo procedury są trudne, długie i kosztowne. Ale skąd pewność, że uprawnione osoby, które potwierdzą, że budynek jest bezpieczny, zrobią to zgodnie ze sztuką? Przyjmując hipotetycznie, że np. konstruktor potwierdzi, że budynek jest bezpieczny, a potem coś się stanie, to kto za to odpowie? Czy prawdą jest, że samowole budowlane to także pensjonaty, hotele, które nie spełniają norm przeciwpożarowych i innych warunków technicznych? Prawo na dziś jest dziurawe i stąd możliwe jest, że działający hotel czy pensjonat jest de facto samowolą budowlaną. Czy nie lepiej wstrzymać ten projekt do czasu załatania dziur prawnych i wprowadzenia przepisów, które uniemożliwią powstawanie samowoli budowlanych? Jakie rząd planuje wprowadzić zmiany w prawie, aby w przyszłości samowole budowlane nie powstawały? I czy kolejną zmianą proponowaną przez rząd nie będzie np. przeznaczanie terenów zielonych zasypanych gruzem na parkingi? Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Bardzo proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju pana ministra Roberta Nowickiego o zabranie głosu.

Wysoka Izbo! Na wstępie chciałbym podziękować za dotychczasowe głosy w dyskusji, za dotychczasowe prace w komisji i podkomisji. Jak ważny i istotny jest ten projekt, pokazuje ilość przeprowadzonych dyskusji i konsultacji.

Jak słyszeliśmy na posiedzeniu komisji: wręcz przeciwnie - wprowadzenie projektu technicznego powoduje pełną zgodność w BIM. My nie wkraczamy, pani poseł, absolutnie w kwestię BIM.

Tak wiele kontrowersji wywołuje tutaj nowela w zakresie 20 lat i postępowania. Otóż zapominamy o jednej ważnej rzeczy, o bezpieczeństwie. Jeżeli przez 20 lat organ administracji.

I na końcu, jeśli mówimy o gospodarce, to nie zapominajmy o inwestorach, a głos inwestorów jest jednoznaczny w zakresie wprowadzanych nowelą poprawek.

Chcę też poinformować, że jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne - tu chodzi o pytanie o zawieszenie tych prac - to 20 stycznia wznowiono pracę zespołu do spraw opracowania ustawy o planowaniu przestrzennym. Myślę, że tutaj przejdę już do konkretnych pytań panów posłów i pań posłanek, odniosę się do nich w kolejności.

Prawo budowlane to sieć połączeń, to sieć połączeń z innymi ustawami, to wpływ na specustawy, to wpływ na infrastrukturę, to wpływ na jakość życia. Jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z głównym inspektorem nadzoru budowlanego i planujemy szerszą reformę nadzoru budowlanego, tak aby to organy A, B... aby inspektor nadzoru budowlanego mógł efektywnie zarządzać swoim zasobem. My pracujemy nad nowym rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych i przyjrzymy się temu problemowi, bo takie sygnały do nas docierały, te głosy są słyszalne.

Dzisiaj trwały rozmowy z Polskim Związkiem Działkowców. Odrzucam też zarzut o bublu, o trybie pospiesznym. To też jest kwestia - jak mówimy, jak domniemywam, jak rozumiem - jakości pracy inspektorów nadzoru budowlanego. Chcę tylko przypomnieć, że rząd PiS w zeszłym roku wprowadził oczekiwaną od kilku lat podwyżkę dla inspektorów nadzoru budowalnego w wysokości 500 zł na każdą osobę i w tym roku w projekcie ustawy budżetowej jest przewidziane 6% wzrostu od kwoty bazowej. To pokazuje jasno, że reforma legislacyjna idzie w parze z kwestią podnoszenia jakości pracy osób, które pracują w służbach inspektorów nadzoru budowlanego. Odpowiadając na pytanie pani poseł Krystyny Sibińskiej: tak. Jednoznacznie mogę odpowiedzieć: tak. Jeśli chodzi o opinię specjalistyczną, w naszej ocenie. To są sprawy szczególne, które regulują i tak przepisy innych ustaw. Przepisy innych ustaw wymagają zachowania odpowiednich procedur, odpowiednich kryteriów - czy wobec materiału, czy wobec procedury stosowania.

My wręcz wymuszamy przepisami koordynację branżową już na etapie powstawania tych projektów, w zakresie specjalności. To jest ważne. To jest ważne, żeby zachować tę spójność. My to odsuwamy i optymalizujemy proces powstawania tego dzieła, i to jest zgodnie z BIM-em. My mamy to wszystko na uwadze, patrząc i wsłuchując się w ten głos, jak podkreślam, 120 organizacji branżowych. Pani poseł Joanna Fabisiak - kwestia przedłużania wydawania zgody.

My oczywiście monitorujemy tę sytuację i staramy się przeciwdziałać różnym mechanizmom, które powodują opóźnienia, bo tak jak powiedziałem, gospodarka to inwestorzy.

Pani poseł, prawo nie dotyczy poczucia estetyki.

Natomiast te 20 lat. Przypomnę to, co mówiła pani poseł Paluch, pani poseł sprawozdawca, w zakresie tych 20 lat. Przy uchwalaniu na poziomie gminy planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest obowiązek inwentaryzacji samowoli, nielegalnych budowli. Jeżeli gminy tego nie zrobiły bądź nie oddziałują na tyle na tereny sąsiednie, na obszary okoliczne, to znaczy, że dajmy tym osobom możliwość wejścia w system. A co to znaczy: wejście w system? To znaczy: być poddawanym okresowym kontrolom, płacić podatki od nieruchomości. Pani poseł Małgorzata Pępek poruszyła tutaj istotną sprawę, natomiast nie jest to kwestia Prawa budowlanego, ale ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W dialogu z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej my też ten temat analizujemy. Jeśli chodzi o wystąpienie pana posła Romualda Ajchlera, to też nie jest kwestia Prawa budowlanego, panie pośle. Zdaję sobie sprawę i wiem, co pan poseł miał na myśli, natomiast nie ma to związku logicznego z procesem projektowania nowych przepisów. Panie pośle, jeśli chodzi o uwagę czy też pytanie pana posła Mariusza Trepki, to odnośnie do projektu technicznego wymaganego przed rozpoczęciem budowy chcę jednoznacznie powiedzieć, że taki projekt techniczny, czyli komplet dokumentów, będzie wymagany. I tutaj chcę szczególnie pochylić się nad przepisem art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy, jako że on nakłada na inwestora obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - a przypominam, że każdy będzie musiał złożyć takie zawiadomienie o zamierzeniu rozpoczęcia prac budowlanych - oświadczenia projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego dotyczącego zamierzenia budowalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

I kierownik budowy zobowiązany jest w przypadku kontroli organu nadzoru do przedstawienia temu organowi, na jego żądanie, aktualnego projektu technicznego. Proszę państwa, podział jest jednoznaczny i pozytywnie przyjmowany przez inwestorów. Projekt techniczny jest projektem szczegółowym, jest projektem, który wymaga często aktualizacji, którego, jeżeli nie ma istotnych odstępstw, nie ma potrzeby aktualizowania na poziomie organu AAB.

Tak, panie pośle, jak powiedziałem na wstępie, patrząc na kwestię zagospodarowania przestrzennego i kwestię ustawy, bardzo ważnej ustawy, bardzo szeroko dotykającej tych spraw, widzimy, że to nie tylko problem zagospodarowania przestrzennego i tej ustawy, to nie tylko problem planów miejscowych, to problem jakości życia, to problem ochrony pewnych dóbr i tkanek miejskich w systemie architektoniczno-budowlanym. Jeśli mówimy o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym, to niezbędne będą zmiany w Prawie budowlanym. Ostatnie pytanie, pani poseł Jagny Marczułajtis-Walczak.

My to ułatwiliśmy. Panie Marszałku! Wysoka Izba! Dziękuję, panie ministrze.

Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo! Chcę podziękować przedstawicielom klubów Koalicji Polskiej oraz Lewicy za deklaracje poparcia omawianego projektu. Powiem to jeszcze raz. Z całą odpowiedzialnością staraliśmy się w ramach procedowania w podkomisji i w komisji słuchać przedstawicieli strony społecznej, słuchać głosów krytycznych, wyciągać z tego wnioski i próbować tak sprecyzować przepisy, żeby rozstrzygać wątpliwości różnych kręgów, bo przecież interesariusze mają prawo wyrazić swoje zdanie.

Proszę państwa, co do kwestii, że nie wprowadzamy nic istotnego w zakresie zgód i przyśpieszenia procedury, to powiem to jeszcze raz.

A więc, są tu przepisy, które dyscyplinują właściwe podmioty i to powinno wpłynąć w oczywisty sposób na przyspieszenie postępowań. Generalnie dziękuję za dyskusję. Jestem przekonana, że ustawa się przyczyni do tego. Proszę państwa, nie. Planowanie przestrzenne odbywa się na poziomie gminnym i musimy podjąć starania w tym kierunku, żeby jednak kształtować przestrzeń publiczną tak, żeby ona nie raziła oczu. Jeżeli się jedzie do Włoch, to całe Włochy wyglądają jakby spod jednych wytycznych architektonicznych wyszły. Czyli trzeba przedsięwziąć takie działania, które będą wpływały na jakość wspólnej przestrzeni. Z drugiej strony słyszeliśmy, że nie mamy tu ładu urbanistycznego. Trzeba w granicach zdrowego rozsądku zapewnić to, żeby przestrzeń była kształtowana w sposób planowy, spójny, taki, który zapewni nam życie w pięknej przestrzeni, i trudno te wysiłki jak gdyby postponować. Oczywiście wszystko należy robić w granicach zdrowego rozsądku, bo z drugiej strony spotykamy się z zarzutami przedsiębiorców, że nadmierne skomplikowanie procesu przygotowawczego dla inwestycji to są wielkie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Rolą ustawodawcy, odpowiedzialnego ustawodawcy, jest równoważyć te różnorakie głosy płynące z różnych stron i starać się, żeby tak kształtować prawo, by każdy mógł bronić swojego interesu i by zapewnić realizację zadań publicznych w taki sposób, żeby społeczność żyła w jak najlepszych warunkach, a te lepsze warunki to jest również życie w pięknej przestrzeni. Dziękuję, pani poseł. Dziękuję posłom i posłankom. Dziękuję panu ministrowi. Proszę państwa, zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 65 i 165) Bardzo proszę pana posła Leszka Galembę o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 65 i 165. Projekt dotyczy wprowadzenia zmiany polegającej na powierzeniu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zadań w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu, produkcji, przetwarzania i dystrybucji.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła więc poprawki w całości. Wnoszę w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uchwalenie tej ustawy wraz z poprawkami. Dziękuję serdecznie, że zmieścił się pan tak super w czasie, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Panie pośle, proszę bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości mam zaszczyt przedstawić co do projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych stanowisko, które dotyczy wprowadzenia zmiany polegającej na powierzeniu Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zadań z zakresu nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu. Mając na uwadze fakt, iż kompetencje w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych należą do inspekcji jakości handlowej, z czego wyłączony został nadzór w obrocie detalicznym sprawowany przez Inspekcję Handlową, zasadne jest wprowadzenie zmiany polegającej na powierzeniu w całości zadań w zakresie nadzoru nad jakością artykułów rolno-spożywczych jednemu wyspecjalizowanemu organowi urzędowej kontroli żywności. Wobec powyższego uzasadnione jest, aby organ urzędowej kontroli żywności sprawujący nadzór nad jakością produkcji i w obrocie detalicznym podlegał ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych. Z kolei prawidłowe stosowanie materiałów i wyrobów będących w kontakcie z żywnością może mieć wpływ na jakość handlową ofiarowanych z użyciem takich wyrobów i materiałów artykułów rolno-spożywczych, dlatego Inspekcja Handlowa weryfikowała stosowanie się przez przedsiębiorców do wymagań dotyczących materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w zakresie, jaki został wskazany w art. 1 pkt 2. Kontrole w zakresie prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością będą przeprowadzane przez IJHARS wyłącznie w ramach sprawowanego nadzoru nad jakością handlową i nie będą obejmowały aspektów zdrowotnych, nad którymi nadzór sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna. Projektowane skoncentrowanie w ramach jednej inspekcji odpowiedzialności za kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych pozwoli na szybsze reagowanie i wyjaśnianie wątpliwości związanych ze spełnianiem przez podmioty produkujące i wprowadzające wyroby spożywcze do obrotu wymagań z zakresu jakości handlowej. Działanie jednej inspekcji skróci czas niezbędny do zakończenia postępowania kontrolnego oraz wyeliminuje możliwą obecnie ewentualność innej interpretacji przepisów prawnych w związku z kontrolą prowadzoną przez jedną albo drugą służbę kontrolną. Pozwoli to w założeniu na szybsze wycofanie z rynku produktów nieodpowiadających wymaganiom przepisów prawnych, co przyczyni się w konsekwencji do lepszego funkcjonowania przedsiębiorstw i ujednolicenia kryteriów oceny. Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dziękuję serdecznie. Pan poseł Tomasz Lenz z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska ma głos. Proszę bardzo. Panie Marszałku!

Chcę powiedzieć, że jest to dobre rozwiązanie. W modelu obecnym, jaki praktykowany jest w Polsce, nadzór całej drogi, jaką przebywa żywność od produkcji po jej sprzedaż detaliczną, wymaga zaangażowania dwóch instytucji, które różnią się usytuowaniem w obecnej chwili w strukturach administracji rządowej. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych podlega ministrowi rolnictwa, zaś Inspekcja Handlowa prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, co oczywiście wpływa na nie do końca ekonomiczne działania tych instytucji, ale także powoduje, że niedostatecznie bronią one interesów konsumentów.

Dał pan cudowny przykład. Zobaczymy, czy z tego przykładu skorzysta pan poseł Marek Rutka z klubu parlamentarnego Lewicy. Proszę bardzo. Panie Marszałku! Dobroduszny Włodzimierzu! Obawiam się, że nie sądzę. Mam zaszczyt w imieniu Lewicy zaprezentować stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw. Połączenie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z Inspekcją Handlową to na pewno słuszny pomysł i krok w dobrą stronę. Niestety jednak krok ten nie jest wystarczający, ponieważ nie porządkuje całościowo kwestii związanych z kontrolą żywności. Do tego, aby móc powiedzieć, że pod względem zarówno jakości, jak i sprawności funkcjonowania aparatu kontrolnego projekt ustawy reprezentuje spójną wizję, brakuje włączenia do niego Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Warto w tym miejscu powołać się na wyniki raportu Najwyższej Izby Kontroli z dnia 3 stycznia 2019 r. Przypomnę, że to jeszcze przed nastaniem tzw. ery kryształowej w tej instytucji. Ten raport mówił o nadzorze nad stosowaniem dodatków do żywności. Ten raport postuluje utworzenie jednolitej, wyspecjalizowanej służby bezpieczeństwa żywności, kompetentnej w ocenianiu każdego elementu jakości produktu przeznaczonego do spożycia, w tym zarówno jakości zdrowotnej, jak i jakości handlowej.

Obecnie sanepid i WIJHARS pracują w systemie 8-godzinnym od poniedziałku do piątku. Inspekcja nie pracuje w święta i dni wolne.

Bez zgody tej instytucji - to jest bardzo ważne - nie da się dokonywać odprawy celnej towaru spożywczego. Tymczasem na granicy lądowej sanepid i WIJHARS działają w systemie 24-godzinnym. A więc można. Aktualnie - mówię na przykładzie Trójmiasta - brakuje wyspecjalizowanych magazynów celnych, gdzie można dokonywać we właściwych warunkach kontroli towarów wymagających utrzymania np. łańcucha chłodniczego. Jedna doba przekroczenia pobytu kontenera w porcie to jest koszt ok. 150 euro, a trzeba pamiętać, że czasami kontrola trwa 4 doby. Te koszty oczywiście ponosi przedsiębiorca.

Groteskowe są badania prób pobieranych przez WIJHARS. To są pracownicy, którzy nie dysponują odpowiednim zapleczem do przeprowadzenia badań chociażby mikrobiologicznych.

Zacytuję ten raport: Truskawka ma charakterystyczny zapach truskawki, jej kształt jest charakterystyczny dla truskawki. To jest całe badanie, jakie przeprowadziła inspekcja. Nie ma badań dotyczących chociażby obecności metali ciężkich w tych truskawkach wyglądających jak truskawki. Co roku powtarzają się sytuacje, że laboratoria są zamykane, bo skończyły się środki. W ubiegłym roku te środki skończyły się w sierpniu. Przedsiębiorcy są obarczani tymi kosztami badań oraz transportu próbek laboratoryjnych. Zdarza się, że koszt transportu przekracza koszt samego badania. Klub Lewicy od samego początku postawił sobie za cel bycie opozycją konstruktywną, otwartą na dobre rozwiązania bez względu na to, kto jest ich autorem.

Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Koalicja Polska - PSL - Kukiz15 mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, a właściwie stanowiska komisji rolnictwa dotyczącego tej ustawy. Nie ulega wątpliwości, że ustawa była wyczekiwana, jest potrzebna i jest odpowiedzią na potrzeby klientów, tak żeby polscy klienci, idąc do sklepów, mieli pewność, że kupują ten produkt, który jest opisany na opakowaniu. Kierunek dobry. Ważne jest również to, abyśmy zwrócili uwagę nie tylko na administracyjne połączenie tych inspekcji, ale również na ich odpowiednie finansowanie. Jest to bolączka wszystkich inspekcji bez pieniędzy. Nawet najładniej opakowana ustawa, nawet najładniej opakowana inspekcja nie sprawdzi się. To jest coś, co nas niepokoi, ponieważ budżet Inspekcji Handlowej był w UOKiK-u i teraz jest obawa, że połączono dwie inspekcje w ramach budżetu ministra rolnictwa i tych pieniędzy jest niewiele więcej, niż było poprzednio, a zadań przybywa więcej.

Taka ustawa była przygotowana już w 2017 r. Niestety nie została przyjęta i w tej chwili procedujemy nad kawałkiem tej ustawy.

Nie był on niestety procedowany. Jest do wykorzystania. Bardzo prosiłbym o skorzystanie również z tego projektu. Chciałbym podziękować panu ministrowi za wczorajsze posiedzenie komisji, dosyć długie, merytoryczne posiedzenie. Jednocześnie padła tam deklaracja o tym, iż Inspekcja Weterynaryjna będzie wzmocniona, zreorganizowana, że będzie więcej pieniędzy na tę inspekcję. Bardzo się z tego cieszę. Chciałbym przy tej okazji zapytać, kiedy moglibyśmy się spodziewać tego nowego projektu ustawy. Reasumując, ustawa jest dobra, potrzebna. Klub Koalicji Polskiej popiera tę ustawę, czekając na wzmocnienie finansowe tej inspekcji, jak również Inspekcji Weterynaryjnej oraz nasiennej. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Zapraszam pana posła Michała Urbaniaka z koła Konfederacja. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Tutaj mówimy o poprawce do ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i niektórych innych ustaw. Otóż generalnie Konfederacja z uznaniem, a jednocześnie z pewnym zdziwieniem patrzy na dynamiczny rozwój ustawodawstwa w wykonaniu rządu tzw. dobrej zmiany.

Ale już tak bardziej na poważnie, cieszymy się, że rząd też widzi możliwości pewnych usprawnień czy ewentualnie uproszczeń. Otóż dzisiaj zostało tutaj powiedzianych wiele słów bardzo merytorycznych, nie będę ukrywał, na temat samej ustawy, na temat instytucji, które tutaj mają pracować. Natomiast nie wiem, czy zwrócili też państwo uwagę w ogóle na samego obywatela. Przedsiębiorca też jest obywatelem. Tutaj możemy mówić o szerokiej gamie przedsiębiorców czy wytwórców w ogóle. Zatem cieszy nas to, że ktoś stwierdził, że warto, aby ci przedsiębiorcy czy wytwórcy byli kontrolowani tylko przez jedną instytucję, a nie przez szereg instytucji, takich jak UOKiK czy też Inspekcja Handlowa. Wszystko będzie się skupiać w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Generalnie rozumiemy, że przy pewnych uchybieniach czy przy niedostosowaniu się do przepisów kary być powinny, mogą ewentualnie. Zatem postulujemy też o jedną naprawdę niewielką poprawkę. W jednym z artykułów mówi się o przedsiębiorcy, który w poprzednim roku rozliczeniowym nie miał jeszcze dochodów. Ten przedsiębiorca w przypadku uchybień byłby karany kwotą minimum 1000 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu posłowi serdecznie. Bardzo proszę, ustalam czas na zadawanie pytania na 1 minutę. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam takie pytanie dotyczące tego organu kontroli, który ma właściwie kontrolować produkcję żywności od pola do stołu. Prosiłbym, żeby pan minister je trochę rozwiał, a być może i całkowicie.

Pan poseł Wojciech Saługa, Koalicja Obywatelska. Panie Ministrze!

Słyszymy: to jest szkodliwe, to jest szkodliwe, to jest szkodliwe, a jednocześnie jest to dopuszczane do obrotu.

Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jarosław Sachajko, klub parlamentarny PSL-Kukiz15. Wysoka Izbo! Znowu mam pytanie o pieniądze, bo każda inspekcja jest na tyle silna, na ile silni i zadowoleni, i wykształceni są jej pracownicy.

Dziękuję. Serdecznie zapraszam panią poseł Dorotę Niedzielę z Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Chcę powiedzieć, że ta ustawa dotyczy tylko i wyłącznie inspekcji jakości handlowej środków spożywczych. Nie mówimy tutaj o bezpieczeństwie żywności, które jest czymś zupełnie innym, bo w procesie sprawdzania bezpieczeństwa żywności biorą udział cztery inspekcje. PiS mówił nam o tym w dwóch swoich programach wyborczych, że złączy je w jedną wspólną inspekcję bezpieczeństwa żywności.

Wtedy byłaby to jedna inspekcja, która sprawdza wszystko.

A więc proszę nie mieszać pojęć. Dziękuję serdecznie.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Teraz będzie to w jednej instytucji i dlatego możemy czuć się bezpieczniej. Oczywiście tak jak zwrócił uwagę pan poseł Sachajko, pieniądze zawsze są ważne i pieniądze w tym wypadku idą za tą częścią Inspekcji Handlowej, która będzie włączona do inspekcji jakości artykułów rolno-spożywczych. One zostały zapewnione na tyle, na ile jest to możliwe, na tyle, na ile było to przewidziane dla Inspekcji Handlowej. Wszystkie te pieniądze tam idą.

Rzeczywiście ta uwaga. Nie można wprowadzać do obrotu żywności, która ewentualnie miałaby szkodzić. W związku z tym żadna żywność, która jest dopuszczona do obrotu, nie może temu zdrowiu szkodzić.

Nade wszystko, pani marszałek, chciałbym podkreślić, że jest to pierwszy krok w kierunku tego kompleksowego nadzoru, od pola do stołu. Witam też wszystkich państwa po przejęciu przeze mnie prowadzenia obrad. Zapraszam sprawozdawcę komisji pana posła Leszka Galembę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Nikt nie powinien mieć obawy. Ta ustawa przynosi przede wszystkim ulgę przedsiębiorcom, ale również zadowolenie konsumentom, bo ten pierwszy etap połączenia inspekcji, tak jak pan minister tutaj powiedział, dzisiaj dzieje się na naszych oczach. Mówiliśmy, że będziemy łączyć instytucje, i łączymy, i tak się dzieje dzisiaj.

Chcę wszystkim klubom podziękować za merytoryczną pracę i proszę Wysoką Izbę o uchwalenie tej ustawy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm skierował ponownie ten projekt do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 155 i 166) Proszę pana posła Kazimierza Gwiazdowskiego o przedstawienie sprawozdania komisji. Zapraszam, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, zawartego w druku nr 155. Marszałek Sejmu w dniu 9 stycznia 2020 r. skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do pierwszego czytania. Podczas pierwszego czytania zgłoszono trzy poprawki, które komisja przyjęła. Dobrostan zwierząt. Tego rodzaju wsparcie polega na rekompensowaniu rolnikowi kosztów związanych z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów, wykraczających ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Działanie to stanowić będzie zachętę do stosowania nieoptymalnego z ekonomicznego punktu widzenia systemu produkcji, gdyż rolnik stosujący lepsze standardy warunków utrzymywania zwierząt uzyska płatność wyrównującą jego dochód w stosunku do rolnika stosującego standardy podstawowe. Projektowane rozwiązania dotyczące wdrażania działania: Dobrostan zwierząt sprzyjać będą stabilizacji warunków prowadzenia działalności rolniczej, a tym samym pozytywnie wpłyną na konkurencyjność polskich gospodarstw oraz na sytuację finansową polskich rodzin rolniczych. Przez wprowadzenie praktyk mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt zwierzętom zapewni się możliwość realizowania potrzeb behawioralnych, a tym samym - lepsze samopoczucie i zdrowie, co stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania społeczne w zakresie warunków utrzymywania zwierząt. Projektowane przepisy wprowadzają rozwiązania korzystne dla rolników, wobec czego Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2020 r. wnosi: Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Oświadczenie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawi Wysokiej Izbie pan poseł Ryszard Bartosik. Zapraszam. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Wysoki Sejmie! Ten projekt, który jest oczekiwany przez rolników, był zapowiedziany już wcześniej.

Dzięki uruchomieniu tego działania rolnicy będą otrzymywać oczywiście wsparcie finansowe za prowadzenie praktyk związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Zapewni to lepsze warunki utrzymywania zwierząt. Pragnę wspomnieć, że działanie to nie było dotychczas w Polsce realizowane. Wsparcie finansowe będzie udzielane na realizację zobowiązań w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa.

Propozycja wdrożenia działania została zaakceptowana przez Komitet Monitorujący PROW i Radę Ministrów. Projekt zmiany PROW został również zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Do projektu ustawy na posiedzeniu komisji wniesiono trzy poprawki, które dotyczą tytułu ustawy, oświadczeń, które będą składać rolnicy zamiast wniosku o przyznanie płatności, oraz terminu wejścia w życie niektórych zapisów ustawy. Projekt umożliwi wsparcie gospodarstw rolnych.

Daje też szansę małym gospodarstwom na rozwinięcie produkcji. Z drugiej strony jest to szansa na zdrowszą żywność i lepsze utrzymywanie zwierząt w warunkach gospodarskich. Klub Prawa i Sprawiedliwości wnosi o uchwalenie tej ustawy wraz z poprawkami, które zostały złożone w pierwszym czytaniu. Proszę w imieniu mojego klubu o uchwalenie tej ustawy. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam pana posła Kazimierza Plocke do zaprezentowania stanowiska Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska. Proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze!

Programy krowa+ i świnia+ osobiście ogłosił prezes Prawa i Sprawiedliwości pan Jarosław Kaczyński. Dzisiaj mamy dzień prawdy. Przed nami leży projekt ustawy w tej sprawie.

Tylko tyle i aż tyle. Zamiast miliardów złotych rząd proponuje rolnikom 50 mln euro na 2 lata. I nie są to żadne dodatkowe środki, tylko środki przesunięte z innego działania w ramach tego samego programu. Rząd postąpi jak zawsze: zabierze jednym, przekaże drugim. Dzięki temu będzie można powiedzieć: dotrzymujemy obietnic. A my mówimy: sprawdzam. W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że z działania może skorzystać 65 tys. gospodarstw, ale najpierw rolnicy będą musieli wydać 1 tys. zł na przygotowanie wniosku przez wskazanego doradcę rolnego. Te koszty zmniejszą pulę środków na dopłaty dla rolników łącznie o 65 mln zł. W tej sytuacji dla rolników na 2 lata zostanie już tylko 150 mln zł. Według danych rządowych w Polsce mamy 6 mln sztuk bydła i 11 mln świń, w tym 7 mln to chów nakładczy pochodzący z Belgii, Niemiec czy Danii. Rachunek jest prosty.

A prawda jest taka, że biorąc pod uwagę konieczność poniesienia wydatków na przystosowanie obór, chlewni, wliczając 1 tys. zł od projektu dla doradcy, koszty w przyszłości mogą przekroczyć wartość otrzymanej pomocy. Nie ulega wątpliwości, że w ostatecznym rozrachunku rolnicy będą musieli się napracować, aby skorzystać z programów krowa+, świnia+. Na koniec, ten wielki program okazał się zwykłym działaniem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, na dodatek słabo przygotowanym i bardzo słabo dofinansowanym. Ta ustawa pokazuje, z jaką propagandą mamy do czynienia na co dzień.

Warto o tym pamiętać. A wiecie dlaczego? Bo te pieniądze rolnikom się należą. Dziękuję, panie pośle. Stanowisko klubu parlamentarnego Lewica zaprezentuje pan poseł Romuald Ajchler. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Oni o tym doskonale wiedzą. I dzisiaj ten, kto jest związany z polską wsią, wie, że rolnicy mówią: no może coś nam przypadnie.

Ale dostajemy.

I teraz jest pytanie: Co dalej, panie ministrze? Co z nową perspektywą? Czy to jest tylko zachęta dla rolników na wsi, aby może kolejny raz wyciągnęli rękę i zagłosowali za PiS-em? Ja nie komentuję tej kwestii, tylko informuję, że rolnicy jednak swój rozum mają. To jest jedna część tego projektu ustawy. Trzeba włożyć ogromne środki finansowe, żeby przystosować polskie rolnictwo i tych, którzy niedawno oddali do użytku obory, chlewnie z maciorami, do tego, żeby byli w stanie te warunki spełnić.

Ale albo to zrobi i zmniejszy produkcję.

To by groziło rozpowszechnieniem tej choroby, a już o bioasekuracji nie byłoby żadnej mowy.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogłaby w tym uczestniczyć i sfinansować pomoc doradcy, który ma przyjechać do rolnika do gospodarstwa.

Reasumując swoją wypowiedź, panie ministrze, ze względu na to, że te 50 mln trafi na polską wieś. Już kończę, pani marszałek. administratorzy, to znaczy ci, którzy będą szkolenia przeprowadzać etc., cała biurokracja też kilkadziesiąt milionów pochłonie. Dziękuję bardzo, panie pośle. I stanowisko klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Kukiz15. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Maliszewski. Wysoka Izbo! Ta ustawa o PROW, o zmianie systemu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wcale nie jest bardzo oczekiwana przez polskich rolników. To jest taki slogan, którego państwo używacie, argumentując swoje nie do końca dobre pomysły. Dlaczego ona nie jest wcale taka dobra dla polskich rolników?

Ale prawdy w tym nie ma, dlatego że nie wszyscy - tylko i wyłącznie ci, którzy będą te zwierzęta hodować w systemie ekstensywnym.

Państwo wspieracie nie rolnictwo intensywne, takie, które spowoduje wzrost eksportu, tylko państwo tym programem wspieracie rolnictwo ekstensywne, które jest archiwum już dzisiaj w skali europejskiej. Małe rolnictwo nic nie pomoże małemu rolnikowi, dlatego że mały rolnik dzisiaj nie jest w stanie zrealizować zasad bioasekuracji w przypadku zwalczania ASF-u. A w tym programie nie ma nic o wsparciu bioasekuracji, zwalczaniu ASF-u. Ten program jest programem ekstensywnym. Zresztą nie tylko dlatego on jest zły. Bo państwo nie dajecie specjalnych środków budżetowych z budżetu krajowego na ten program krowa+ i świnia+, tylko manipulujecie przy środkach Unii Europejskiej. I myślę, że podstawową przyczyną jest nie realizacja waszego programu wyborczego, chociaż może w części tak, ale przede wszystkim przyspieszenie wydatkowania środków Unii Europejskiej, bo pod tym względem Polska jest na szarym końcu. Jeszcze niedawno było to tylko 29% zakontraktowanych środków w ramach PROW z tej perspektywy finansowej. A teraz: komu zabieracie? Skoro nie dajecie z budżetu krajowego, to komuś zabieracie w ramach PROW. Otóż zabieracie właśnie intensywnym rolnikom, bo zabieracie grupom producentów rolnych, taka była informacja na posiedzeniu komisji. Skoro zabieracie grupom producentów rolnych, to zabieracie intensywnym rolnikom, takim, którzy chcą zainwestować albo zainwestowali po to, żeby wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną na rynku. Bo dzisiaj jak można wzmocnić pozycję rolnika na rynku? Nie słowami, nie tym oczekiwaniem przez polskich rolników. Można to wprowadzić tylko wtedy, kiedy się ich zmusi albo zachęci do wspólnego gospodarowania, żeby na rynku się umieli przeciwstawić dużym odbiorcom. A skoro te środki zabieracie, to, po pierwsze, nic nie zrobiliście w kierunku wzmocnienia polskich rolników na rynku.

Jako dowód kolejny - kolejny wskaźnik. Nie tak dawno, bo w ubiegłym roku, przedstawiliście tutaj projekt ustawy o spółdzielniach rolniczych, który miał z kopyta ruszyć ich powstawanie, organizowanie się rolników w tej rzeczywiście dobrej formie, jaką jest forma spółdzielcza. Chciałbym, żeby tu któryś z ministrów powiedział, ile spółdzielni w oparciu o tę ustawę powstało. Ja mam wiedzę, że żadna. Jeżeli żadna nie powstała, to ten program, który w tej chwili przedstawiacie, jest tak wiarygodny jak Radio Erewań, które mówiło, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają moskwicze. To wszystko była prawda, tylko że nie w Moskwie, a w Leningradzie, nie rozdawali, a kradli, i nie moskwicze, tylko rowery. I wasz program jest dokładnie taki sam. To nie jest program oczekiwany przez rolników, [[Oklaski]] bo zabieracie tym intensywnym rolnikom, a chcecie dać tym, którzy nie mogą sobie na rynku poradzić, i ten program nic im w tym nie pomoże. Gdybyście tym programem wsparli bioasekurację, tobyśmy poparli ten projekt dwoma rękoma. My go i tak poprzemy.

Gdybyśmy nie poparli tego projektu i gdybyście go nie przedstawili, to jestem przekonany, że nie wykorzystalibyśmy środków z Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa. Jeszcze jedna rzecz, która także tu się pojawiła, mianowicie taka - wyraźnie nawet w uzasadnieniu jest to napisane - że aby ten program mógł funkcjonować, jest potrzeba przeszkolenia pracowników doradztwa rolniczego i przeegzaminowania. I znowu mówicie, że to wspiera doradztwo. Gdyby to wspierało doradztwo, to byłoby to zrobione ze środków budżetu krajowego. A wy po prostu z pieniędzy unijnych, nie przeznaczając na doradztwo większych pieniędzy. Wprowadzacie znowu grabież środków unijnych, po to żeby tych pracowników, których powinniście wspierać z własnego budżetu, sfinansować z budżetu Unii Europejskiej. Powiedziałem, że ten projekt poprzemy.

Dziękuję, panie pośle.

Szanowni Panowie Posłowie, Panie Posłanki, Posłannice, Poślice! Nie ma czegoś takiego jak unijne pieniądze. Unia Europejska nie ma maszynki do produkowania pieniędzy, które może później rozdać, tylko Unia Europejska ma te pieniądze, które ciężko pracujący obywatele, w tym ciężko pracujący Polacy, muszą wypracować i wpłacić do Unii Europejskiej. Ale ja chciałbym powiedzieć o rzeczy ważniejszej. Otóż francuski ekonomista Fryderyk Bastiat, francuski ekonomista, pamflecista ekonomiczny, powiedział kiedyś rzecz, wydawałoby się, oczywistą, że są na tym świecie rzeczy, które widać, i rzeczy, których nie widać. W Polsce widać tysiące wielkich, białych tablic, które informują o tym, co powstało dzięki Unii Europejskiej. A czego nie widać? Nie widać tysięcy czerwonych tablic, które powinny stać wszędzie tam, gdzie coś nie powstało przez unijną biurokrację i podatki, którymi zasilamy unijny budżet. Najpierw narzucacie polskiemu rolnikowi, hodowcy idiotyczne przepisy, gąszcz idiotycznych, szkodliwych, niepotrzebnych przepisów, które utrudniają polskiemu rolnikowi pracę, które sprawiają, że koszty pracy polskiego hodowcy są większe, a później przychodzicie, pojawiacie się na białym koniu i łaskawie pochylacie się nad marnym losem rolnika i obsypujecie go złotem. Robicie w ten sposób z siebie łaskawców. Godząc się na system, w którym najpierw Polska wpłaca ogromne pieniądze do Unii, a później polski rolnik musi się starać o odzyskanie tych pieniędzy w ramach projektów unijnych, wniosków o dopłatę, wniosków o finanse unijne - robicie z polskich rolników żebraków. Tymczasem polscy rolnicy nie są żebrakami, a wy nie jesteście łaskawcami, bo jedyne pieniądze, które wy macie, macie dlatego, że zabraliście polskiemu rolnikowi w podatkach. Polska, oddając część budżetu państwa Unii Europejskiej w składkach, oddała w tej części suwerenność, pozwalając Unii decydować, jak te pieniądze zostaną wydane. I kilka dni temu mieliśmy tego strzelisty przykład - zwracam się tu do rządu Prawa i Sprawiedliwości, które narzeka, słusznie, że Unia Europejska wtrąca się w to, jak polski rząd chce zreformować sądownictwo, a kilka dni temu Unia Europejska zapowiedziała, że jak reforma polskiego sądownictwa nie zostanie wstrzymana, to Unia przestanie nam wypłacać odpowiednią ilość pieniędzy. Ale to wy, Prawo i Sprawiedliwość, pozwoliliście Unii na ten szantaż finansowy, podpisując traktat lizboński. To wy ukręciliście na siebie ten bicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie pośle. To może pan, nie wiem, na posiedzeniu klubu czy swojego koła. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mówimy tutaj o 50 mln euro, które zostaną wydane w ciągu 2 lat. Mówimy tutaj o tym, że składki polskich obywateli zostaną ponownie przetransferowane po prostu do rolników. Dziś tak naprawdę jeśli spojrzymy na tę ustawę dotyczącą dobrostanu zwierząt, to możemy powiedzieć jasno, że to jest po prostu ustawa, która jest podkładką dla rządu Prawa i Sprawiedliwości przeciwko środowiskom, które zajmują się ekologizmem, tym ekoterrorystom czy bambinistom, którzy mówią o szeroko pojętym dobrostanie zwierząt, a ten dobrostan już dzisiaj każdy rolnik zapewnia swoim świniom, krowom czy zwierzętom w gospodarstwach.

My się na to nie zgadzamy. Uważamy po prostu, że ta ustawa też jest zwyczajną podkładką. Proszę spojrzeć na to, że rząd buduje tutaj mechanizmy biurokratyczne w przypadku wypłaty każdej dotacji. ARiMR będzie wszystko kontrolował, ARiMR będzie dostarczał doradców -każda dopłata będzie wiązała się z szeregiem kosztów poniesionych szybciej. Jeśli tak mają wyglądać programy świnia plus czy krowa plus, to my na pewno nie będziemy głosować za. Przechodzimy do pytań. Zamykam listę posłów zapisanych do zadania pytania. Wyznaczam czas: 1 minuta.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wiele mądrych słów padło z tej mównicy. Szanowni Państwo! Poseł Maliszewski mówił o grupach producentów rolnych. Czy tak naprawdę w Polsce zależy nam na rozwijaniu towarowych, konkurencyjnych gospodarstw? Chciałbym się zapytać, panie ministrze, gdzie ta obietnica narodowego holdingu spożywczego. Gdzie te podwojone dopłaty, na które czekają polscy rolnicy? Ale naprawdę, szanowni państwo, przede wszystkim powinniśmy patrzeć na to, że powinniśmy wspierać rolnictwo towarowe, rolnictwo, które będzie konkurencyjne w Europie. Kilka miesięcy nie będziemy mogli w ogóle się dowiedzieć, ile osób z tego skorzystało, bo wdrożenie tego programu będzie chyba (Dzwonek) kosztowało więcej niż to, co rolnicy zyskają. Dziękuję bardzo.

215 mln na 6 mln bydła i 11 mln świń. 215 mln zł pomniejszone o 65 mln obsługi.

Natomiast moje pytanie: Czy pan prezes Jarosław Kaczyński wie, że podpisał się pod hasłem krowa+ i świnia+, myśląc o dobrostanie zwierząt?

Duńczycy też dostaną te pieniądze? Pan poseł Tadeusz Tomaszewski, klub Lewica. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Szanowni Przedstawiciele Rządu! W trakcie debaty pojawiła się sprawa niewykorzystania środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Czy to prawda? Na jakim jesteśmy etapie? Czy istnieje zagrożenie niewykorzystania tych środków na wcześniej przyjęte przez polski Sejm programy?

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Wysoka Izbo!

Dobrostan zwierząt jest to bowiem zaspokajanie podstawowych potrzeb zwierząt dotyczących m.in. dostępu do wody, żywienia, higieny, pomieszczeń, w których są zwierzęta chowane. Jeżeli nie będziemy o tym pamiętali, to nie będziemy pamiętali, że z tych zwierząt również korzystamy. Dzięki uruchomieniu takich działań rolnicy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe na prowadzenie praktyk związanych z podwyższeniem dobrostanu zwierząt. Chciałbym zapytać: Jak dzisiaj będzie dokładnie wyglądało finansowanie tego programu z podziałem na województwa, ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego? Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Klimczak, Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Zapraszam. Wysoka Izbo! Szanowni Przedstawiciele Rządu! Chciałbym zapytać, dlaczego państwa projekt nie jest tak jasny i przejrzysty jak wtedy, kiedy prezentowaliście go wiosną tego roku podczas kampanii wyborczej. Proszę jasno i wyraźnie wytłumaczyć polskim rolnikom, dlaczego nie wszyscy, którzy hodują krowy i świnie, będą mogli skorzystać z proponowanej dopłaty. Dlaczego w kampanii wyborczej nie mówiliście, że koszt skorzystania z programu będzie aż tak duży? I nie mówię tylko o opłacie dla eksperta, którą można by załatwić przez ODR przy wsparciu rządowym, ale bardziej chodzi o dostosowanie pomieszczeń tak, aby nie było potrzeby ograniczenia liczebności stada. Bardzo proszę. Będę kontynuował wypowiedź pana posła Tomaszewskiego. Otóż pan poseł Tomaszewski - zresztą w swoim wystąpieniu klubowym również o tym mówiłem - pytał o kontynuację tegoż programu w nowej perspektywie finansowej.

Bo byłoby nieporozumieniem dzisiaj przystosować gospodarstwa, jeśli w nowej perspektywie nie będzie kontynuacji tego programu. Chciałem mieć pewność, z jakich środków to będzie, czy macie państwo gwarancję, że na ten program (Dzwonek) środki będą. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Na pytania szanownych państwa w imieniu rządu odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan minister Ryszard Kamiński. Zapraszam, panie ministrze.

Wysoka Izbo! Dziękuję za wszystkie pytania. Rzeczywiście przy wprowadzaniu nowego działania uzupełniającego dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, co jest, myślę, dosyć naturalne, zadajmy sobie pytanie, jak to będzie realizowane.

Obiecujemy, że ona zostanie przygotowana w najbliższym czasie. Na powtarzające się zresztą pytanie pani Niedzieli o obsługę programu odpowiedzmy tak: szkolenia, bo to wielokrotnie tutaj padało, już od 2 tygodni są prowadzone ze środków ministerstwa rolnictwa, dokładnie centrum doradztwa rolniczego prowadzi już szkolenia i doradcy rolniczy już są przygotowywani. Pieniądze przeznaczone na ten program nie będą zabierane z dotacji dla rolników.

Musimy nad tym pracować. Różnego rodzaju inicjatywy są podejmowane. Natomiast jeżeli te pieniądze miałyby zostać niewykorzystane, to została podjęta taka decyzja, że one lepiej będą służyły podniesieniu dobrostanu.

Konsumenci oczekują wiedzy o tym, w jakich warunkach zwierzęta żyły, były utrzymywane, jak były karmione.

Nie ma regionalizacji, ale jest założenie, że wszyscy, którzy zgłoszą się do tego programu, będą mogli nominalnie z tego skorzystać.

Otóż podstawową sprawą dzisiaj jest to, że rolnicy masowo rezygnują z hodowli w związku z zagrożeniem chorobami, w związku z konkurencją ponadnarodowych koncernów, które stworzyły hodowlę przemysłową w Polsce, i z tym, że opłacalność jednostkowa maleje. W każdej wsi prawie w każdym gospodarstwie są niewykorzystane budynki. Mało tego, codziennie są podejmowane przez rolników decyzje o rezygnacji z hodowli, kolejnych rolników. W związku z tym rolnikom, którzy zastanawiają się, czy ma to jeszcze sens utrzymywać trzodę, czy bydło mleczne czy mięsne, mówimy: jeżeli macie budynki, jakie macie, niewykorzystane, zastanówcie się, policzcie, oceńcie te budynki, często puste już dzisiaj, to, czy w nich nie można by przywrócić czy kontynuować produkcji, bo przecież przy tych waszych budynkach z tą dodatkową płatnością ta kalkulacja produkcji będzie nieco inna. Ja nie mówię, że zwiększymy o 100% opłacalność produkcji, ale na pewno, jak wielu z państwa podkreślało, ta opłacalność relatywnie, szczególnie dla drobnych gospodarstw, wzrośnie.

Pan poseł Ajchler zwracał uwagę na to, zadawał pytanie, czy myślimy o nowym okresie programowania.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Gotowość odpowiedzi na pytanie zgłosił również sprawozdawca komisji pan poseł Kazimierz Gwiazdowski. Bardzo proszę. Ja chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim klubom za merytoryczną dyskusję.

Ta ustawa oczywiście jest skierowana do pewnej grupy, tych, którzy będą w ponadnormatywnych warunkach utrzymywać zwierzęta. Dzisiaj dyskutujemy, że 50 mln euro to jest za mało.

Tak że należy się z tego cieszyć, że kolejna grupa rolników będzie mogła skorzystać z tych rekompensat, z tych środków. Tak że wszystkim dziękuję za merytoryczną dyskusję i proszę o przegłosowanie tej ustawy w Sejmie. Dziękuję bardzo. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 8. porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 38) Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pana Mieczysława Kasprzaka. Pan w roli obywatela, panie pośle. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Nie udało się chyba ze względu na krótki czas, krótki okres, bo pierwsze czytanie tego projektu w ubiegłej kadencji odbyło się w dniu 7 listopada 2018 r., później były wybory i chyba z tego powodu projekt ten nie został przeprocedowany. Dzisiaj przedstawiam go po raz kolejny i dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tę inicjatywę. Tak jak obiecaliśmy wcześniej w Polskim Stronnictwie Ludowym - kiedy nasz projekt został odrzucony, nasz projekt klubowy, inicjatywa obywatelska, bo o to zwrócili się do nas emeryci i renciści - aby ten projekt przeprowadzić, dzisiaj po raz kolejny go przedstawiam. Poparło go ponad 140 tys. emerytów i rencistów, ale nie tylko, bo pod projektem podpisali się również ludzie młodzi. W dniu dzisiejszym sytuacja jest o tyle poważniejsza, jeżeli chodzi o ten projekt, w stosunku do tego, co prezentowałem przy poprzednim pierwszym czytaniu, że sytuacja emerytów i rencistów znacznie się pogorszyła odnośnie do tego, co było półtora roku temu, dlatego też, szanowni państwo, pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na ten temat. Skąd się wziął ten projekt? Otóż rządzący zapomnieli o emerytach i rencistach. Kiedy dostrzegane są wszystkie grupy społeczne, to niestety trzeba stwierdzić, że emeryci i renciści zostali zapomniani. Nie wiem, skąd się to bierze.

Dzisiaj emeryci i renciści stają przed problemem przeżycia następnego miesiąca. Skąd się to bierze? Skąd takie dane? Otóż to jest proste. Wzrasta zadłużenie emerytów i rencistów, i to w trybie bardzo szybkim. Emerytów oczywiście uspokaja się, że będą dodatkowe świadczenia, dodatkowe trzynastki, czternastki, ale jednocześnie zabiera im się co miesiąc z ich przyznanych świadczeń. Później przez cały rok mówi się: wypłacimy wam, przez pół roku, wypłacimy wam trzynastkę, przez kolejne pół roku wypomina im się: a wypłaciliśmy wam trzynastkę, o co macie pretensję, dlaczego domagacie się jeszcze dodatkowych środków? Realna wartość świadczeń emerytalnych spada z roku na rok. Otóż waloryzacja nie zabezpiecza wartości realnej. Mało tego, waloryzacja przychodzi z rocznym albo półtorarocznym opóźnieniem i przykład mamy w tej chwili. Mamy galopującą już inflację, bo tak trzeba przyznać, wzrastają ceny żywności, wzrastają ceny energii, wzrastają ceny usług, ceny leków, i to w galopującym tempie, bo w przypadku żywności w niektórych przypadkach jest to nawet i 20%. Więc pytanie: za co emeryt, rencista mają przeżyć? My proponujemy proste rozwiązanie: uprościć system świadczeń, po prostu nie pobierać podatku, bo emeryci i renciści przez całe swoje życie pracowali, wywiązywali się ze swoich zobowiązań, płacili podatki, wszystkie podatki płacili, nie mieli nawet czasu na wyjazdy zagraniczne, bo w wielu przypadkach nie było takiej możliwości, i dzisiaj państwo nie docenia tego, co zrobili. Budowali Polskę, odbudowywali Polskę, ale kiedy przychodzi do zapłaty w ich dorosłym życiu, to mówi się: no zrobiliście swoje, to my wam rzucimy coś na otarcie łez, rzucimy wam minimum socjalne, rzucimy tę minimalną emeryturę i ratujcie się sami. Dlatego też emeryci i renciści są zawiedzeni tą sytuacją, mówią: dość już oszukiwania nas, oszukiwania naszych rodzin, bo to, co nam obiecano, nie jest realizowane.

Jest tych problemów dość dużo, więc bardzo często rodzi się pytanie, i to pytanie jest zadawane, skąd wziąć na to pieniądze.

Jeżeli płaciliście całe życie, to może w tej chwili nie będziemy już od was pobierać tego podatku. To, co przyznaliśmy wam, to, co jest głoszone na co dzień, że emeryt dostaje 1200 zł, 1300 zł, że to jest prawdą. Bo na dzień dzisiejszy to jest nieprawdą. Bo to jest nieprawdą.

Skąd pieniądze? Dzisiaj słyszymy, że gospodarka rozwija się wspaniale.

się rozwija.

Budżet nam się zrównoważył, nie mamy zadłużenia. Przez tyle lat było źle, bo budżet był. Z drugiej strony emeryci mówią tak: Państwo nie pilnuje tych wydatków, bo na wszystko jest, każdemu się należy. Tym się należało, tym się należało.

O tych aferach słyszymy na co dzień.

Dzisiaj przedsiębiorcy mówią, że jest coraz gorzej, a to właśnie oni są jedynym gwarantem zabezpieczenia dochodów budżetu państwa. Więc zadbajmy o przedsiębiorców, pokażmy, że można rozwijać, a nie zwijać przedsiębiorstwa, to będą pieniądze. I tak moglibyśmy szukać wielu miejsc w naszym życiu codziennym, w naszych budżetach, gdzie znalazłyby się pieniądze. Oczywiście mamy świadomość, że tego nie da się zrealizować w krótkim okresie. Ale przystąpmy do konkretnej dyskusji o sytuacji emerytów i rencistów, bo z dnia na dzień przybywa nam emerytów, którzy żyją na poziomie minimum socjalnego. Te wszystkie dodatkowe świadczenia nie zabezpieczają tego, tak jak powiedziałem. Rozpocznijmy poważną dyskusję nad przyszłością polskich emerytów i rencistów. To dotyczy wszystkich, my w tej ustawie mówimy o wszystkich emerytach i rencistach, całego systemu okołoemerytalnego. W skrócie mówimy: ustawa o emeryturze bez podatku, ale dotyczy to wszystkich, również emerytur rolniczych.

Skorzystajmy z tych rozwiązań, bo oni już od kilkudziesięciu lat mają taki system i to funkcjonuje, i to się sprawdza. To jest system bardzo oszczędny, bo likwiduje pobór podatku, czyli całą tę administrację, i później dodatkowe wydawanie, całą tę promocję, którą robimy. My nie jesteśmy przeciwni i emeryci nie są przeciwni jakimś dodatkowym świadczeniom, one są mile widziane. Ale to jest rozwiązanie systemowe, które daje pewność, że z miesiąca na miesiąc, z roku na rok emerytura będzie w takiej wysokości, jak została przyznana, i tyle emeryt dostanie do kieszeni. Bo emeryt, idąc do sklepu, nie płaci brutto, tylko płaci tym, co dostał do kieszeni, czy tym, co mu przelano do banku i co ma na karcie bankowej. Szanowni Państwo! Wrócę do tego, co spotkało mnie w niedzielę. Otóż pewna emerytka podchodzi od mnie i mówi tak: Panie pośle, zróbcie coś, niech emerytury będą w końcu realne, niech one pozwolą nam na godne życie. Mam siedmioro wnuków i te wnuki przyjdą do mnie z laurkami, przyniosą jakieś małe prezenciki, a mnie nie stać na to, żeby im kupić jakąś czekoladę i podziękować za to.

Mi złotówka nie zostaje, muszę dobrze kombinować i zaciskać pasa, żeby zmieścić się w tej kwocie. I dodaje jeszcze: przecież tych siedmioro wnuków zapracuje na moją emeryturę, bo ja poprzez swoją rodzinę dałam państwu potencjał, który będzie pracował dla Polski, dla obywateli, dla mojej rodziny, i chciałabym, żebym to odczuła. Zróbcie coś w tym zakresie. Dlatego, szanowni państwo, przedstawiając ten projekt w imieniu 140 tys. Polaków, którzy pod nim się podpisali, proszę o skierowanie go do komisji i o dalsze procedowanie nad nim. Jest to projekt obywatelski. Proszę również o to, aby był on w możliwie szybkim terminie rozpatrywany, bo sytuacja jest trudniejsza, niż była wcześniej, kiedy przedstawialiśmy ten projekt, żebyśmy mogli zacząć rzeczowo dyskutować (Dzwonek), bo życie ucieka, czas ucieka, a każdy z nas będzie emerytem, każdy z nas.

Dlatego też, szanowni państwo, my jako Polskie Stronnictwo Ludowe deklarujemy, że nie spoczniemy i że ten projekt wcześniej czy później - taką inicjatywę - przeprowadzimy w Wysokiej Izbie. Panie pośle, przypominam, że pan był przedstawicielem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, a nie klubu Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale dziękuję panu. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Bardzo proszę. Panie Ministrze!

Projekt ustawy, nad którym procedujemy, zakłada zwolnienie emerytów i rencistów z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przypomnę, że składki na ubezpieczenie społeczne, w tym składki emerytalne, są odliczane od wynagrodzenia przed potrąceniem składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Co to oznacza? Oznacza to, że wynagrodzenie przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne jest nieopodatkowane. Po wielu latach składki te wracają do ubezpieczonego w postaci emerytury. Ponieważ dochód ten nie został opodatkowany przy odprowadzaniu składek, podatek jest pobierany przy wypłacie emerytury. Wysoka Izbo!

Polskie Stronnictwo Ludowe, które, odkąd sięgamy pamięcią, uczestniczyło w sprawowaniu władzy, raz z SLD, raz z PO, dzierżyło w swoich rękach odpowiedzialność za system emerytalny, w tym za sytuację emerytów i rencistów, w swoich szeregach miało dwóch ministrów pracy. I wówczas podnieśliście wiek emerytalny. Pytaliście wtedy Polaków? Do kosza wyrzuciliście miliony podpisów. Łataliście dziurę budżetową pieniędzmi z OFE i z wyprzedaży majątku narodowego. Teraz wnioskodawcy wyliczają, że wejście w życie ustawy spowoduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa o blisko 35 mld zł. Źródłem pokrycia tej kwoty według autorów projektu ma być m.in. wzrost dochodów z podatku VAT. Co za hipokryzja. Za waszych rządów z budżetu państwa wyciekło 260 mld zł właśnie z podatku VAT. Wysoka Izbo!

Proponowane zmiany nie przyczynią się do znacznej poprawy sytuacji osób pobierających świadczenia najniższe. Progresywna skala podatkowa powoduje, że najniższe świadczenia wzrosną w znacznie mniejszym stopniu niż świadczenia najwyższe. Zmiany mają negatywny wpływ zarówno na system ubezpieczeń społecznych, jak i na system świadczeń zdrowotnych, wprowadzają negatywne skutki dla systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, negatywnie wpływają na budżet państwa. W opinii Biura Analiz Sejmowych w sprawie zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej, która przecież dla was jest wyrocznią, napisano, że proponowane rozwiązanie jest niezgodne z art. 18 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczącym zakazu dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. Projekt został negatywnie zaopiniowany również przez prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, bo jak napisano, dyskryminacją byłoby przyznawanie zwolnień podatkowych jedynie grupie otrzymującej świadczenia emerytalno-rentowe bez względu na wysokość świadczenia. Co więcej, projekt ustawy może być sprzeczny z art. 84 konstytucji, który stanowi, że każdy jest zobowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków. Prawo i Sprawiedliwość swoimi rządami udowodniło, że w sposób szczególny troszczy się o najsłabszych, o emerytów i rencistów. Dużo można byłoby wymieniać rzeczy, które wprowadziliśmy za naszych rządów.

zaraz podniesiecie wiek emerytalny i każecie im pracować aż do śmierci. Prawo i Sprawiedliwość w odpowiedzialności za cały system emerytalny i w związku z tym, że jest odpowiedzialnym ugrupowaniem, proponuje przesłać ww. projekt do dalszych prac w komisji. Dziękuję bardzo, pani poseł.

A więc zapraszam pana posła Michała Szczerbę, by przedstawił stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska, czyli również w imieniu pana posła Rutnickiego. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Obywatelski projekt ustawy Emerytura bez podatku. Szanowni państwo, czym jest ten projekt? Po pierwsze, jest to zwolnienie z PIT-u na stałe, co miesiąc, bez względu na kaprysy władzy i ich wyborcze kalkulacje, i nie kosztem innych grup, bo największą część osób z niesamodzielnościami, niepełnosprawnością stanowią osoby starsze. Wysoka Izbo! W Koalicji Obywatelskiej inicjatorzy projektu mają swoich sojuszników. Chcemy pracować nad tym projektem w komisjach sejmowych, wypracować najlepsze i najbardziej sprawiedliwe rozwiązania. Wypracowali swoje emerytury. To, czego oczekują od swojego państwa, to przede wszystkim warunki do godnego starzenia się w dobrym zdrowiu. Będzie rokiem drożyzny, ponieważ drożeją koszty pracy, drożeje prąd, drożeje żywność.

Uważamy, że te rozwiązania, które powinny zostać wypracowane, powinny być rozwiązaniami na stałe. Szanowni Państwo! Dochody emerytów w Polsce nie wystarczają na godne życie. Wczoraj otrzymaliśmy dane z Krajowego Rejestru Długów. Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo! Dlaczego takie zadłużenie? Dlaczego polscy emeryci na starość muszą się obawiać komornika, muszą się obawiać windykacji, muszą się obawiać wejścia na ich wypracowane emerytury? Dlatego że w systemie ochrony zdrowia, w systemie publicznym nie uzyskują usług, na które oczekują. Polacy wydają blisko 50 mld zł na prywatne usługi medyczne i leki. To oznacza, że każdy emeryt i każda emerytka 1500 zł rocznie płaci na prywatne wizyty u lekarzy specjalistów, prywatną rehabilitację, prywatne zabiegi i leki, które również kosztują. Leki kosztują również te osoby, które nie mają 75 lat. Dzisiaj jest Dzień Dziadka. Czy Wysoka Izba wie, jaki jest przeciętny wiek życia mężczyzny? To 73 lata. I ten wiek po raz pierwszy od ubiegłego roku się obniża. W zeszłym roku po raz pierwszy od wielu, wielu lat zmniejsza się wiek przeżycia Polek i Polaków. Szanowni Państwo! Kolejna sprawa. Chcemy również reprezentacji osób starszych. Mamy ustawę o osobach starszych, mamy ustawę, która precyzuje, czym są gminne rady seniorów. Stworzyliśmy przedstawicielstwo osób starszych jako Obywatelski Parlament Seniorów, który tutaj zainicjował swoją aktywność w 2015 r. Tego typu formy przedstawicielskiej aktywności, dialogu społecznego nie są przez rząd realizowane. Co więcej, rząd PiS-owski odmawia pracy nad Konwencją ONZ dotyczącą praw osób starszych. To jest, szanowni państwo, niebywałe. Rzecznik praw obywatelskich jest jedynym organem konstytucyjnym, który uczestniczy w pracy nad tą konwencją ONZ. Polski rząd odmawia konsekwentnie tego udziału. Szanowni Państwo! Uważamy również, że trzeba tworzyć zachęty dla osób starszych, które już wchodzą w wiek emerytalny, ale świadomie decydują się, że chcą pracować dłużej. Uważamy, że żeby zachęcać do takiej aktywności, powinno się zwolnić ze składki na ubezpieczenie społeczne te osoby, które kontynuują pracę i nie pobierają emerytury. Wreszcie osoby o ograniczonej samodzielności. Uważamy, że potrzebna jest ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym. Uważamy, że sprawy osób starszych powinny być bardziej zauważane przez rząd. Dziękuję, panie pośle. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Przedstawiciele Komitetu Inicjatywnego! W imieniu klubu parlamentarnego Lewicy pragnę przedstawić stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu ustawy Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ustawy określa w szczególności zwolnienie od podatku dochodowego oraz składki zdrowotnej świadczeń osób pobierających emerytury, w tym emerytury służb mundurowych, rolników, żołnierzy zawodowych, nauczycieli, oraz rent, w tym rent socjalnych. Podstawowym celem przedmiotowego projektu ustawy jest likwidacja obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne. W rezultacie mówimy o grupie 9 mln Polek i Polaków.

Projektodawcy szacują, że spadek wpływów do budżetu państwa będzie równy ok. 15 mld zł, a wpływy ze składek zdrowotnych spadną o ok. 20 mld zł. Od zawiązania się Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej minęły prawie 2 lata. Na pewno podczas prac w komisji należy przejrzeć przepisy zmienione przez emeryturę bez podatku oraz wskazać źródła jej finansowania. W poczuciu sprawiedliwości społecznej i w myśl zasad współżycia społecznego, mając na celu poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów, za konieczne należy uznać wprowadzenie rozwiązań podwyższających otrzymywane przez nich świadczenia.

Projekt ustawy w szczególności zasługuje na uwagę, jeśli chodzi o pochylenie się nad dobrem wspólnym i poziomem życia fundamentalnej grupy społecznej, zwłaszcza że jest to obywatelska inicjatywa ustawodawcza, a zatem reprezentuje ona bezpośredni głos społeczeństwa. Warto zwrócić uwagę na kilka argumentów potwierdzających wagę składanego projektu ustawy. Argument pierwszy: szanowni państwo, gwarancje prawne daje seniorom przede wszystkim Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejska Karta Społeczna. Art. 67 konstytucji stanowi: „Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego”

To efekt tego, że rząd przyjął najniższy z możliwych wskaźników waloryzacji świadczeń. Trzeci argument: obywatele Holandii i Chorwacji po przejściu na emeryturę otrzymują ponad 100% wynagrodzenia. W Polsce 35% ostatniego wynagrodzenia otrzymują mężczyźni, a kobiety - tylko 27%. Jesteśmy na szarym końcu. Argument czwarty: w grudniu 2018 r. prawie 750 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż bycie emerytem. Spośród nich prawie 500 tys. podlegało także ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. W ciągu ostatnich 4 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ok. 30%. Podsumowując, emerytura bez podatku to jeden z ważniejszych postulatów, na których realizację oczekują wszyscy obywatele. Lewica popiera projekty, które poprawiają sytuację materialną emerytów i emerytek, dlatego złożyliśmy projekt zakładający podniesienie emerytury minimalnej do 1600 zł. Projekt ten został odrzucony na wniosek Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy dalej walczyć o godne życie osób starszych, dlatego aktywnie włączymy się w prace nad projektem Emerytura bez podatku na poziomie komisji. Szanowni Państwo! Na koniec pozwolę sobie przypomnieć słowa Magdaleny Samozwaniec, które bardzo pasują do sytuacji: „Starość posiada te same apetyty co młodość, tylko nie te same zęby”

Bardzo proszę. Wysoka Izbo! To jest dla nas bardzo ważny dzień. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich emerytów, rencistów, wszystkich z komitetu ustawodawczego, którzy są też obecni na dzisiejszym posiedzeniu. Pozdrawiam szczególnie UTW z Otwocka, panie, które od lat wspierają tę inicjatywę.

Uważają to za jeden z najważniejszych postulatów, jakie trzeba spełnić w obecnej kadencji. Nie udało się w poprzedniej, ponieważ większość rządząca nie chciała dać wyższych emerytur zwolnionych z podatku wszystkim obywatelom. Fajnie i dobrze, że go poparliście, że jesteście za dalszymi pracami. To jest już pierwszy sygnał. Na to liczą emeryci i renciści. Popiera związek emerytów i rencistów, wielka organizacja skupiająca setki tysięcy emerytów, rencistów i inwalidów z Polski. Popierają związkowcy, np. z OPZZ. Popierają rady seniorów: gminne, powiatowe, wojewódzkie.

Kiedyś wprowadzono podatki, ubruttowiono emeryturę. Tego nie robiliśmy my podczas naszych rządów, tylko robiliście to wy, szanowni państwo z prawej strony sali politycznej, bo rządziliście w Polsce przez 15 lat. Wprowadzaliście OFE, które teraz będziecie likwidować. Chcemy to zmienić. Idziemy za tym wzorem, który dla was powinien być najlepszym przykładem, czyli wzorem budapesztańskim. Inne kraje, kraje nadbałtyckie. Nie przypuszczałem, że będziecie takimi obrońcami Unii Europejskiej.

Będziecie się teraz troszczyć o rzeczy, które można poprawić w komisji, doprecyzować. Naprawdę, dajcie tylko szansę, nie bójcie się. 85% Polaków, nie tylko emerytów i rencistów, ale również emerytów i rencistów, bardziej popiera emeryturę bez podatku niż trzynastą emeryturę. My się cieszymy z każdego wsparcia. My o was potrafimy powiedzieć dobre słowo. Dobrze, że jest wsparcie w postaci trzynastej emerytury. Niedobrze, że nie jest to wsparcie systemowe, że ono nie jest trwałe, tylko zależy od widzimisię, od tego, czy jest rok wyborczy. Bardzo ważne jest, żeby emeryci mieli poczucie bezpieczeństwa. Ceny rosną. Ostatnie dane Eurostatu pokazują, że Polska jest na szóstym miejscu pod względem wzrostu cen towarów i usług. To pokazuje, jak mocno dzisiaj trzeba stanąć po stronie emerytów i rencistów. Nie spoczniemy, dopóki ten projekt nie wejdzie w życie. Zrobimy wszystko, żeby wszedł w życie projekt Emerytura bez podatku, emerytura i renta wyższa dla każdego, dla wszystkich obywateli. Zrealizujemy to. Dziękuję, panie przewodniczący. W imieniu Koła Poselskiego Konfederacja pan poseł Artur Dziambor. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Emerytura bez podatku to jest coś, o czym wspominaliśmy już tutaj podczas jednej z rozmów na temat trzynastej emerytury. Chciałbym tylko przypomnieć, że Konfederacja to jest ta formacja polityczna, która mówi o tym, że nie tylko emerytura powinna być bez podatku, ale też umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, wszelkie zarobki, wszelka działalność. Wszyscy powinni być tak naprawdę odpodatkowani, ponieważ podatek dochodowy docelowo nie powinien istnieć. Proponowaliśmy, żeby rozwiązać to systemowo i po prostu stworzyć stawkę, kwotę wolną od podatku na poziomie dwunastokrotności najniższej krajowej. To tak naprawdę bardzo by odpodatkowało emerytów. O tym też nie było w naszej Izbie dyskusji, ponieważ rozmawialiśmy o propagandowym projekcie trzynastej emerytury, który ma po prostu pomóc kandydatowi partii rządzącej w wyborach prezydenckich. Będziecie ponosili jakieś tam konsekwencje za to, podobnie jak będziecie ponosili konsekwencje za przegłosowanie 2 mld zapomogli dla telewizji, która ma opiekować się propagandą. Natomiast tutaj jest sytuacja, w której można zrobić naprawdę wielki gest dla emerytów i zrobić pierwszy krok ku temu, żeby podatek dochodowy docelowo zlikwidować. Uważamy, że podatek dochodowy jest karą za to, że się pracuje. Uważamy, że podatek dochodowy nie powinien istnieć. Chcielibyśmy o tym poważnej dyskusji. Jeżeli pierwszym krokiem może być odpodatkowanie emerytów, to jesteśmy za, ponieważ uważamy, że takimi krokami należy doprowadzić do tego, żeby system został rozwiązany ostatecznie, tak jak mówimy, całkowicie bez podatku. Konfederacja będzie oczywiście głosowała za tym projektem. Mamy nadzieję, że będzie miał ostatecznie, już po przejściu przez komisję i przez czytania, również poparcie partii rządzącej. To będzie gigantyczny krok dla dobrej zmiany w Polsce. Tak że polecam go gorąco partii rządzącej. Dziękuję bardzo, panie pośle. Przechodzimy do pytań. Do pytań zapisały się 34 osoby.

Zapraszam.

Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Chciałem się dopytać, w jaki sposób i o ile dokładnie wzrośnie ta emerytura, biorąc pod uwagę emeryturę najniższą, średnią i jakąś emeryturę wysoką, kominową. Otóż wiadomo, że jest kwota wolna od podatku.

Czy nie będzie tak, że te niższe kwoty wzrosną minimalnie albo też wcale, natomiast wzrosną wysokie emerytury? Dziękuję bardzo, pani marszałek. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Presja ma sens. Pamiętacie państwo, jak w ubiegłym roku Wysoka Izba przyjmowała to jednorazowe świadczenie, jakim jest trzynasta emerytura. Wówczas ta trzynasta emerytura była opodatkowana.

Czyli Wysoka Izbo, można? Można. Wtedy kiedy jest presja. I druga sprawa, która mnie osobiście, szanowni państwo, zabolała. Jedna z posłanek mówiła, że wprowadzenie zniesienia opodatkowania świadczeń emerytalnych może być niezgodne z konstytucją. Szanowni Państwo! W poprzedniej kadencji dokonaliście zwolnienia z podatku PIT dosyć dużej grupy, a mianowicie osób poniżej 26. roku życia. Można? Można. Nie używajmy dzisiaj argumentów, które nie są merytoryczne. Jeżeli jest dobra wola - a z naszej strony jest taka wola pracy w komisji nad tym projektem - to wszystko jest możliwe. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Jako przedstawicielka Lewicy i jako posłanka osobiście cieszę się z każdego rozwiązania, które miałoby odciążyć Polki i Polaków, sprawić, by żyli godnie i na sprawiedliwych zasadach otrzymywali swoje świadczenia. A moje pytania wynikają z chęci zweryfikowania słuszności jej założeń i efektywności jej działania. Każda ustawa gwarantująca świadczenia socjalne bądź działania prowadzone wokół tych świadczeń, takie jak zwolnienie z podatku emerytur i rent, powinny się osadzać na swoistej sprawiedliwości i ugodzie społecznej. Czy zwolnienie wszystkich emerytów i emerytek, rencistów i rencistek z podatku od dochodu, z płacenia składek zdrowotnych od tych świadczeń spełnia to kryterium społecznej sprawiedliwości? Większość emerytek i emerytów to ludzie ubodzy. Należy zadbać o ich los. Jednak większość to nie wszyscy. Moje pytanie zatem brzmi (Dzwonek): Czy wedle inicjatorów najistotniejszym kryterium zwolnień z podatków i opłat składek jest sytuacja materialna, czy źródło dochodu, od którego należy odprowadzić dane zobowiązania? Dziękuję. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Z dużym zadowoleniem usłyszałem wypowiedzi przedstawicieli wszystkich tych klubów, którzy mówili ciepło o projekcie obywatelskim, ale również to zapewnienie, że nad tym projektem będziemy pracowali w komisji i później, po raz kolejny - mam nadzieję, w Sejmie. Szanowni Państwo! W pierwszej kolejności płaci swoje zobowiązania za mieszkanie, później wykupuje leki, a później zamyka się w swoich czterech ścianach, bo już na więcej go nie stać. Szanowni Państwo!

Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Adamczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Emerytura bez podatku, emerytura i renta bez podatku - to marzenie wszystkich polskich emerytów i rencistów. Ci ludzie przez całe życie płacili podatki, a dziś większość z nich ma głodowe emerytury, zwłaszcza w kontekście spóźnionej i niskiej waloryzacji, drożyzny, wysokich cen prądu, usług, leków, a także niewydolnego systemu zdrowotnego, za co muszą płacić właśnie z emerytur. Uważam, że w poczuciu sprawiedliwości społecznej, szacunku do ich ciężkiej i długiej pracy, emeryci i renciści w Polsce nie powinni płacić podatku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Zabrakło woli politycznej, by zadbać o godne życie tej wykluczonej grupy. Jak najbardziej z tego powodu jest wart poparcia. Ale co z prawie połową polskich emerytów i emerytek, którzy otrzymują świadczenie niższe niż wynagrodzenie minimalne? Świadczenie mężczyzn to średnio 2600, kobiet - 1600, jest to o ponad 60% różnicy. Kiedy wreszcie nasz system emerytalny stanie się systemem sprawiedliwym, opartym na zasadzie solidarności społecznej, gwarantującym wysokość świadczenia, a nie tylko wysokość składki? Co zamierza zrobić rząd, by te świadczenia były wreszcie równe dla kobiet i mężczyzn (Dzwonek) i na poziomie nie niższym niż minimalna pensja?

Zapraszam.

Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Witam również panie emerytki, które przyjechały dzisiaj do nas z Otwocka i nie tylko. Otóż ustawa Emerytura bez podatku jest już po raz kolejny procedowana w Sejmie. Emeryci czekają na wynik tego głosowania. Badania jasno wskazują, że 85% emerytów i rencistów jest za emeryturą bez podatku. Jest za takim rozwiązaniem, jakie proponuje Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe. Ta ustawa budzi wielkie zainteresowanie w środowisku.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Zapraszam. Pani Marszałek! Panie Ministrze!

Pan kandydat na prezydenta Kosiniak-Kamysz pięknie mówi, że to ważny dzień, bo my możemy emerytom przypomnieć, bo jesteśmy przed wyborami prezydenckimi, więc warto coś zaoferować.

Panie Ministrze! Proszę wypunktować i powiedzieć, ile dobrego za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości zostało zrobione dla polskich emerytów po to, żeby godnie żyli, bo to, że żyje im się coraz gorzej, i to, że są tak bardzo zadłużeni, jak powiedział tutaj jeden z posłów, to niestety wynik waszych fatalnych 8-letnich rządów. Pan poseł Mateusz Bochenek, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! Jestem przedstawicielem najmłodszego pokolenia pracującego w parlamencie, pokolenia, dla którego perspektywa emerytury jest niezwykle odległa, niemal trudna do wyobrażenia.

Nie zmienia to jednak faktu, że od najmłodszych lat powinniśmy pamiętać o edukacji, o edukowaniu młodego pokolenia, dlatego tak potrzebna jest zmiana w tym zakresie. Musimy w końcu zacząć myśleć o przyszłości, i to od najmłodszych lat. Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, a niestety dotyczy to tak wielu Polek i Polaków, że emeryt po przepracowaniu 40 lat zastanawia się, czy wystarczy mu pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Pytam zatem Radę Ministrów, pana premiera: Jakie działania zamierza podjąć rząd w zakresie zmiany aktualnej sytuacji i poprawy jakości życia emerytów? Jakie zamierza podjąć działania w zakresie edukacji? Dziękuję bardzo. Przepraszam, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Doceniam to, że skierowane są do Sejmu projekty, które mają poprawić los emerytów. To jest niezwykle istotne.

To by dało emerytom dodatkowe pieniądze. Tak się nie stało.

I zapowiedziany już wcześniej pan poseł Jan Łopata, Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W niejako preambule do tego projektu ustawy czytamy, że w poczuciu sprawiedliwości społecznej, mając na celu poprawę sytuacji finansowej emerytów i rencistów, za konieczne należy uznać wprowadzenie rozwiązań właśnie podwyższających

Tak więc w duchu tej preambuły, którą tutaj przed chwilą przedstawiłem, chciałem zapytać pana ministra o rzecz podobną, też dającą możliwość podwyższenia emerytur.

I w związku z podwójnym ubezpieczeniem istniała również możliwość pobierania świadczeń emerytalnych zarówno z powszechnego, jak i rolniczego systemu, tzw. półtorakrotności tych świadczeń, ale to już jest historia. Mówię o roku urodzenia. otrzymywać połączonych emerytur. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Omawiany projekt ustawy dotyczący zwiększenia rent i emerytur poprzez zwolnienie z obowiązku płacenia podatku przez rencistów i emerytów to rozwiązanie systemowe i zapewniające wzrost tych świadczeń. Dyskusja na temat świadczeń dla starszego pokolenia Polaków w czasie, gdy obchodzimy w Polsce Dzień Babci i Dzień Dziadka - przy okazji składam jak najlepsze życzenia - powinna być kontynuowana. Być może złożony projekt nie jest idealny, ale z pewnością można i trzeba prowadzić nad nim merytoryczną dyskusję. Renty i emerytury muszą wzrosnąć, czego obecnym i przyszłym świadczeniobiorcom życzę. To jest obywatelski projekt ustawy, w związku z czym proszę, abyśmy skierowali go do odpowiedniej komisji i prowadzili dalszą dyskusję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę.

Wysoka Izbo! Pytam posłów PiS: Dlaczego państwa nie ma w tej chwili na sali albo jest was jakaś garstka? Klub Lewicy złożył tydzień temu projekt podwyższenia najniższych emerytur do minimum 1600 zł. Niestety głosami PiS, głosami PSL, Kukiz, a także PO czy KO został ten projekt odrzucony. Dzisiejszy projekt, projekt obywatelski, jest godny tego, ażeby się nad nim pochylić, może wprowadzić poprawki. Prawdą jest, że emeryci całym sercem są za tym projektem.

Dziękuję bardzo. Pan poseł Dariusz Klimczak, klub parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Czy w związku z tym, że obecna ekipa rządząca ma ogromne problemy legislacyjne z wypłatą trzynastej emerytury, która de facto trzynastą emeryturą nie jest, tylko jej minimalną częścią, nie przyszedł najwyższy czas na to, żeby w Polsce zastosować rozwiązania systemowe dotyczące wypłacania emerytur bez podatku? Taki projekt leży.

Czy z tego względu (Dzwonek) nie należałoby ukłonić się Polakom i znieść podatek od rent i emerytur? Pani poseł Ewa Kołodziej, Koalicja Obywatelska. Zapraszam. Wysoka Izbo! W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że obywatelski projekt ustawy zmierza do likwidacji obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenia zdrowotne. To niewątpliwie dobry kierunek i cieszy fakt, że debata o systemowych rozwiązaniach, dobrych dla seniorów, toczy się w naszym parlamencie. W uzasadnieniu projektu czytamy również, że budżet państwa odnotuje zmniejszone wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o ok. 15 mld zł, natomiast wpływy ze składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego będą niższe o ok. 20 mld zł. Wnioskodawcy wskazują jednak, że biorąc pod uwagę zwiększenie świadczeń emerytalno-rentowych, wpływy do budżetu zostaną zwiększone poprzez wzrost dochodów z podatku VAT. Stąd moje pytania: Czy wnioskodawcy posiadają symulację lub analizy, o ile dochody z podatku VAT mogą wzrosnąć?

Pani poseł Wanda Nowicka, klub parlamentarny Lewica. Zapraszam. Nie ma?

Pani Marszałek! Szanowni Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego! Panie Ministrze! Zamiast nieprawdziwe uwagi czy oskarżenia kierować tu, w stronę polityków dzisiejszej opozycji, dobrze, jakby wykorzystała ona ten moment i chociażby przeprosiła polskich rolników za to, że w 2017 r. państwo podnieśliście im emerytury. Podnieśliście wiek emerytalny polskim rolnikom. Mogłaby pani też wykorzystać to jako dobrą okazję i przeprosić za swoich kolegów, którzy byli prominentnymi politykami w czasach AWS-u i wtedy, tak jak to dzisiaj mówiono, ubruttowili emerytury, czyli tak de facto opodatkowali. A pytanie mam do posła wnioskodawcy. Czy prawdą jest, że w najbliższym czasie będziemy mieli do czynienia (Dzwonek) z najwyższą inflacją w ostatnich kilkunastu latach, co przełoży się jeszcze na pogorszenie sytuacji emerytów? Pani poseł Katarzyna Osos, Koalicja Obywatelska. Zapraszam. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Z pewnością wszyscy powinniśmy dążyć do tego, aby zapewnić naszym emerytom, naszym seniorom godne życie. Podczas wielu spotkań z seniorami i rozmów o ich potrzebach, o ich oczekiwaniach postulat zniesienia podatku od emerytury pada najczęściej. Wskazują oni, że jest to rozwiązanie dla nich najkorzystniejsze, że będzie to realne wsparcie, realna pomoc i że przy tym będą to najprostsze rozwiązania. My jesteśmy tutaj, aby słuchać obywateli i wychodzić naprzeciw ich oczekiwaniom. Tak że liczę na to, że podczas prac komisji wszyscy pochylimy się nad tym projektem i wypracujemy najlepsze rozwiązania dla naszych emerytów, ażeby już żaden emeryt nie musiał dokonywać wyboru, czy opłacić czynsz, czy wykupić leki. Mamy wypracować te przepisy z myślą o naszych emerytach. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Środowisko emerytów i rencistów z uznaniem przyjmuje przedłożony projekt ustawy dotyczący emerytur i rent wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie powinno być tak, że emeryci odprowadzają składki przez kilkadziesiąt lat, a później nadal odejmuje się je od zwykle niewielkich świadczeń. Te dodatkowe pieniądze mogłyby pomóc wykupić leki czy opłacić rachunki. Projekt ten został podpisany przez wyborców różnych partii. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy przekazał na moje ręce apel skierowany do parlamentarzystów o podjęcie tej inicjatywy, pisząc, że zniesienie podatku przyczyni się do poprawy sytuacji bytowej wszystkich emerytów i rencistów w Polsce, którzy płacili przez całe swoje życie zawodowe podatki. Dziękuję bardzo.

Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Padło tu wiele oskarżeń pod adresem tych wcześniejszych rządów, które ustanowiły taki czy inny system emerytalny, ale od takich oskarżeń naprawdę emerytura nie wzrośnie i nie znikną problemy związane z systemem emerytalnym, przed którymi właśnie w tej chwili staje ten rząd. I bardzo państwu oczywiście z tego powodu współczuję.

Był to jeden z głównych powodów tego, że w tej chwili emerytury mają jedną z niższych stóp zastąpienia w Europie. To jest po prostu prawdziwy wstyd. Polskie emerytury mają jedną z najniższych stóp zastąpienia, jeżeli chodzi o wynagrodzenie.

Obecnie rządzący deklarowali walkę z ubóstwem w Polsce, troskę o najsłabszych oraz tych najbardziej potrzebujących wsparcia. A walczycie państwo, walczycie i co? Ano nic. Liczba osób zagrożonych ubóstwem w Polsce rośnie i to jest niestety wina rządzących. Coraz większa inflacja, często drastyczne podwyżki cen żywności, usług, prądu, leków najmocniej uderzają w tych, którzy często na przeżycie mają kilkaset złotych miesięcznie, uderzają w polskich emerytów i rencistów. Dlatego apeluję do sumienia rządzących: nie odwracajcie się od nich i w poczuciu solidarności społecznej, odpowiedzialności przyjmijcie ten projekt obywatelski. A do pana ministra kieruję pytanie: Czy zapewni pan polskich emerytów i rencistów, że ten projekt nie ugrzęźnie w komisjach sejmowych, ale zostanie potraktowany równie priorytetowo jak inne projekty, których legislację skracacie nieraz do jednego dnia, do kilku godzin, i przyjmujecie na tym samym lub na następnym posiedzeniu Sejmu? Pytanie to kieruję również do wszystkich posłów partii rządzącej, bo wasze zachowanie w tej sprawie będzie waszym testem na polityczną wiarygodność. Pani poseł Paulina Matysiak, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Jako posłanka Lewicy jestem i zawsze będę po stronie milionów emerytek i emerytów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i społecznej. Nie będzie więc zaskoczeniem, jeśli tak jak inni posłowie Lewicy przypomnę, że to Lewica zgłosiła projekt dotyczący ustalenia minimalnej emerytury na poziomie 1600 zł netto, który niestety podobno opiekuńczy rząd Prawa i Sprawiedliwości bez mrugnięcia okiem odrzucił. Dlatego popieram skierowanie projektu ustawy emerytura bez podatku do prac w komisji, żeby dokładnie oszacować koszty budżetowe tej ulgi i zastanowić się, czy nie powinno się wprowadzić górnego limitu wysokości emerytur zwolnionych z podatku. Dziękuję bardzo. Pani poseł Iwona Maria Kozłowska, Koalicja Obywatelska. Zapraszam, pani poseł. Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Ale to, co proponują nasi polityczni konkurenci, czyli emeryturę bez podatku, uważam za pomysł niesprawiedliwy. Co by oznaczało jej wprowadzenie? To, że ci, którzy mają wysokie świadczenia, np. 4000 zł czy 5000 zł, dostaliby wysoki dodatek, ale ci, którzy mają bardzo niewielkie emerytury, np. 1000 zł czy 1500 zł, prawie nie odczuliby zwolnienia z podatku. Czy sprawiedliwie oznacza, że wszyscy mają otrzymać równą kwotę wolną od podatku, czy sprawiedliwość wymaga, aby regulacja była równa dla wszystkich i dawała równe szanse odpowiednio do wypracowanej emerytury, czy jest to może też propozycja, aby spłaszczyć świadczenia emerytalne? Dzisiaj być może to jest mało istotne pytanie, ale ma jednak fundamentalne znaczenie dla obywateli, którzy w płaceniu składek na ZUS widzą swoją (Dzwonek) przyszłość i zabezpieczenie. Dziękuję bardzo. I pan poseł Krzysztof Gawkowski, klub parlamentarny Lewica. Wysoka Izbo! Projekt emerytur godnościowych, bo tak trzeba mówić o wszystkich projektach, które mają podnieść uposażenie emerytów, powinien być rozpatrywany nie tylko w tym wąskim zakresie dotyczącym zwolnienia z podatku, choć to dobra droga, ale przede wszystkim w zakresie budowy odpowiedzialności za cały system, który umożliwia godne, normalne życie na emeryturze. Lewica zgłosiła projekt ustawy, który miał dać szansę, że godne życie na emeryturze będzie na poziomie minimum 1600 zł. Zwracam się z zapytaniem do pana ministra, ale chciałbym również skierować apel do parlamentarzystek i parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwość.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Gdyby rząd PiS poważnie traktował emerytów, to pieniądze na trzynastą emeryturę byłyby zapisane w projekcie budżetu. Ale nie były. Gdyby rząd PiS traktował poważnie osoby z niepełnosprawnościami, toby nie zabrano z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ich pieniędzy właśnie na wypłatę trzynastej emerytury. A jednak zabrano. Gdyby rząd PiS w poprzedniej kadencji przyjął do prac parlamentarnych projekty ustaw emerytura bez PIT Platformy Obywatelskiej i Emerytura bez podatku PSL, to obywatele nie musieliby zbierać podpisów i składać projektu obywatelskiego. A jednak musieli i zebrali ponad 140 tys. podpisów. Panie Premierze! Zawsze podkreślacie, że słuchacie suwerena. To właśnie ten głos suwerena, na który tak często się powołujecie. Tu i teraz obywatele mówią wam: sprawdzam. Czy rząd PiS wysłucha tym razem suwerena?

Zamrażarka to nie nasza specyfika. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Niewątpliwie emeryci więcej wpłacają do systemu, niż z niego otrzymują. Po pierwsze, jeżeli płacą składkę, ona wchodzi do obrotu funduszu emerytalnego, a każdy obrót pieniądza jest oskładkowany, czyli oprocentowany. Te nie są. One po prostu idą na emerytury tych, którzy dzisiaj są.

Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Dziękuję w imieniu Nowoczesnej za zgłoszenie tego projektu. Ten projekt powinien być przyjęty nie tylko dlatego, że jest poparty przez 140 tys. obywateli, ale też dlatego, że chociaż minimalnie zapewnia uczucie, że obecna władza dba o godność emerytów i rencistów w Polsce. Emeryci od dawna domagają się takich zmian. Największe problemy ze spłatą zobowiązań mają osoby, które dopiero przeszły na emeryturę, a to ta grupa społeczna jest jedną z najbardziej zadłużonych. Ja tylko przypomnę jeden fakt.

Wtedy PiS ten projekt poparł i twierdził, że przecież to państwo odpowiada za sytuację materialną i poziom życia obywateli, tak mówił ówczesny przedstawiciel PiS-u. Dzisiaj mówię: sprawdzam waszą wiarygodność. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! To bardzo ważny z punktu widzenia społecznego projekt, który daje nadzieję na poprawę sytuacji materialnej emerytów i rencistów, w szczególności tych, którzy są w trudnej sytuacji, mają niskie świadczenia, często prowadzą jednoosobowe gospodarstwo rodzinne. Sojusz Lewicy Demokratycznej, klub Lewicy zgłosił ten projekt dotyczący podwyższenia minimalnej emerytury do 1600 zł, ale mamy w naszym programie także projekt dotyczący emerytury wdowiej, czyli części po zmarłym małżonku. To jest również bardzo istotne, bo jak wspomniałem, ta bieda dotyka często pozostających samotnych emerytów i rencistów.

Dziękuję. Pan poseł Jakub Rutnicki, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Cytując klasyka, zapytam, czy ten projekt emerytom się należy. Tak, oczywiście, że się należy.

To jest m.in. wasza wina, szanowni państwo, dlatego że szaleje inflacja, szaleje drożyzna. Wzrost cen leków, wzrost cen artykułów spożywczych, wzrost czynszu. Pani poseł mówiła o dotrzymywaniu słowa. A kto obiecał, a kto zapewniał wszystkich Polaków, przede wszystkim emerytów, że ceny prądu nie wzrosną? Z tej mównicy mówił to premier Morawiecki. Potem powtarzał to minister Sasin, że ceny nie wzrosną. A co się stało? Wzrosły, szanowni państwo. Dlatego trzeba konkretnych rozwiązań systemowych. Ten projekt ustawy (Dzwonek) emerytom po prostu się należy. Dziękuję. Pan poseł Dariusz Wieczorek, klub parlamentarny Lewica. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Rzeczywiście to jest projekt ustawy, o którym możemy jako Lewica powiedzieć: jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Rzeczywiście nasz projekt ustawy przepadł w komisji.

Pani poseł Monika Rosa, Koalicja Obywatelska. Bardzo proszę. Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Czy konieczne jest zwiększenie wysokości rent i emerytur dla Polek i Polaków? Tak, jest konieczne z wielu powodów, dlatego mam pytanie do posła wnioskodawcy: Czy prawdą jest, że to renciści i emeryci są w Polsce jedną z najbardziej zadłużonych grup społecznych? Jakie są powody tego zadłużenia? Czy prawdą jest, że powody są bardzo prozaiczne? Po pierwsze, te długi wynikają z konieczności wykupienia leków, na których ich nie stać. Po drugie, z konieczności szukania prywatnej pomocy specjalistycznej u lekarzy, która nie jest dostępna ze względu na fatalny stan geriatrii w Polsce. Po trzecie, ze względu na poszukiwanie prywatnej rehabilitacji, która w Polsce jest bardzo słabo dostępna. I to są rzeczy najważniejsze, ale mamy także szalejącą drożyznę, wzrosty cen prądu, wzrosty cen kolejnych usług.

Pan poseł Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kraj mój widzę dostatni, a ludzi - żyjących szczęśliwie. Te słowa powinny przyświecać wszystkim posłom, a szczególnie posłom opcji rządzącej, i każdą chwilę spędzoną w tym parlamencie powinniśmy wykorzystywać do tego, żeby mówić opcji rządzącej, że emeryci i ludzie niepełnosprawni to są dwie grupy, które są najsłabsze społecznie, są niedofinansowane i potrzebują pomocy państwa. Państwo, które nie dba o swoich emerytów, państwo, które nie dba o ludzi niepełnosprawnych, właściwie nie powinno przybierać miana państwa. To jest jakieś konsorcjum dla swoich, konsorcjum dla klientów, konsorcjum dla bogatych.

Pani poseł Małgorzata Chmiel, Koalicja Obywatelska. Wysoka Izbo! W Polsce mamy ok. 9 mln emerytów i rencistów. Dochody emerytów w Polsce nie są wystarczające na godne życie, wzrastają ceny usług, żywności, brakuje na leki. Chciałam się zapytać, czy rząd, zamiast wypłacać kolejne trzynaste emerytury tuż przed kolejnymi wyborami, po to, żeby przekupić, nie mógł zwolnić emerytów z podatku? Szanowni Państwo! To jest nasz podstawowy obowiązek, żeby dbać o emerytów. Im naprawdę jest ciężko, a to pozwoli zaoszczędzić minimum 300 zł od jednej emerytury. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Obowiązkiem każdego obywatela, zwłaszcza w sile wieku, jest wspieranie osób słabszych, w szczególności dotyczy to osób potrzebujących: dzieci, ale także emerytów. To jest projekt, który daje godność życia emerytom. Tak często państwo powołujecie się - mówię o partii rządzącej - na emerytów, to dla was dzisiaj jest naprawdę wielki sprawdzian. Emeryci nie mogą czekać na wybory, emeryci nie mogą czekać na czyjąś łaskę, czy rząd będzie łaskawy, czy da trzynastkę czy nie. To im się po prostu należy. Proszę państwa, ostatnia rzecz: wszyscy wiemy, że ceny rosną, emeryci wydają coraz więcej środków finansowych na leki, zatem niech to będzie nasze wspólne dzieło. Wszyscy poprzyjmy ten projekt. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, mówienie o emerytach to nie jest tylko kwestia pustych deklaracji i twierdzenia, że trzeba coś zrobić, że my stawiamy na emerytów, że potrzebna jest dla nich opieka czy inne wsparcie. Trzeba w tych sprawach bardzo konkretnie działać, rzeczywiście trzeba podjąć takie działania, które w realny sposób dadzą wsparcie emerytom, zwłaszcza tym, którzy mają najgorzej, którzy są na poziomie poniżej wszelkich standardów życia, przeżycia, nie mówiąc już o godnym życiu. Dlatego też nie będę pytała, ale chciałabym bardzo serdecznie zaapelować do strony rządowej, żeby ten projekt poparła, żeby przychyliła się do założeń tego projektu, bo trzeba skończyć mówić, trzeba zacząć działać, i to jest właśnie ten moment. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos w trybie sprostowania poprosiła również pani poseł Urszula Rusecka. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Sprawozdawcą tej ustawy, przypomnę, który wykonał całą czarną robotę, był wasz przewodniczący prezes Kosiniak-Kamysz. Bardzo dobrze, że pani poseł, pani posłanka mówi o tym, że sprawy emerytów są bardzo ważne, trzeba do nich podejść systemowo.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. W pierwszej kolejności na pytania odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pan minister Stanisław Szwed. Zapraszam, panie ministrze. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Tu jeden z panów posłów zarzucał któremuś tam z rządów, który wprowadzał te zmiany.

To jest pierwsza rzecz. Mogę tutaj jeszcze kilka przykładów podać, ale to taki chyba bardzo ważny przykład, bo on dotyczy 9800 tys. emerytów, którzy są uprawnieni do świadczeń. Mówimy o najniższym świadczeniu. Najniższa emerytura. No to przypomnijmy sobie rok 2015, ile wynosiła najniższa emerytura - 880 zł. Wzrost najniższej emerytury o prawie 37%. To jest realny wzrost świadczeń, jeśli chodzi o najniższą emeryturę.

W tym roku będzie kwota gwarantowana minimum 70 zł.

Zmiana zasad waloryzacji, która będzie również obowiązywała w tym roku, czyli waloryzacja kwoto-procentowa. Najniższa wysokość waloryzacji - 70 zł.

Do tego trzynasta emerytura, która będzie dotyczyła wszystkich uprawnionych emerytów i rencistów, czyli 9800 tys. uprawnionych. A więc łączne środki, które będą w tym roku przeznaczone na wsparcie dla emerytów w tym zakresie, czyli trzynasta emerytura, waloryzacja, to jest prawie 22 mld zł. Jeśli chodzi o inne rozwiązania, zastosowaliśmy w ubiegłym roku po raz pierwszy emeryturę 4+, czyli świadczenie dla tych mam, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci i nie miały uprawnień do żadnego świadczenia bądź miały uprawnienia wynikające z mniejszego stażu emerytalnego.

Tego świadczenia nie było. Z tego mogą korzystać, jak powiedziałem, mamy, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci - oczywiście ojcowie też, jeżeli mamy już w tym przypadku nie ma. Nie ma lepszej metody, żeby wspierać tych, którzy mają najniższe dochody, jak podnoszenie kwoty wolnej od podatku.

Państwo mówicie o sprawiedliwości społecznej. No już tutaj widzę, że po stronie Lewicy jest jakaś chwila refleksji. To państwu podam przykłady, jak wygląda sprawiedliwość społeczna w tym projekcie. Emerytura brutto - 1200 zł, zysk z podatku - 175 zł. Emerytura w wysokości 5 tys., podatek - 868 zł.

Jeżeli państwo mówicie o sprawiedliwości społecznej, to tej sprawiedliwości społecznej w tym projekcie akurat nie ma. Szukajmy innych rozwiązań, a nie w tym systemie. To jest jakby ta najważniejsza rzecz, która wynika z tego projektu.

Jeżeli chcemy wspierać, tak jak wspieramy przez nasze projekty - czy to zmiana zasad waloryzacji, czy jednorazowe świadczenie, czy za kilka tygodni będzie przedstawiony projekt czternastej emerytury, który też będzie wychodził naprzeciw dodatkowym środkom dla emerytów - to szukajmy w takich rozwiązaniach, bo to rozwiązanie nie jest rozwiązaniem systemowym. Ono powoduje, że jeszcze bardziej zwiększamy różnicę między najbogatszymi emerytami a tymi najsłabszymi, zwalniając z tej kwoty.

Tu oczywiście pan poseł pytał o emerytury rolnicze. Po zmianie systemu emerytury rolniczej, jeżeli ktoś ma wypracowane 25 lat, mówię o mężczyznach, to ma emeryturę rolniczą, plus te, które ma wypracowane w systemie powszechnym, ale już nie ma tego liczenia, zostało to zmienione w 1998 r. Dzisiaj jest dokładane do tego za ten okres to.

Ten projekt nie jest sprawiedliwy społecznie i w takim kształcie, w jakim jest zaprezentowany, trudny jest do zaakceptowania. Jest decyzja dotycząca skierowania projektu do prac w komisji i również w tej komisji będziemy nad tym projektem pracować. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Zapraszam do zabrania głosu przedstawiciela komitetu inicjatywy obywatelskiej pana Mieczysława Kasprzaka. Tylko, panie pośle, proszę nie mylić znowu roli. Komitet inicjatywy obywatelskiej. Bardzo proszę. Pani marszałek, ja jestem z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To, że przygotowaliśmy ten projekt i on jest praktycznie identyczny z tym, co państwo odrzuciliście, to zasługa tych państwa, którzy tam siedzą i popierają to rozwiązanie. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za podjęcie tematu i taką rzeczową dyskusję, która pokazuje rzeczywiście, jak trudno żyje się dzisiaj emerytom. Bo rzecz nie w tym, że wprowadziliśmy jakieś rozwiązania, że staramy się, tylko sytuacja z dnia na dzień, z roku na rok staje się coraz gorsza. Spróbuję odnieść się do kilku rzeczy, omówię je mniej więcej tak, jak tutaj pojawiały się te pytania i ta dyskusja. Poczucie sprawiedliwości. No właśnie emeryci oczekują tego poczucia sprawiedliwości i podatek jest tym elementem. Tak, płaciłem całe życie, chodziłem do pracy, nie chodziłem na chorobowe, nigdzie nie wyjeżdżałem, pracowałem od świtu do nocy i teraz jeszcze muszę płacić podatek.

Składka emerytalna w jakimś sensie też jest tym podatkiem, bo ona trafia do ZUS-u czy do budżetu państwa. Myśmy przewidzieli, że samorządom zrekompensujemy ten ubytek, nie tak jak jest przy wszystkich innych ustawach, gdzie likwiduje się obciążenia podatkowe, ale zapomina się o samorządach i one tracą. Dzisiaj mamy efekt tego, że w wielu przypadkach obniżono podatek, obniżono PIT, ale nie zrekompensowano samorządom.

Myśmy tutaj to przewidzieli. Ona wtedy, gdy projekt był tworzony, była mniej więcej w tej wysokości, w tej chwili jest wyższa.

To jest do rozpatrzenia, dopracowania w trakcie prac w komisji. Oczywiście projekt jest niedoskonały, bo na etapie tworzenia tak trudnego projektu, bo to jest projekt systemowy, on obejmuje wszystkich. System emerytalny w Polsce nie jest prosty, jest rozwarstwienie, to się zgadza. Z tym że ja bym tutaj nie demonizował, bo od pewnego czasu zaczęło się takie napuszczanie, a ci biedni emeryci to oni dostaną coś tam, natomiast ci tam, którzy mają po 5 tys., to zagarną całą pulę. Nie, nieprawda.

Jednak to nie jest tak, że akurat ci najbogatsi zagarną, jak to się mówi, całą pulę tych środków, które przeznaczymy na obniżkę podatków od świadczeń emerytalnych, natomiast biedni, ci seniorzy, którzy mają niższe świadczenia, na tym nie skorzystają.

Te składki były wyższe. Naprawdę dzisiaj emerytom i rencistom żyje się coraz trudniej. Coraz trudniej. Nie mieliśmy.

No tak, tylko że w tamtym czasie nie było inflacji, tylko była deflacja. Deflacja. A w tej chwili mamy do czynienia już z galopującą inflacją. No galopującą, bo jeżeli ceny śmieci rosną o 60%. Rosną? Kto za to zapłaci? Obywatel za to płaci. Ceny prądu rosną. A ceny usług rosną? Rosną, bo te ceny prądu przekładają się na ceny wszystkich świadczeń.

Emeryt kupuje tę żywność. 1200 zł to jest minimum socjalne.

Czyli brakuje tych pieniędzy. Zmniejsza się wysokość świadczenia emerytalnego. Wszyscy o tym wiedzą i wszyscy o tym mówią: z roku na rok. Za kilkanaście czy za 20 lat to będzie drastycznie niski poziom.

Kiedy ubóstwo będzie na poziomie kilkudziesięciu procent?

Ale rolnicy czekają. Nie mają pretensji, że ktoś więcej uzyska na zwolnieniu od podatku, bo to też jest określony gest w kierunku rolników.

Proszę mi pokazać jedną kobietę, która by przeszła na emeryturę w takim wieku. Nie było takiego przypadku.

Podwyższyliście?

Najdłuższe urlopy macierzyńskie w Europie, [[Oklaski]] najdłuższe urlopy macierzyńskie. Były osoby, które nie miały żadnego prawa do zasiłku macierzyńskiego.

My się od tego nie odcinamy, tylko nie róbcie z tego polityki partyjnej, bo wy robicie politykę partyjną. Jak wam trzeba głosów do wyborów, to będziecie przez pół roku mówić: damy trzynastkę, a później przez pół roku: daliśmy wam wszystko. Po co robić takie szopki? Wprowadzić systemowe rozwiązanie, znieść podatek od emerytów i rencistów, to byłoby prostsze. Nie musielibyście jeździć autobusami, busami, krzyczeć: emerytura, trzynasta emerytura.

Pochylmy się nad tym naprawdę i przemyślmy to do końca, jakie oszczędności z tego tytuły by były.

Kupią sobie żywność, pokryją wydatki, zadłużenia, które mają.

W dużej części trafią do budżetu.

Nie będzie tak, że trzeba wyciągnąć gotóweczkę, gotowe środki z budżetu, żeby dać emerytom. Szanowni Państwo! Dziękując za tę rzetelną i uczciwą dyskusję, bo uważam, że ona była uczciwa, wszyscy pochylili się nad tym. Dzisiaj nie oglądajmy się, co było 20 lat temu ani kto to wprowadził 20 lat temu. Dzisiaj żyjemy w cywilizowanym świecie, gdzie należy pochylić się nad emerytami. Może kiedyś była trudniejsza sytuacja.

To nie jest, jak zaznaczyłem w pierwszym wystąpieniu, idealne rozwiązanie, które załatwi problem wysokości świadczeń dla emerytów. Trzeba szukać innych rozwiązań. My też jesteśmy otwarci i też będziemy zgłaszać inne propozycje. My będziemy popierać te propozycje, naprawdę będziemy popierać te propozycje. 500+, którym się chwalicie na okrągło - przecież myśmy to popierali, przecież myśmy wcześniej też mówili o trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o rodziny, rodziny wielodzietne. Wracam jeszcze do jednego tematu. Ono do końca też nie jest sprawiedliwe, bo do mnie przychodzą panie i mówią tak: wychowałam piątkę dzieci i praktycznie ani dnia nie byłam na urlopie wychowawczym, pracowałam, ratowałam się jak można i mam takie samo świadczenie jak kobieta, która nie przepracowała może w ogóle ani jednego dnia. Więc też trzeba by się zastanowić, czy to jest sprawiedliwe, czy to jest uczciwe.

Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, proponuje, aby Sejm skierował obywatelski projekt ustawy Emerytura bez podatku oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawarty w druku nr 38, do Komisji Finansów Publicznych oraz do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu rozpatrzenia. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (druki nr 128 i 168) Proszę pana posła Jerzego Polaczka o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z satysfakcją pragnę przedłożyć Wysokiej Izbie sprawozdanie odnośnie do rządowego projektu zmiany ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, który jest zawarty w druku nr 128.

Po pierwsze, sam model wsparcia funkcjonuje od ok. 10 lat. Warto odnotować, że w tym czasie łączne nakłady ze strony budżetu państwa na wsparcie tych zadań przekroczyły sumę 527 mln zł, natomiast łączna wartość inwestycji odnoszących się do termomodernizacji i remontów przekroczyła 3 mld 300 zł.

Po pierwsze, jest to zwiększenie efektów programu wspierania termomodernizacji i remontów poprzez objęcie wsparciem kolejnych celów, takich jak remonty budynków, tak jak powiedziałem wcześniej, z wielkiej płyty oraz remonty budynków komunalnych. Te podstawowe rozwiązania, które zawiera sam projekt, w szczególności dotyczą dodatkowego wsparcia dla właścicieli i zarządców budynków z wielkiej płyty na wykonanie dodatkowych połączeń między warstwą nośną a warstwą fakturową ścian zewnętrznych. Według proponowanej przez rząd regulacji premia będzie wynosiła 50% kosztów zaprojektowania, zakupu i montażu kotew wzmacniających, a inwestycja taka musi być realizowana wspólnie z inwestycją termomodernizacyjną, która będzie objęta wsparciem w wysokości 16% kosztów.

Co również z satysfakcją należy odnotować, zwiększenie takiej premii do 60% będzie dotyczyło obiektów zabytkowych lub obiektów, które znajdują się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. Wspominałem już na początku o rozszerzeniu katalogu podmiotów uprawnionych, które mogą się ubiegać o premię remontową. Ta nowelizacja ustawy włącza do kręgu podmiotów uprawnionych wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. Ta nowelizacja również zwiększa premię termomodernizacyjną z 16% do 21% wartości przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przypadku zainstalowania odnawialnego źródła energii w budynku, który jest poddawany termomodernizacji. Efektem ustawy zgodnie z informacją rządu ma być poddanie pracom remontowym ok. 30 tys. budynków komunalnych i, co ważne, nie mniej jak 4 tys. budynków z wielkiej płyty.

W bieżącym roku nie będzie wymagane dodatkowe wsparcie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, gdyż na koniec 2019 r. na jego koncie odnotowano wolne środki w kwocie ok. 248 mln i ta kwota wystarczy na sfinansowanie wszystkich zadań funduszu w bieżącym roku. Chcę jeszcze odnieść się do kilku wątków, które były referowane przez przedstawicieli różnych klubów w ramach dyskusji nad tym projektem. Przede wszystkim warto odnotować, iż de facto wszystkie kluby parlamentarne wysoko oceniły projekt rządowy, udzieliły mu wsparcia. Z satysfakcją odnotowano zwiększenie wsparcia, które jest zapisane w projekcie, które wzrasta odpowiednio do 50% bądź 60% kosztów danego projektu, jeśli dotyczy to budynków gminnych, w których wszystkie lokale należą do mieszkaniowego zasobu gminy.

Gminy według informacji strony rządowej posiadają aktualnie 35 600 budynków wielorodzinnych, w których znajduje się ponad 255 000 mieszkań.

Pozwala to przyjąć założenie, że wsparciem zostanie objętych ok. 30 tys. budynków z zasobów gminnych, tj. ok. 85% tych zasobów.

Dotychczas objęte nim były spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty z większościowym udziałem gminy.

Ale to nie dotyczy oczywiście wprost samego projektu.

Po pierwsze, jednym z warunków uzyskania takiego wsparcia w wysokości 50% jest zapewnienie w budynku wyremontowanym ze wsparciem budżetowym, że źródła ciepła spełniają współczesne standardy i nie przyczyniają się do emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery. Tutaj poprawkę w trakcie prac nad projektem zgłosił pełnomocnik rządu ds. czystego powietrza. Po drugie, gminy mogą osiągnąć ten cel poprzez wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej lub zamianę źródła energii. Wspominałem tutaj o preferencji w wysokości premii termomodernizacyjnej, jeśli są uwzględniane aspekty odnawialnych źródeł energii.

Można założyć, że zachowanie tych standardów realizacji inwestycji spowoduje jeszcze większą poprawę efektywności energetycznej, co przyczyni się do zmniejszenia opłat za ciepło oraz poprawy komfortu cieplnego mieszkańców. Reasumując, pragnę w imieniu Komisji Infrastruktury wyrazić podziękowanie dla strony rządowej za dialog, który prowadziliśmy w trakcie prac. Dziękuję również przedstawicielom Biura Legislacyjnego.

A to na pewno wpłynie w sposób, można powiedzieć, bardzo konkretny, wymierny na strategię mieszkaniową, którą przyjmuje gmina raz na 5 lat. Można oczywiście spodziewać się szeregu decyzji inwestycyjnych i pewnej korekty polityki mieszkaniowej, której głównymi beneficjentami - w szczególności, jeśli chodzi o gminy - będą te zasoby, które są w 100% własnością gminy, ale również oczywiście wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy (Dzwonek), które na podstawie tej ustawy również z tych środków publicznych będą mogły korzystać. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła.

Wznawiam obrady. Szanowni Państwo! Wysoka Izbo!

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Dziękuję bardzo. Wracamy do punktu 9. porządku obrad. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, druki sejmowe nr 128 i 168. Projekt dotyczy zwiększenia efektywności interwencji publicznych realizowanych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów, co ma na celu poprawę stanu technicznego zasobów mieszkaniowych i poprawę warunków mieszkaniowych społeczeństwa, co przyczyni się równocześnie do realizacji innych priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości, takich jak poprawa efektywności energetycznej, walka ze zjawiskiem smogu i walka z ubóstwem energetycznym. Potrzeba przeprowadzenia proponowanej nowelizacji wynika z oceny skutków funkcjonowania w okresie ostatnich 10 lat zasad udzielania wsparcia na termomodernizację i remonty oraz ich wpływu na poprawę stanu technicznego budynków. W ubiegłym roku rząd Prawa i Sprawiedliwości uruchomił program pilotażowy dotyczący termomodernizacji domów jednorodzinnych. Obecnie dążymy do tego, by ustawa po 10 latach została znowelizowana, co oznacza pomoc w przypadku termomodernizacji bloków, czyli budynków z wielkiej płyty, większe wsparcie dla inwestycji samorządowych oraz kompleksowych termomodernizacji. Proponowana nowelizacja stanowi odpowiedź na następujące problemy: niezadowalający stan techniczny ścian zewnętrznych budynków wykonanych w technologii wielkopłytowej, wymagający interwencji w przypadku wykonywania docieplenia; zmianę uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i środowiskowych, w związku z którymi powinno się promować głęboką termomodernizację i kompleksowe prace termomodernizacyjne; konieczność wsparcia samorządów gminnych w przedsięwzięciach poprawiających stan techniczny mieszkaniowych zasobów komunalnych; zwiększenie efektów działań wspierających remonty budynków; ograniczenia w dostępności premii kompensacyjnej.

Podstawowe rozwiązania przewidziane w projekcie to: dodatkowe wsparcie dla właścicieli i zarządców budynków z wielkiej płyty na wykonanie dodatkowych połączeń między warstwą nośną a warstwą fakturową ścian zewnętrznych; premia w wysokości 50% kosztów zaprojektowania, zakupu i montażu kotew wzmacniających, przy czym inwestycja taka musi być realizowana wspólnie z inwestycją termomodernizacyjną, która będzie objęta wsparciem w wysokości 16% kosztów; wsparcie samorządów gminnych w przedsięwzięciach remontowych; premia remontowa dla gmin przy wykonywaniu remontów budynków, w których znajdują się mieszkania wchodzące w skład zasobu komunalnego, przy czym wysokość premii - 50% wartości przedsięwzięcia remontowego; zwiększenie premii do 60% w przypadku obiektów zabytkowych lub znajdujących się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, poszerzenie katalogu podmiotów mogących ubiegać się o premię remontową, umożliwiające włączenie do grona beneficjentów instrumentu m.in. wspólnot mieszkaniowych z większościowym udziałem gminy; zwiększenie premii termomodernizacyjnej z 16% do 21% wartości przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w przypadku zainstalowania instalacji odnawialnych źródeł energii w budynku poddawanym termomodernizacji.

Dodatkowo budżet będzie nadal finansował aktualne inwestycje termomodernizacyjne i remontowe w kwocie ok. 100 mln rocznie.

Wysoka Izbo! Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość popiera rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Będziemy głosowali za przyjęciem tego projektu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska głos zabierze pan poseł Dariusz Joński. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej mam przyjemność przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Projekt ustawy ma na celu poprawę stanu technicznego, o którym była mowa, zasobów mieszkaniowych i warunków mieszkaniowych społeczeństwa, ale w ustawie jest też mowa o poprawie efektywności energetycznej, walce ze zjawiskiem smogu, w walce z ubóstwem energetycznym. Można by było powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości obudził się po paru latach z letargu, bo na polu ochrony środowiska, co jak co, ale PiS zderzył się ze ścianą w ostatnich latach. Najlepszym przykładem był 2017 r., kiedy wpłynął do Sejmu projekt zmian o odnawialnych źródłach energii, który tak de facto w ogóle zastopował rozwój odnawialnych źródeł energii. Prawie 1 tys. małych przedsiębiorców wstrzymało jakiekolwiek działania inwestycyjne, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Dopiero w 2019 r. pan minister Tchórzewski ogłosił, że dziś możemy startować z OZE, bo: była niepewność co do przyszłości źródeł węglowych - to cytat. Dobrze, że ten projekt ustawy się pojawił.

Natomiast mamy też dwa kolejne założenia.

Mówimy tu o premii, która może wynieść 50% kosztów przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych.

I jest ten trzeci obszar dotyczący wielkiej płyty.

Pan poseł mówił m.in. o tym, że można wymieniać tę termomodernizację na grubszą itd., ale przecież większość przede wszystkim spółdzielni mieszkaniowych już to wykonała, więc nie będzie tego robiła po raz drugi. A sprawa faktycznie jest dość istotna, bo chodzi o tzw. kotwy łączeniowe, które zagrażają bezpieczeństwu, i to powinno zostać poprawione, bo same płyty mają się nieźle. Krótko mówiąc, projekt jest godny poparcia, przy czym warto zauważyć, i chcę z tego miejsca o tym powiedzieć, że albo rząd przygotuje dodatkową propozycję, tak aby objąć tym budynki użyteczności publicznej, albo po prostu klub Koalicji Obywatelskiej złoży oddzielny projekt ustawy, tak żeby mogły być podjęte termomodernizacja i remont tych budynków.

Dziękuję bardzo, panie pośle. Zapraszam. Panie Ministrze! My również odnosimy się bardzo pozytywnie do omawianej ustawy, do rozszerzenia listy podmiotów, które będą mogły z niej korzystać.

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mówimy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, druki nr 128 i 168.

Zawsze się mówiło, że jest to relikt komunizmu, ale w tych blokach żyje wiele Polek i Polaków, żyją ludzie, którzy mają bardziej bądź mniej zasobne portfele, emeryci, o których dzisiaj tak dużo mówiliśmy, i trzeba to realizować. Dobrze też, że pojawia się kwestia spięcia termomodernizacji z tymi projektami, w których będą uwzględnione inwestycje w odnawialne źródła energii, panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe na tych blokach. To jest potrzebne. Brakuje mi jednego jeszcze - gniazd do ładowania samochodów elektrycznych, bo gdzie te milion aut będziemy ładować? Przy każdym z takich dużych bloków powinno się takie gniazdo znaleźć.

Myślę, że też dzisiaj nie przyspieszy aż tak mocno realizacja tego programu. Zostały w ostatnich latach wyrzucone duże projekty OZE, chociażby wykorzystujące energię wiatrową, miały funkcjonować duże farmy wiatrowe. Dzisiaj się to próbuje zastąpić jakimiś tam mikroinstalacjami, a tak naprawdę nie wiemy, jak będą one funkcjonować w miastach, gdzie mamy różne natężenie tego. Czekamy, że to pozytywnie wpłynie na zmiany.

Tu padają duże liczby. Pojawia się kwestia chociażby zabytków. Też faktycznie warto pomyśleć o tym, żeby zająć się wymianą stolarki okiennej, drzwiowej, spiąć to wszystko razem.

Dlatego też jako klub Koalicja Polska - Polskie Stronnictwo Ludowe - Kukiz15 będziemy głosować za wprowadzeniem tej zmiany ustawy, traktując to jako projekt ważny i oczekiwany przez Polki i Polaków po to, żeby wszystkim żyło się lepiej, bezpieczniej w tych blokach z dużej płyty. Mam nadzieję, że przynajmniej po przeprowadzeniu tych inwestycji Polacy będą płacić mniej za energię elektryczną (Dzwonek), którą dogrzewają się w tych blokach. Czas na zadanie pytania - 1 minuta. Jako pierwszy pytanie zadaje pan poseł Przemysław Koperski, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. W takim razie pan poseł Jarosław Gonciarz, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Uzasadnienie projektu ustawy wskazuje, że o podwyższoną premię można się ubiegać w przypadku przedsięwzięć, które dotyczą m.in. wyłącznie budynków wielorodzinnych, których jedynym właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego. Praktyka pokazuje jednak, że w ciągu ostatnich lat wykupiono wiele mieszkań komunalnych, a liczba budynków, w których gmina jest jedynym właścicielem, jest coraz mniejsza. Prosiłbym o doprecyzowanie, czy ten przepis dotyczy budynków, gdzie gmina ma 100% swoich mieszkań, czy też budynków komunalnych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, ale w których wykupiono przynajmniej jedno mieszkanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Dyduch, klub parlamentarny Lewica. Bardzo proszę. Wysoki Sejmie!

Ja nie mówię, że ten, ten jak każdy następny.

Jest pytanie, ile tutaj szacujemy oszczędności z tego tytułu dla mieszkańców, przy tym nakładzie x, który będziemy przekazywać, ile oni zaoszczędzą.

Dziękuję. Pan poseł Mirosław Suchoń, Koalicja Obywatelska. Nie widzę. W takim razie lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Na pytania odpowie podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju pan minister Robert Nowicki. Zapraszam serdecznie.

Wysoka Izbo! Na początku chciałbym podziękować wszystkim parlamentarzystom, szczególnie panom posłom sprawozdawcom w zakresie tej ustawy w komisji. Myślę, że ta ustawa jest niezmiernie potrzebna, ponieważ ona celuje właśnie w te warstwy, gdzie jest najbardziej potrzebna pomoc, to znaczy w warstwy, gdzie gminy gospodarują swym zasobem. To wciąż, jak przypomnę, 35 tys. budynków, więc to nie znaczy: tylko, to znaczy: aż. 35 tys. budynków to kilkaset tysięcy mieszkańców. Efektywność energetyczna.

To jest ok. 200 tys. do termomodernizowania, z tego 35 tys., gdzie 100% udziałów w strukturze właścicielskiej ma gmina, a 95 tys., gdzie jest współwłasność z innymi podmiotami. Ile oszczędzą mieszkańcy? To jest 43% efektywności według danych.

W tym punkcie mamy wyraźnie powiedziane, jak rząd wspiera samorządy w walce z ubóstwem energetycznym, [[Oklaski]] w walce dotyczącej kwestii jakości powietrza w gminach. Chcę powiedzieć też w odniesieniu do wystąpienia pana posła Dariusza Jońskiego - niestety nie mam możliwości bezpośrednio skierować tego do pana posła - że to nie jest tak, że tylko budynki mieszkalne mogą korzystać ze wsparcia, z premii termomodernizacyjnej. Z premii termomodernizacyjnej mogą także korzystać obiekty użyteczności publicznej. Dodatkowo, o czym nie było mowy, środki NFOŚ są do wykorzystania też na obiekty użyteczności publicznej.

Jak wynika z analiz, obiekty komunalne często są substandardowe.

Pozostałe to jest 15%. Mam na myśli te, gdzie nie ma tej 100-procentowej struktury. To przewiduje nowela. Tego nie ma dzisiaj, to należy wyraźnie podkreślić i komunikować.

Różna struktura właścicielska może być w spółce. A jeżeli nie ma 100%, to dostaje 15%.

A w kolejce do realizacji tego programu termomodernizacji czy też remontów są budynki znacznie starsze.

Walka związana z jakością powietrza, ze zdrowiem, panie pośle - kieruję to do pana posła Dariusza Jońskiego - to nie tylko 2019 r., bo jeśli spojrzeć na dane z 2016 r., to instalacji fotowoltaicznych było ok. 16 tys. W 2019 r. w pierwszym kwartale było 85 tys. Znakomity wzrost ilości instalacji fotowoltaicznych. A więc widać ewidentnie na przykładzie tych lat, jak możemy walczyć w kwestii tego miksu energetycznego.

Dziękuję bardzo, panie ministrze. Do głosu zapraszam też sprawozdawcę komisji pana posła Jerzego Polaczka. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Jak powiedziałem, przede wszystkim ona rozszerza krąg podmiotów uprawnionych. To są, po pierwsze, samorządy terytorialne, czyli jednostki samorządu terytorialnego, jakimi są gminy, po drugie, uwzględnia się w tych rozwiązaniach możliwość wsparcia wspólnot mieszkaniowych, czyli zasobu komunalnego zarządzanego przez gminę, który ma już tę strukturę własnościową mieszaną, po trzecie, daje wyjątkowo wysoką premię remontową, do wysokości 50% wartości projektu, w przypadkach budynków zabytkowych nawet do wysokości 60% - tego nie było, po czwarte, przede wszystkim zwiększa nakłady na ten cel, jakim jest obniżenie kosztów utrzymania w zasobach mieszkaniowych.

One należą głównie do spółdzielni mieszkaniowych.

Chcę również jako poseł sprawozdawca rozszerzyć tę krótką informację, o której już wspomniał pan minister: to nie jest jedyne źródło finansowania tych przedsięwzięć, bo pamiętajmy, iż zarówno program operacyjny związany z likwidacją niskiej emisji finansowany przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska w tej perspektywie europejskiej daje beneficjentom, wśród których są również m.in. wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, inni zarządcy, możliwość uzyskania premii inwestycyjnej w wysokości 45% całkowitego kosztu przedsięwzięcia.

Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia dodatkowego sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (druki nr 159 i 175) Proszę panią poseł Annę Paluch o przedstawienie sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Wysoka Izbo! Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, które przepisy należy stosować do postępowań administracyjnych wszczętych przed dniem 31 grudnia 2014 r. i dotychczas niezakończonych dotyczących udzielenia koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 1 Prawo geologiczne i górnicze, tzn. objętych własnością górniczą, z wyłączeniem złóż węglowodorów. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem zawartym w omawianym projekcie ustawy stosowane będą przepisy w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2014 r., co pozwoli na wyeliminowanie jakichkolwiek niepewności interpretacyjnych w tym zakresie. Przyjęta reguła intertemporalna potwierdza poszanowanie praw nabytych stron pozostających nadal w toku postępowań koncesyjnych. Pozostaje ona również w zgodzie z zasadą zaufania obywateli do państwa i do prawa. Wysoka Izbo!

Ta ustawa zmieniająca Prawo geologiczne i górnicze zawiera szereg przepisów przejściowych odnoszących się m.in. do postępowań w zakresie węglowodorów, zatwierdzania dokumentacji hydrogeologicznych, dokumentacji geologiczno-inżynierskich czy też postępowań dotyczących opłat eksploatacyjnych. Nie zawiera natomiast żadnych przepisów dotyczących postępowań o udzielenie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin objętych własnością górniczą, oczywiście z wyłączeniem złóż węglowodorów. Wysoka Izbo!

W VIII kadencji przepisy tej ustawy z 11 lipca 2014 r. były trzykrotnie nowelizowane i poprawiane ustawami, których projekty zawarte były w drukach nr 364, 996 i 2551. Błędy w przepisach uniemożliwiały prawidłowe prowadzenie postępowań koncesyjnych. Konieczne było wprowadzanie samoistnej podstawy prawnej w przypadku zmiany koncesji, żeby nie korzystać z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Dokonano korekty przepisów przejściowych regulujących kwestię koncesji udzielonych na podstawie przepisów sprzed wejścia w życie nowelizacji z 2014 r., w tym spraw dotyczących ważnych praw nabytych. Wysoka Izbo! Dokonywano również modyfikacji przepisów regulujących zasady wykonywania koncesji i naliczania opłaty koncesyjnej, podział pomiędzy uprawnione podmioty. Te zmiany, które były dokonywane, jak mówię, w VIII kadencji, dały możliwość objęcia przepisami wykonawczymi koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów z wniosków złożonych przed dniem 30 września 2014 r., a udzielonych po tej dacie. I pytanie, skąd ta data się wzięła. Ano z przepisu o charakterze retroaktywnym, który był zawarty w art. 11 ust. 2 tej ustawy z 2014 r., który umorzył wszystkie wnioski o wydanie koncesji złożone w okresie 3 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy.

Umorzono postępowania z wniosków złożonych po 30 września, ale były wszczęte postępowania z wniosków złożonych wcześniej. Nie było przepisów, które umożliwiłyby prawidłowe naliczenie opłat eksploatacyjnych, koncesyjnych, podziału tych opłat między uprawnione podmioty, nie było podstaw prawnych do egzekucji. Można by jeszcze długo mówić o tych błędach. Wracam do tej działalności prawodawczej z ubiegłej kadencji, ponieważ omawiany projekt ustawy zawarty w druku nr 159 odpowiada również na komplikacje i problemy wywołane przez tę nieszczęsną nowelizację z 11 lipca 2014 r.

Postępowania te toczą się na tym etapie na skutek orzeczeń sądów administracyjnych uchylających poprzednie rozstrzygnięcia ministra środowiska kończące te postępowania. Natomiast postępowania przed sądami administracyjnymi w każdej z tych spraw, które się toczą, toczyły się ok. 4 lat.

Wysoka Izbo! Ustawa o zmianie Prawa geologicznego i górniczego z 2014 r. odmiennie uregulowała zasady dotyczące udzielania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin objętych własnością górniczą, wprowadzając tzw. procedurę open door. To znaczy, że w przypadku złożenia wniosku koncesyjnego ogłasza się możliwość składania kolejnych wniosków koncesyjnych w sprawie wykonywania tej samej działalności w tej samej przestrzeni. Organ ocenia wówczas wszystkie złożone wnioski. Na tym polega procedura open door. Ona pozwala na przeprowadzenie postępowania koncesyjnego na wniosek przedsiębiorcy, przy czym to minister wyznacza czas i obszary, dla których chce udzielić koncesji. To jest procedura dużo sprawniejsza i tańsza, więc warto było ją wprowadzić.

W porządku prawnym obowiązuje zasada działania nowego prawa wprost, tzn. w przypadku braku przepisu przejściowego, który odnosi się jednoznacznie do danych stosunków, zastosowanie w tym przedmiocie mają przepisy nowej ustawy, więc po prostu musimy to rozstrzygnąć ustawą, o której tutaj rozmawiamy. Ta zasada stosowania nowych przepisów nie ma charakteru bezwzględnego. Są sytuacje, gdy nowych przepisów po prostu nie da się zastosować. Wówczas powinno się stosować dotychczasowe przepisy.

Nie wiemy, proszę państwa, jaką interpretację w tym zakresie przyjęłyby sądy administracyjne, które będą badać rozstrzygnięcia w II instancji, bo należy zakładać, że będzie się toczył proces odwoławczy czy dalsza kontynuacja w trybie sądowym. Minister klimatu ze względu na wagę tych postępowań koncesyjnych musi mieć pewność, jakie przepisy należy zastosować do tych postępowań, a tę pewność dają właśnie przepisy ustawowe, które jednoznacznie przesądzają, że postępowania będą się toczyć na podstawie przepisów, które obowiązywały w momencie ich wszczynania. Wysoka Izbo! Przypominam, że dzisiaj odbyło się pierwsze czytanie tego projektu. To jest projekt bardzo krótki, 2-artykułowy. W trakcie szczegółowych prac nad projektem przyjęto poprawkę proponowaną przez Biuro Legislacyjne, odnoszącą się do tytułu ustawy.

Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa uprzejmie proszę o uchwalenie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, zawartego w sprawozdaniu komisji ochrony środowiska z druku nr 175. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i koła. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pani poseł sprawozdawca komisji bardzo wyczerpująco omówiła ten punkt, ponieważ faktycznie projekt nowelizacji jest krótki. On właściwie dotyczy wyłącznie wprowadzenia przepisu przejściowego do ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Przepis ten jest konieczny ze względu na nadal będące w toku postępowania koncesyjne toczące się przed Ministerstwem Klimatu w II instancji na skutek orzeczeń sądów administracyjnych uchylających poprzednie rozstrzygnięcia. Ze względu na to, iż ww. postępowania były wszczęte przed wejściem w życie ustawy o zmianie Prawa geologicznego i górniczego na podstawie przepisów wówczas obowiązujących, a obecnie w II instancji nie można zastosować nowych regulacji, należy rozstrzygnąć ustawowo, iż te postępowania powinny zakończyć się na podstawie tych samych regulacji, na podstawie których zostały wszczęte. Minister klimatu ze względu na wagę ww. postępowań koncesyjnych musi mieć pewność, jakie przepisy należy zastosować do tych postępowań, a tę pewność dają jedynie regulacje ustawowe. Zresztą tych postępowań - bo takie też były pytania - jest zaledwie kilka. Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Koalicja Obywatelska wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Natomiast dzisiejsze posiedzenie komisji, które odbyło się o godz. 8.30 i trwało 30 minut, wzbudziło szereg wątpliwości posłów i posłanek zasiadających w komisji. Zadaliśmy państwu proste pytanie: Jakie podmioty, które złożyły swoje wnioski przed 31 grudnia 2014 r., będą podlegać tym zmianom? Jakich podmiotów to będzie dotyczyć? Przez ponad pół godziny tych pytań padło z sali pewnie pięć albo dziesięć. Nie mogliśmy się doprosić o tę odpowiedź. W związku z tym rodzą się wątpliwości, które podmioty będą beneficjentami tej nowelizacji. Czy nie jest to czasem próba ominięcia przepisów, które w tej chwili obowiązują po tamtej nowelizacji, i cofnięcia się do przepisów z 2014 r. Czy nie jest to również próba obejścia sądów i ich rozstrzygnięć na temat tego, które przepisy powinno się stosować - czy te sprzed nowelizacji, czy te po nowelizacji?

Ten wniosek nie został przegłosowany. Padł kontrwniosek pani poseł Paluch, żeby zakończyć dyskusję. Nie został przegłosowany pozytywnie, nie został przyjęty. Nie rozumiemy, dlaczego w takiej sytuacji ucina się dyskusję.

W związku z tym nie mam pewności, że to jest kompletna lista. Co więcej, minister klimatu wprost przyznaje, że de facto chcemy stosować przepisy sprzed nowelizacji, czyli z roku 2014, do postępowań, które będą ponownie rozpatrywane. Chyba powinny być rozpatrywane już zgodnie z nowymi przepisami, skoro te nowe przepisy zostały przegłosowane. Nie mieliśmy czasu, ponieważ to pismo wpłynęło bardzo późno, aby zapoznać się szczegółowo z tymi konkretnymi przypadkami, sprawdzić, czy czasem nie będzie tam naruszony jakiś interes mieszkańców, jeżeli chodzi o to, że te wnioski będą procedowane wedle tych starych przepisów, a nie nowych. Na koniec chciałbym powiedzieć o wątpliwościach Biura Legislacyjnego, które wprost stwierdza, że wątpliwości budzi propozycja dodania nowego przepisu w art. 18 ustawy. Przepis ten jest przepisem częściowym. Takie rozwiązanie budzi wątpliwości co do jego zgodności z konstytucyjnymi zasadami pewności prawa oraz zakazu retroakcji. I w tej sprawie wydaje się konieczne zasięgnięcie opinii Biura Analiz Sejmowych, o którą to opinię również się zwróciliśmy. Takiej opinii nie dostaliśmy. Co więcej, nasze wątpliwości budzi również to, iż projekt, który powinien być procedowany w trybie ministerialnym, jest procedowany w trybie poselskim. Państwo uciekacie od odpowiedzi na nasze pytania. W związku z tym w imieniu Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni na podstawie art. 45 ust. 2 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej wnoszę o odrzucenie w drugim czytaniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ten projekt ustawy wygląda niewinnie. Akt prawny liczy ok. 100 słów. Do tego jest krótkie uzasadnienie. Niewiele, zważywszy na to, ze cały projekt ustawy, cały akt prawny Prawo geologiczne i górnicze liczy sobie 266 stron. Z pozoru wszystko wygląda rzeczowo. W uzasadnieniu czytamy, że projekt ustawy doprecyzowuje postępowania administracyjne i pozwoli na wyeliminowanie niepewności interpretacyjnych. Tak też tutaj zostało to przedstawione. Dla niepoznaki dodaliście w uzasadnieniu zdanie, że ustawa pozostaje w zgodzie z zasadą zaufania obywatela do państwa. Świetnie, tylko że to jest oszukiwanie obywateli. Jak podaje Biuro Legislacyjne, projekt nie został zaopiniowany przez żadną z instytucji, które są do tego powołane na mocy różnych ustaw, tj. Krajową Radę Radców Prawnych, Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Izbę Gospodarczą, Radę Dialogu Społecznego, prokuratora generalnego. I wy macie czelność uzasadniać tę ustawę zasadą zaufania obywatela do państwa? A to nie koniec. Biuro Legislacyjne wyraziło również wątpliwość, czy ta zmiana ustawy jest zgodna z konstytucyjnymi zasadami pewności prawa oraz zakazu retroakcji, czyli działania prawa wstecz. Rekomendacją biura jest, aby w tej sprawie zasięgnąć opinii Biura Analiz Sejmowych. Tej opinii nie otrzymaliśmy. Wbrew wszelkim zasadom przepychacie kolanem ten projekt. Czy na tej podstawie można budować zaufanie obywatela do państwa? Żartujecie sobie z nas, posłanek i posłów, żartujecie sobie z obywateli. Nasuwa mi się pytanie: Dlaczego? Dlaczego pomimo negatywnej opinii idziecie jak walec z tą ustawą? Dlaczego nie konsultujecie jej z instytucjami, które są do tego powołane? My tego nie wiemy. Nasuwają się przypuszczenia, że rząd próbuje coś ukryć lub wpłynąć na wyroki sądowe w sprawach, które jeszcze się toczą. Prawo geologiczne i górnicze powstało po to, aby wyważyć interesy stron, przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości gruntowych. Przepisy z jednej strony zapewniają przedsiębiorcy łatwiejszy dostęp do złoża, a z drugiej chronią właścicieli nieruchomości, zapewniając możliwość występowania z roszczeniem. A wy chcecie to zmienić. Z niewiadomych powodów chcecie bronić praw korporacji, a nie obywateli.

Czyich bronicie interesów? To, co robicie, to są kpiny z procesu tworzenia prawa. Przypomnę, ta ustawa ma 266 stron.

W tym bałaganie nie da się dobrze stanowić prawa i wy dobrze o tym wiecie. Więcej, o to wam właśnie chodzi, ponieważ w tym bałaganie łatwiej ukryć błędy i celowe niszczenie prawa, tak żeby chroniło was, rządzących, a nie obywateli. Klub Lewicy nie będzie popierał prawa, które jest źle przygotowane i nie jest skonsultowane. Wnosimy o odrzucenie projektu ustawy. Dziękuję bardzo, pani poseł. Dziękuję. W imieniu klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego - Kukiz15 pan poseł Andrzej Grzyb. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Taka mała nowela a tyle emocji, jak również krytycznych ocen.

W ocenie wnioskodawców nie można zakończyć tych postępowań, ponieważ nie można zastosować przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2015 r. To zostało potwierdzone również przez resort środowiska, przez wiceministra tego resortu oraz głównego geologa kraju.

Było to związane z brakiem informacji w uzasadnieniu, ale również w wyjaśnieniach w pierwszym czytaniu, które nie przyniosły oczekiwanej klarowności, kto będzie beneficjentem tej zmiany.

Stąd też myślę, że to nie jest nawet zamierzona złośliwość wobec wnioskodawców, tylko kwestia rzeczywistego wyjaśnienia. No i otrzymaliśmy to wyjaśnienie. Odnotowałem - akurat komisja do spraw środowiska i zasobów naturalnych przesłała to wyjaśnienie bodajże o godz. 18 z minutami - że dotyczy to pięciu postępowań, przy czym są wymienione obszary koncesyjne.

No, ale to wyjaśnienie otrzymaliśmy.

W chwili obecnej chcielibyśmy jeszcze dokonać pewnej oceny tego wszystkiego, co mamy, łącznie z całym przebiegiem dyskusji, wtedy podejmiemy decyzje co do naszego ostatecznego stanowiska. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.

Jako Konfederacja z nieukrywanym zdziwieniem przyjmujemy do wiadomości to, że na posiedzeniu komisji nie ujawniono, jakich konkretnie podmiotów dotyczy omawiana ustawa.

Dobrze wiemy, że został on jednak opracowany w ministerstwie, a nie przez posłów. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli jednoznacznie wynika, że bez rozpoznania pozostaje powyżej 13% wniosków o udzielenie lub zmianę koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż miedzi, a kolejne 2,5% to sprawy w toku.

Światowe wydobycie opiera się w tej chwili na rynkach, które bądź są niestabilne, czyli mają niestabilną sytuację polityczną, bądź - tak jak chociażby Chiny - blokują zewnętrzny dostęp. Należy podkreślić, że to właśnie poprzedni rząd nie zadbał o należyte przepisy intertemporalne w projekcie zmian własnej ustawy z 2014 r. W konsekwencji tych niedomagań z uwagi na kolejną implementację przepisów unijnych blokowane są dziś nawet wnioski złożone na 4 lata przed nowelizacją z 2018 r. Koło Poselskie Konfederacja opowiada się za uproszczeniem procedur dotyczących koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie złóż miedzi, aby skorzystać z koniunktury na te dobra naturalne, ponieważ dzisiaj cena miedzi jest bardzo wysoka, a nikt z nas nie wie, jak będzie za 10, 15 czy 20 lat. Ja jako poseł z ziemi lubuskiej. Nam szczególnie na tym zależy, ponieważ w naszym okręgu złoża miedzi są ogromne i chcielibyśmy, aby były jak najszybciej wydobywane, ponieważ byłaby to gwarancja ogromnego rozwoju dla całego województwa lubuskiego. Dodatkowo uważamy, iż nadwyżki pochodzące z opodatkowania rud miedzi lub ze sprzedaży tego surowca powinny na wzór norweski stanowić zabezpieczenie przed dramatycznie pogarszającą się w Polsce sytuacją w systemie ochrony zdrowia i ubezpieczeń społecznych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do pytań zapisało się pięcioro parlamentarzystów. Wyznaczam czas na zadanie pytania - 1 minuta.

Wysoka Izbo! Wydaje mi się, że państwo wnioskodawcy stosujecie sztuczki prawne. Nie wiem, pytam.

Tymczasem Ministerstwo Klimatu wydaje kolejne koncesje na wydobycie choćby węgla kamiennego nawet na terenach tak cennych przyrodniczo jak Rezerwat Biosfery UNESCO Polesie Zachodnie w otulinie Poleskiego Parku Narodowego, na terenach torfowisk chronionych konwencją Ramsar itd., itd.

Kolejne pytanie zada pan poseł Krzysztof Gawkowski, Lewica. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Panie Ministrze! Mam taką wątpliwość co do tego aktu prawnego. Co wy chcecie w nim ukryć? Dlaczego nie chcecie odpowiedzieć na pytania, które stawiać można przecież w wypadku każdej ustawy, ale ta z perspektywy inicjatywy poselskiej powinna być jasna i otwarta. Dlaczego nie powiecie jasno, że chodzi o kasę? Bo przecież chodzi o kasę. Tylko kto na tym zyska? Dlaczego podajecie obszary, a nie podajecie firm, które mogą być uprzywilejowane w związku z przyjęciem tego aktu prawnego, który de facto będzie nielegalny, bo to jest prawo, które ma działać wstecz. Mam konkretne pytanie: O jakie podmioty chodzi i o jakie pieniądze, jeśli ta ustawa zostanie przyjęta i kto na tym konkretnie będzie mógł skorzystać? Dziękuję bardzo. Pani poseł Małgorzata Janowska, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo!

Dziękuję bardzo. Pan poseł Marek Dyduch, Lewica. Pani Marszałek! Mam takie pytanie. Pani sprawozdawca, pani przewodnicząca Paluch powiedziała, że to jest wina tych wszystkich, co przyjęli nowelizację w 2014 r.

Tam była cała lista instytucji, które czekały na decyzję. Wiem, że chodzi o sprawy sądowe. Uważnie słuchałem. No to jak wracamy do starej ustawy, to po co było wszystko inne przez te lata? No po co to było? Dziękuję. Pan poseł Grzegorz Lorek, Prawo i Sprawiedliwość. Wysoka Izbo! Muszę powiedzieć, że to jest długo oczekiwana ustawa. Na każdą ścianę potrzebna jest koncesja. Co 5 lat kopalnia prosi o wydanie tej koncesji. Wiem, że członek klubu PSL jest byłym dyrektorem i on bardzo dobrze wie, jaką walkę musiał toczyć co 5 lat, żeby tę koncesję uzyskać. My jeszcze walczymy o Złoczew, pani poseł. Myślę, że pracownicy kopalni węgla brunatnego ucieszą się z pani słów. Natomiast chcę powiedzieć pani to, co pani poseł sprawozdawca powiedziała, mianowicie, że wreszcie mamy szansę to uporządkować, te działania, które są bardzo długotrwale robione w różnych instancjach.

Dziękuję. Dziękuję bardzo. W imieniu rządu na zadane pytania odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu pan minister Piotr Dziadzio. Proszę bardzo.

Szanowni Państwo! W odpowiedzi na dyskusję, bo tak to nazwę, dyskusję, którą w pewnym sensie można uznać za dyskusję niepotrzebną wobec potrzeby dokonania zmiany, która była przygotowana przez klub poselski Prawa i Sprawiedliwości i zreferowana tutaj przez panią Annę Paluch, posła sprawozdawcę, której bardzo dziękuję za przekazanie tych informacji Wysokiej Izbie. Szanowni Państwo! Odniosę się może bardzo całościowo do spraw, które zostały poruszone. Postaram się to syntetycznie państwu przedstawić, niemniej jednak szereg zarzutów, które tutaj usłyszeliśmy, to zarzuty tak naprawdę bezpodstawne, jeśli chodzi o przygotowanie, ukrywanie czegokolwiek. Zmiana ustawy, która jest proponowana, uporządkuje i umożliwi przeprowadzenie wydania koncesji poszukiwawczych i rozpoznawczych - jak tutaj już padło, państwo słyszeliście - w obszarze bogatych złóż miedzi. Szanowni Państwo!

W pierwszej kolejności powinniśmy zakończyć postępowania, które umożliwią nam wydanie koncesji poszukiwawczych i rozpoznawczych, to jest ten pierwszy element, żebyśmy mogli zrobić krok do przodu.

Szanowni Państwo! W zeszłym roku uzyskaliśmy wyroki, stąd tak długi proces. Dzisiaj, żebyśmy mogli zrobić krok jeszcze raz do przodu, powinniśmy przyjąć tę ustawę, która pozwoli podmiotom, które starają się o koncesje - jeszcze raz - na poszukiwanie i wydobywanie złóż rud miedzi i srebra, je uzyskać.

To jest proces, który wymaga spełnienia wszystkich obowiązków i całej procedury.

Czyli podmioty gospodarcze, które starają się o te koncesje, nie mogą stać w niebycie, powinny dostać możliwość skończenia i uzyskania koncesji, koncesji na poszukiwanie i wydobywanie. Jeszcze raz: przyznaję i potwierdzam.

Pozwólmy wydać te koncesje i przeprowadzić proces koncesyjny.

Potwierdzam to. Było również pytanie odnośnie do wydawania koncesji na wydobywanie węgla. Oczywiście, proszę państwa, ta sprawa nie dotyczy wydawania koncesji węglowych.

Dziękuję bardzo panu posłowi Krystianowi Kamińskiemu z Konfederacji, który wspiera przyjęcie tych rozwiązań.

Ustawa, która jest proponowana, nie jest w jakiejkolwiek sprzeczności z prawem unijnym, nie zagraża bezpieczeństwu obywateli, a w szczególności właścicieli nieruchomości.

My chcemy te koncesje wydać, ażebyśmy mogli świadomie udostępniać zasoby naturalne i z nich korzystać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Ale bardzo proszę, pani poseł, naprawdę, jeśli mogę apelować o krótkie.

Szanowni Państwo! Dziękuję przedstawicielowi PSL za rozsądne stanowisko, bo to przede wszystkim rozsądku trzeba w takich ściśle technicznych czy proceduralnych ustawach. To nie jest próba obejścia sądów. Przecież sądy, rozstrzygając, muszą brać pod uwagę przepisy prawa.

Co do wątpliwości Biura Legislacyjnego, to spodziewam się, że takie same wątpliwości Biuro Legislacyjne wyrażało w momencie procedowania nad ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. Wtedy ówcześnie rządzącej większości, którą dzisiaj reprezentował pan poseł z Platformy Obywatelskiej, nie drgnęła powieka, żeby dziesiątki wniosków złożonych 3 miesiące przed terminem wejścia w życie ustawy wyrzucić do kosza i, że tak powiem, nikt się wtedy nie przejmował retroaktywnością.

Więc, proszę państwa, dziękuję tym klubom i tym posłom, którzy wykazali się zdrowym rozsądkiem, bo przede wszystkim tym powinniśmy się kierować, procedując nad tak ważnymi ustawami.

W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w całości. Proponuję, aby Sejm nie odsyłał tego projektu ustawy ponownie do komisji. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważała, że Sejm propozycję przyjął. O, jest sprzeciw. W takim razie do głosowania w tej sprawie przystąpimy w bloku głosowań.

Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie jeszcze wygłosić oświadczenie? Nikt się nie zgłasza. Listę posłów zgłoszonych do oświadczeń uważam zatem za zamkniętą. Może ktoś z państwa byłby skłonny złożyć oświadczenie na piśmie. Byłabym naprawdę bardzo zobowiązana.

Zapraszam, pani poseł. Wysoka Izbo!

Chodzi o poprawienie dostępności dla pacjentów, ale także o zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ciągłości i stabilności finansowej szpitali. Tymczasem w praktyce powstał system na wskroś niewydolny. Nie poprawia się ani sytuacja ekonomiczna szpitali, w myśl tej ustawy, ani dostępność dla pacjentów, a wręcz odwrotnie. Bardzo negatywnie oceniana jest też praca na tzw. szpitalnych oddziałach ratunkowych, a także dostępność dla pacjentów. Należy zatem ocenić tę ustawę jako nieprzemyślaną, jako eksperyment na żywej komórce, na pacjentach. Podstawowym założeniem tej ustawy miało być bardzo elastyczne zarządzanie pieniędzmi, a także stopniowe wychodzenie szpitali z zadłużenia. Niestety większość placówek, które miały zadłużenie przed wejściem reformy, tylko je powiększyła po wprowadzeniu, a właściwie po wejściu ustawy o sieci szpitali.

Należy zatem zadać pytanie, co dalej, jakie rząd proponuje rozwiązania i czy weźmie pod uwagę opinie, a właściwie sugestie Najwyższej Izby Kontroli, która w wyniku przeprowadzenia kontroli po wejściu w życie ustawy o sieci szpitali pisze: Błędem było nieuwzględnienie podczas tworzenia sieci ani aspektów społecznych, ani możliwości terapeutycznych i diagnostycznych poszczególnych jednostek służby zdrowia, nie uwzględniono także aspektów demograficznych, epidemiologicznych ani też stopnia dostosowania infrastruktury poszczególnych placówek do obowiązujących przepisów prawa. Niestety obecnie przyjęty system finansowania, szanowni państwo, nie nadąża za zmieniającymi się błyskawicznie realiami finansowymi. Szpitale, w myśl umów, które realizowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zadłużają się, ponieważ umowy nie uwzględniają lawinowo rosnących kosztów. Dzieje się tak, szanowni państwo, że zarządy województw, marszałkowie tną koszty poprzez likwidację poszczególnych oddziałów szpitalnych - oddziałów onkologicznych, kardiologicznych, oddziałów, które ratują zdrowie i życie - po to aby ograniczyć koszty personalne, ograniczając tym samym dostęp pacjentów do świadczeń medycznych. To bardzo przykre, bo taka sytuacja ma miejsce w województwie lubelskim, a konkretnie w Lublinie, gdzie w czterech szpitalach robi się tzw. reorganizację poprzez likwidację bardzo ważnych, bardzo potrzebnych i bardzo obleganych oddziałów, do jakich należy oddział chirurgii piersi, gdzie specjaliści - specjaliści rangi krajowej, ogólnopolskiej, ale także międzynarodowej - niestety są albo właściwie będą zwalniani. Dziś doszła do mnie informacja, że kilku ordynatorów złożyło dymisję, ponieważ zostali zobligowani do tego, aby wskazać listę osób do zwolnienia. Szanowni Państwo! Bardzo proszę, najwyższy czas, aby rząd podjął konkretne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Moje oświadczenie dotyczy jednego z największych problemów ekologicznych, by nie powiedzieć: bomby ekologicznej na Górnym Śląsku. Toksyczne odpady po zlikwidowanych Zakładach Chemicznych Tarnowskie Góry uznawane są za jeden z największych problemów ekologicznych. Funkcjonujące od 1922 r. przedsiębiorstwo było jednym z największych w kraju producentów chemicznych związków nieorganicznych. Jego odpady poprodukcyjne przez całe dziesięciolecia deponowane były na zwałowiskach wokół zakładu bez odpowiedniego zabezpieczenia, a doprowadziło to do skażenia zarówno gleby, jak i wód powierzchniowych i podziemnych. Sytuacja ta jest jednym z najbardziej wyrazistych przykładów obrazujących to, w jaki sposób zakłady chemiczne, jeśli na czas nie podejmie się środków zaradczych, mogą negatywnie wpływać na środowisko naturalne regionu.

Z analizy wyników badań pozyskanych w ramach prowadzonego monitoringu wód podziemnych stwierdzono wysokie stężenia takich pierwiastków jak arsen, bar, bor, cynk, kadm, ołów czy stront. Wszystkie odpady poprodukcyjne zakładów chemicznych zalicza się do grupy odpadów szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. Co warto podkreślić, wciąż zalegające odpady stwarzają realne niebezpieczeństwo dla mieszkańców gmin położonych w zasięgu oddziaływania głównego zbiornika wód podziemnych nr 330 Gliwice, który stanowi rezerwuar wody pitnej dla północno-zachodniej części aglomeracji górnośląskiej. Popierając zabiegi, jakie w tej sprawie podjął powiat tarnogórski oraz rady gmin Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Zbrosławice, Tworóg, Wielowieś, Rudziniec, Pyskowice, Gliwice, Zabrze oraz zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, zwracam się do władz Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o podjęcie natychmiastowych oraz skutecznych działań mających na celu ostateczną likwidację zagrożeń, jakie stwarzają odpady po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne Tarnowskie Góry w Tarnowskich Górach w likwidacji. Czas najwyższy, aby niebezpieczne odpady zostały wreszcie całkowicie usunięte.

Dziękuję bardzo, pani poseł. Bardzo proszę. Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Ust. 1 art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej mówi: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Wielokrotnie mówi się, wręcz alarmuje, że ten podział w Polsce jest zagrożony. W Polsce polskie władze łamią konstytucję. 21 stycznia do Kancelarii Sejmu przybył sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, by wykonać prawomocne postanowienie sądu, czyli dokonać wglądu do list poparcia sędziów nowej KRS.

Powinno to głośno wybrzmieć: Cofnięcie delegacji nie jest i nie może być cofnięciem prawomocnego postanowienia sądu. Kancelaria Sejmu miała i wciąż ma obowiązek przedstawienia tych list poparcia. Kolejną niepokojącą sytuacją jest zachowanie prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie - czyli cofnięcie delegacji - i, co istotne, członka nowej rady Macieja Nowackiego, który specjalnie przerwał urlop, by cofnąć delegację sędziemu Juszczyszynowi, co jest ewidentnym utrudnieniem wykonywania czynności służbowych przez podległego mu sędziego. Skłaniam się do refleksji, że i prezes Nowacki prawdopodobnie narusza ten sam artykuł konstytucji. Zgodnie z prawem, a potwierdza to rzecznik olsztyńskiego sądu rejonowego, sędzia Juszczyszyn przebywał w Kancelarii Sejmu w pełni legalnie i należało okazać mu listy.

Ten przykład obrazuje patologię i fasadowość rządów prawa w Polsce. Cieszę się z jednej strony, że w TVP powstał nowy program interwencyjny nagłaśniający nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji publicznych w Polsce. Mam nadzieję, że już niedługo usłyszymy w nim o tym przypadku. Jak widać, kasty PiS-u w Polsce mają się bardzo dobrze.

Dziękuję. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pozwólcie państwo, że powiem o kilku sprawach, które dotyczą Pomorza Zachodniego, a dokładnie rzecz biorąc, gospodarki morskiej, bo to jest dla nas, dla tego miasta, dla tego regionu bardzo ważne. Zacznę od tego, że mamy fabrykę, która, szanowni państwo, miała produkować morskie podstawy do elektrowni wiatrowych, czyli właściwie to, co będzie nam w niedługim czasie bardzo mocno potrzebne - wydaje się, że tak powinno być - a zarząd tej spółki, w której 80% ma fundusz Mars, ogłasza upadłość. Szanowni Państwo! Ludzie w styczniu, na koniec stycznia nie będą mieli wypłat.

Drugi przykład, o którym chciałem powiedzieć - bo mówię o gospodarce morskiej i tak naprawdę będę się odnosił do działań Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - to Stocznia Szczecińska. Szanowni Państwo!

Tak było, szanowni państwo. Dzisiaj tam hula tylko wiatr. Swego czasu pan premier Pawlak mówił, że to nasze srebro narodowe, a dzisiaj, obawiam się, bardzo mocno zagrożone, jedno z dwóch pozostałych przedsiębiorstw państwowych.

Jeden z mniejszych programów unijnych, które wdrażamy w tej perspektywie, z mniejszym budżetem, a najbardziej zagrożony, jeśli chodzi o zasadę n+3. Co z Odrzańską Drogą Wodną, tak szumnie zapowiadaną wielką inwestycją za wielkie miliardy? Nic się, szanowni państwo, nie dzieje. Żadnych rozmów się nie prowadzi, a ostatnio 80 mln zł, które były przeznaczone na Międzyodrze, które miało zabezpieczać częściowo Szczecin przed wysoką wodą, zostało przesunięte nie wiadomo, w które miejsce.

A dodatkowo, szanowni państwo, mamy jeszcze zagrożenie zwrotem unijnych środków, bo ta fabryka powstała m.in. dzięki środkom z Unii Europejskiej, ale mieliśmy zagwarantować i miejsca pracy, i produkcję. Bardzo proszę pana premiera o zajęcie się tym tematem, bo naprawdę jest on bardzo trudny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Rada Powiatu Tucholskiego w województwie kujawsko-pomorskim zajęła stanowisko, w którym wyraża swoje zaniepokojenie sytuacją, w której Szpital Tucholski nie ma możliwości zapewnienia we właściwej formie nocnej i świątecznej opieki medycznej. Informacja przedstawiona przez prezesa Szpitala Tucholskiego na sesji rady powiatu jednoznacznie wskazuje, że problem z właściwą realizacją opieki jest związany z brakiem kadry medycznej.

37 absolwentów w pełni przygotowanych do tego zawodu trafiło na rynek pracy. Niestety w szkołach na poziomie powiatowym nie można kształcić innej kadry medycznej.

Szpitale powiatowe nie powinny same realizować nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Rada Powiatu Tucholskiego apeluje o podjęcie działań, które rozwiążą problem w sposób systemowy, co wpłynie na poprawę sytuacji związanej z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Dziękuję, pani marszałek. Dziękuję bardzo, panie pośle.

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Sprawa jest prosta. Kiedyś czytaliśmy i oglądaliśmy polskie komedie i śmialiśmy się z opisów świata i rozwiązań w tych komediach prezentowanych. Dzisiaj okazuje się, że to nie jest takie śmieszne, bo zarządzacie państwem i problemami, które sami najpierw tworzycie, tak jak to zostało pokazane właśnie w tych komediach. Przypomnę problem cukru rozwiązany przez prezesa Dyzmę, który bronił polskiego cukru i zgodził się zostać prezesem, cytuję: żeby pomagać ludziom takim jak wy. Prezes Dyzma kupował cukier od cukrowni po to, aby go zmagazynować. Magazynów nie musicie kupować, pieniędzy też nie musicie mieć, prezes Dyzma już wam ten problem rozwiązał. Oglądaliście, czytaliście, to wiecie. Podsumujmy kilka faktów i danych. Grozi to wstrzymaniem wydobycia i wysłaniem górników na przymusowe postoje. Po drugie, zwały w górnictwie są trzy razy wyższe niż na początku 2018 r. i wciąż rosną. Po trzecie, węgiel z Rosji zalewa Polskę. 9 mln t węgla z Rosji sprowadzono do Polski w 2019 r., nie uwzględniając oczywiście grudnia. Rok 2018 był rekordowy na przestrzeni ostatniej dekady pod względem importu do kraju węgla kamiennego.

Ale sprowadzamy też węgiel z Mozambiku czy z Kolumbii. Po czwarte, kiedyś chcieliście, pod publiczkę oczywiście, blokować import. Związkowcy sami przypominają wam, że przed dojściem do władzy to właśnie Jarosław Kaczyński krytykował sytuację, w której, cytuję: w Polsce więcej się węgla kupuje, niż sprzedaje. Po piąte, polskie społeczeństwo płaci wysoką cenę za podtrzymywanie przez was przestarzałych rozwiązań. Płaci za waszą nieudolność. Mowa tutaj tylko o kosztach dopłat do energetyki węglowej. A gdzie koszty zdrowotne, które wynoszą ponad 62 mld euro? A gdzie przyszłość górnictwa? Po szóste, jednocześnie nigdy w historii nie sprowadzaliśmy do Polski tyle prądu, co przez ostatni rok. Dwukrotnie pobiliśmy rekord importu energii elektrycznej. Te pieniądze wypływają poza Polskę. To tyle, jeśli chodzi o wspieranie przez was polskiej gospodarki. Kasa wam ucieka, bo nie umiecie w gospodarkę, nie umiecie w węgiel, nie umiecie w energetykę. Wreszcie po siódme, jedyne, co umiecie zrobić, to przewieźć węgiel z jednego miejsca na drugie, z jednej hałdy na drugą i ładnie to nazwać: centralny magazyn rezerw węgla energetycznego. Wiecie, jak to się nazywa? To jest klasyczne zamiatanie problemu pod dywan. Za chwilę zrobicie polski centralny magazyn rezerw. Albo zaczniecie go przechowywać pod ziemią. Kto za to płaci? Jak chcecie systemowo rozwiązać ten problem? Ludzie, wy chcecie przewieźć węgiel z jednego miejsca na drugie i nazywacie to rozwiązaniem problemu. Prezes Dyzma rozwiązał problem z cukrem lepiej, a w każdym razie śmieszniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Swoje dzisiejsze oświadczenie chciałbym poświęcić Fordonowi, największej dzielnicy Bydgoszczy, a 100 lat temu samodzielnemu miastu.

Jego zadaniem było zabezpieczenie mostu kolejowo-drogowego na Wiśle. Jeszcze wówczas nie przeczuwał, jak ważną rolę będzie pełnił w historii miasta Fordon, którego potem został burmistrzem. Niemiecki burmistrz Fordonu jeszcze w listopadzie 1919 r. wyjechał z miasta. Komisarycznym burmistrzem został restaurator i przedsiębiorca Konstanty Krygier. W skład komitetu miasta Fordon weszli m.in. Jan Bross, rektor szkoły Stanisław Born czy restaurator Franciszek Płotka. Przewodniczący rady miejskiej przekazał zarząd w ręce Konstantego Krygiera, a chwilę później nauczyciel Jan Bross wygłosił do zgromadzonych tłumnie mieszkańców płomienne przemówienie. Ludzie spontanicznie zaśpiewali „Rotę” oraz wznieśli trzykrotny okrzyk na cześć Polski. Następnie wszyscy zgromadzeni ruszyli z pochodem przez Fordon. Ulice były odświętnie przybrane, wisiały flagi, girlandy oraz patriotyczne hasła. Uniesieni duchem wolności ludzie obeszli dosłownie całe miasto, jakby ich obecność miała podkreślić, kto tu jest gospodarzem.

Ludzie spontanicznie zrobili zbiórkę pieniędzy na rzecz polskich patriotów z Górnego Śląska. W ten sposób chcieli podzielić się radością z dopiero co uzyskanej wolności z tymi, którzy musieli o wolność walczyć. Podniosły i historyczny dzień zakończył się wspólnym obiadem dla wszystkich uczestników manifestacji. Lokalni restauratorzy postanowili podjąć mieszkańców poczęstunkiem oraz zorganizowali dla nich wspólną zabawę.

Przez cały okres międzywojnia był to najdłuższy w Polsce most na Wiśle. Swoje dzisiejsze oświadczenie chciałem dedykować dwóm osobom, które niezwykle dbały i dbają o historię Fordonu: panu Henrykowi Wilkowi, autorowi wielu publikacji na temat historii Fordonu i najstarszej fordońskiej parafii, parafii pw. św. Mikołaja, oraz panu Damianowi Amonowi Rączce, autorowi jedynego przewodnika po Fordonie, człowiekowi, który społecznie oprowadza wycieczki po Fordonie i który na bieżąco prowadzi Starofordoński Spichlerz Historii poświęcony właśnie historii Fordonu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Bardzo proszę. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Moje dzisiejsze oświadczenie będzie mieć nieco inny charakter niż zwykle, będzie przede wszystkim zacytowaniem treści stanowiska Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w sprawie prób anarchizacji państwa przez środowiska prawnicze: „Prawo jest wyrazem woli narodu, jest narzędziem porządkującym życie społeczne. Natomiast prawo wyrażone w Konstytucji jest nie tylko punktem odniesienia wszelkich działań formalnych, ale jest głosem naszej polskiej, tysiącletniej tradycji. Jest najważniejszym głosem naszego narodu, ponieważ prawo jest z narodu i dla narodu. Tymczasem w ostatnich tygodniach jesteśmy świadkami ataków części środowiska sędziowskiego i szeroko rozumianego prawniczego na porządek prawny w Polsce. Działania tzw. 'Kasty nadzwyczajnej' zdumiewają nie tylko Polaków, takie działania są niespotykane w cywilizowanym świecie. Polityczne protesty, często inspirowane przez lobbystów, przez tajemnicze grupy, są w wykonaniu tego środowiska niedopuszczalne. To są działania, które w swej istocie są łamaniem prawa i prowadzą prosto do anarchii i zniszczenia polskiego państwa. Kto ma w tym interes? Kto inspiruje atak na polskie państwo? Prawnicy, a zwłaszcza sędziowie, powinni rozumieć literę i ducha prawa polskiego. Powinni. Bo nie może być tak, że urzędnicy, a nimi są przecież prawnicy, pytają się innych państw o zgodność polskiego prawa z polską Konstytucją. Nie może być tak, że jedno środowisko może decydować o całym państwie i narodzie. Nie może być tak, że prawnicy są bezkarni, a zwykły obywatel za 'batonika' idzie do więzienia. My, jako Związek i jako niepodlegli Polacy, nie zgadzamy się na działania tej części środowiska prawniczego, która kontestuje obowiązujący porządek prawny. W naszym odczuciu w prostej linii wywodzą się one z tradycji zdrajców przedrozbiorowych i komunistycznych. NSZZ 'Solidarność' zrodziła się z potrzeby niepodległości i wolności. Solidarność' zawsze stała na straży Polski wolnej, niezależnej i samorządnej, nigdy nie przestanie bronić naszej Ojczyzny. Dlatego w tym miejscu zajmujemy wyraźne stanowisko broniące polskiej racji stanu. Sprzeciwiamy niebezpiecznym próbom tworzenia porządku prawnego w naszej ojczyźnie przez instytucje zagraniczne, często nieprzychylnie ustosunkowane i zainteresowane destabilizacją społeczną w Polsce. Wąska grupa społeczna rości sobie prawo bycia ponad władzą ustawodawczą i wykonawczą, ponad państwem polskim i ponad naszym narodem. Solidarność' na to nigdy się nie zgodzi. Polska - nasza Ojczyzna, jest naszym największym dobrem, zawsze Jej bronić, dlatego mówimy głosem sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego - 'non possumus', ani kroku dalej - nie zgadzamy się na niszczenie Polski. Jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej, ale też prawie od 30 lat członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” dziękuję za te słowa. Niech w tych ważnych dniach będą słyszalne i niech będą wyrazem wsparcia dla nas, parlamentarzystów, w podejmowaniu tak ważnych dla Polski decyzji dotyczących polskich sądów. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie pośle. Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Kryzys klimatyczny jest faktem, a naukowcy od wielu lat podkreślają, że jego podstawową przyczyną jest emisja gazów cieplarnianych spowodowana niestety ludzką działalnością. Co roku Polska traci 150 mld zł. Umiera ponad 45 tys. ludzi. Śmiało można powiedzieć, że Polska choruje na smog. Tak duże zanieczyszczenie spowodowane jest m.in. ilością pieców węglowych niespełniających norm emisyjności, tzw. kopciuchów. Tylko w Bydgoszczy jest ich ponad 23 tys. Wszystkie trzeba pilnie wymienić.

Skuteczna walka ze smogiem wymaga nakładów finansowych. Dlatego zwracam się o przeznaczenie dodatkowych środków z narodowego funduszu ochrony środowiska oraz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska na rzecz termomodernizacji budynków, wymiany pieców węglowych oraz programów osłonowych w zakresie dopłat do wyższych kosztów ogrzewania innego niż węglowe, które byłyby dedykowane dla Bydgoszczy i okolicznych gmin. Bez tych działań i inwestycji skazujemy dziesiątki tysięcy ludzi na choroby i śmierć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Szanowna Pani Marszałek! Koleżanki i Koledzy Posłowie! Drodzy Lubuszanie! Oto dziś, 22 stycznia, ponownie wróciłem do Sejmu, by sprawować zaszczytną funkcję posła Rzeczypospolitej, dlatego teraz chciałbym zwrócić się do was z trzema refleksjami. Pierwsza koncentruje się na dobru i podziękowaniach wobec tych 8 tys. Lubuszan, którzy uznali 12 października minionego roku, że zasługuję na ich zaufanie, głosowali na mnie w czasie wyborów. Dziękuję i doceniam, szczególnie za pomoc i wsparcie każdej i każdego z was, którzy towarzyszyliście mi w tym 3-miesięcznym okresie swoistego czyśćca poza Sejmem, gdzie życzliwość konkurowała z zawiścią i złem, uczciwość z podstępem, czyny haniebne z chlubnymi. Skupiam się na dobru. Za każdy chwalebny czyn, dobre słowo i wsparcie dziękuję. Dziś odwzajemniam się tym samym, za dobro będę rewanżował się dobrem. Jednocześnie w drugim akapicie dziękuję wojewodzie lubuskiemu panu Władysławowi Dajczakowi za decyzję, która umożliwiła mi powrót do Sejmu. Pracy przed panem wojewodą wiele, wsparcie i żarliwe zabieganie o sprawy ziemi lubuskiej w Sejmie, w gabinetach ministerialnych jest konieczne. Dlatego też, Władku, dziękuję za twoją decyzję i deklaruję ścisłą współpracę i pomoc tu, w Warszawie, jak i rozsądne towarzyszenie na ziemi lubuskiej.

Ono zobowiązuje mnie na kolejne 4 lata w przypadku problemów czystego powietrza w Żarach, obwodnicy Krosna Odrzańskiego, innych obwodnic ziemi lubuskiej, zjazdów z A18 w gminie Wymiarki, szpitala w Ciborzu, spraw dotyczących problemów edukacji samorządów lokalnych, małej i średniej przedsiębiorczości i w ogóle indywidualnych obywateli. Mam dla was dobrą nowinę: wracam. A wy? Identyfikacja, którą wam rekomenduję na najbliższy czas, to Kurzępa - polityk z klasą.

Nie dostaliście tej szansy na powrót na Wiejską. Wiem, jak się czujecie. Wiem, jak gęste emocje was nachodzą. Dlatego też proszę i apeluję do waszych macierzystych środowisk: nie opuszczajcie ich, nie cofajcie gorliwości, wsparcia i pomocy. Czasami duma własna powoduje wycofywanie się, natomiast wielu z nich realnie potrzebuje pomocy. Apeluję więc: bądź dobry i czyń dobro. Pomóżmy koleżankom i kolegom. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. Zamykam stawkę dzisiaj. Moje oświadczenie dotyczy jakości pracy naszego parlamentu. Parę rzeczy mnie trochę irytuje, więc chciałem je dzisiaj wyrazić. Po pierwsze, cały czas słyszę tutaj, że wracamy do przeszłości, tak jakbyśmy ją tutaj budowali. Przecież my budujemy przyszłość. Ale cały czas słyszę: A wyście to zrobili, a wyście tego nie zrobili, a wyście czegoś innego jeszcze nie zrobili albo zrobiliście coś źle, dlatego my dzisiaj możemy robić to samo. Otóż jeżeli się komuś coś wytyka, to się nie robi tego samego, tylko robi się lepiej. Poza tym warto byłoby popatrzeć na to, że my wszyscy mamy jakiś udział w tworzeniu tej Polski demokratycznej. Na początku lat 90. lewica, która funkcjonowała w innym systemie, musiała dopasować prawo do państwa, do rynku, do państwa demokratycznego. To była ironia losu, ale to się stało. Wiele ustaw, dziesiątki ustaw z tamtego czasu dzisiaj jeszcze funkcjonuje, czyli dobrze to wykonała lewica. Później przyjęliśmy konstytucję, a następnie rządziła prawica, która robiła wiele reform - mówię tu o AWS-ie, zostawiła tzw. dziurę budżetową, ale nikt nie jest przecież doskonały. Później przyszła ta lewica i naprawiała to, ale to przecież wszystko robiliśmy dla naszego kraju. I potem było wejście do Unii Europejskiej. To wszytko się toczyło. Teraz jest pytanie: Czy wszyscy byli źli w tamtym czasie i trzeba im to wytykać? Oczywiście, że wiele osób i wiele instytucji popełniło błędy, ale wszyscy razem uczyliśmy się i tej demokracji, i tej gospodarki rynkowej, wzajemnych relacji, stworzyliśmy samorządy, stworzyliśmy pewien ustrój państwa, które funkcjonuje, i moim zdaniem całkiem nieźle to wygląda. Po drugie - i to zjawisko jest złe, bo ono dzieli Polaków i dzieli Polskę - drugi element to jest tworzenie prawa dzisiaj. Kiedyś 99% projektów ustaw trafiało z rządu, 1% to były ustawy poselskie, dzisiaj 95% to są projekty poselskie. Posłowie dobrze nie przygotują tych ustaw. Tylko rząd ma instrumenty, ma instytucje, które mogą to dobrze zrobić.

To wy się odnosicie do tego, że gdzieś popełniliście błąd, robiliście te ustawy na kolanach, nie przewidzieliście paru sytuacji. Wzywam wręcz do tego, żeby wrócić do dobrej tradycji, żeby projekty ustaw przygotowywał rząd, bo to jest prawidłowa droga, żebyśmy nad tym pracowali. Świat nam nie ucieknie. Mam wrażenie, że wszyscy wszystkich tu chcą ograć, koalicja rządząca opozycję, opozycja koalicję rządzącą. Mówię to po to, bo nie ma dialogu. Nasz parlament to jest arena dialogu i sporu.

Jeden dobry przykład: pani marszałek Witek usiadła z posłami Lewicy już po posiedzeniu i rozmawialiśmy. Mówię o tym, bo istota parlamentu to jest dialog, to jest poszukiwanie rozwiązań i ten spór oczywiście. Ale jak wykluczymy to z naszej działalności, z naszych relacji, jak się będziemy tu nienawidzić. Tak będzie w Polsce, przecież nie będzie inaczej. Więc chciałbym, żeby ta arena, która się nazywa Sejm, była areną sporu i dialogu, ale sporu i dialogu albo dialogu i sporu, żeby nie była teatrem, tanim teatrem ze złym spektaklem, bo przecież my oddziałujemy na ludzi, oni nas obserwują, patrzą, jaką jakość my im przekażemy, oni będą tacy sami. Jeżeli powiedzą, że ci, których wybraliśmy, nie potrafią się porozumieć, nie ma dialogu, nie umieją ze sobą rozmawiać, to jak inni będą rozmawiać? No nie będą rozmawiać i to jest smutne. Ja tu nie będę do nikogo apelował, nawoływał, bo nie ma takiego sensu, ale mówię to - do pustej sali - żeby była jakaś refleksja, bo przecież to się nagrywa gdzieś tam, bo może kiedyś taka refleksja przyjdzie i jakoś inaczej urządzimy ten nasz parlament. Dziękuję. Zapewniam, że się nagrywa.